Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Marcina Duszka, Magdalenę Łośko, Karolinę Pawliczak i Pawła Rychlika. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Magdalena Łośko i Karolina Pawliczak. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Karolina Pawliczak i Paweł Rychlik. Proszę wyznaczonych posłów sekretarzy o zajęcie miejsc. Witamy panią poseł sekretarz i zwracam się do pani z prośbą o odczytanie komunikatów. Bardzo dziękuję. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Finansów Publicznych - godz. 9, - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 9, Zdrowia - godz. 9.30, - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 10, - Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 10, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 10, - Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - godz. 10.30, - Łączności z Polakami za Granicą - godz. 11, - Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - godz. 12.15. W dniu dzisiejszym odbędzie się również posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej - godz. 14.30. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani poseł sekretarz. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Zatem przystępujemy do realizacji naszego punktu. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 7 lat temu PiS, dochodząc do władzy, szedł z hasłem walki z mafią paliwową i mafią węglową. Opowiadaliście wtedy ludziom o tym, jak będziecie walczyć ze wszystkimi przekrętami na paliwie i na węglu, jak będziecie ścigać złodziei. Dzisiaj, po 7 latach waszych rządów widzimy, że tak naprawdę szydło wyszło z worka i nie złapaliście nikogo, za to udało wam się wyhodować własny układ węglowy. Nie boję się powiedzieć - mafię węglową. To właśnie jest prawdziwa mafia węglowa, której tak szukaliście. Pod pretekstem wojennego chaosu i kryzysu na rynku energetycznym szajki spekulantów wywindowały ceny tego surowca do absurdalnych poziomów. Moje pytanie jest bardzo proste: Dlaczego pozwoliliście na powstanie mafii węglowej i na nielegalny obrót węglem w Polsce? Dlaczego, kiedy wybuchła wojna, nie zabezpieczyliście rynku surowców energetycznych przed spekulantami? Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Kretkowska. Pytanie zasadnicze: Kiedy rząd odblokuje rozwój zielonej energii z odnawialnych źródeł w Polsce, takich jak fotowoltaika, dzięki której w polskich domach mogłyby być tani prąd i tanie ciepło? Kiedy przestaniecie oszukiwać Polaków i Polki, że przyszłością Polski jest węgiel?

Pan premier, nadpremier Kaczyński ma niewątpliwie trzy sukcesy w polskiej energetyce: najpierw uśmiercił energetykę wiatrową, 6 lat temu, potem usłużni posłowie na polecenie Kaczyńskiego (Dzwonek) zmienili ustawę o fotowoltaice i uczynili ją nieopłacalną, a potem wyhodował mafię węglową, wcześniej uzależniając biedniejsze polskie rodziny, 2 mln polskich rodzin, od dostaw węgla. Skąd? Z Rosji. Z Rosji. Kiedy będą dopłaty do węgla dla tych ludzi, których dzisiaj skazaliście na ogrzewanie węglem? Kiedy odblokujecie fotowoltaikę? Kiedy zaczniecie inwestować w sieci przesyłowe, w pompy ciepła w zielony wodór? Kiedy przywrócicie korzystny dla prosumentów system rozliczania tej fotowoltaiki? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Te pytania były kierowane do prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego będzie odpowiadał pan minister Jacek Ozdoba. Bardzo proszę pana ministra. Szanowny Panie Marszałku! Jeżeli chodzi o argumenty, właściwie pytanie czy tezę, którą postawił pan poseł Iwaniak, ja się z nią nie zgodzę, dlatego że organy państwa działają, jeżeli chodzi o zwalczanie wszystkich możliwych funkcjonujących zorganizowanych grup przestępczych, a nazywanie mafią np. Unii Europejskiej - bo rozumiem, że do tego się odnosi sugestia związana z brakiem wcześniej embarga na rosyjski węgiel - jest co najmniej nie na miejscu. Trzeba pamiętać o tym, że do tej pory Unia Europejska nie nakładała na surowce embarga i jakikolwiek wyłom mógłby spowodować konsekwencje wobec Polski. Polska jako jeden z pierwszych krajów po 24 lutego wprowadziła takie embargo, co jest czymś oczywistym może nie we wszystkich krajach europejskich. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie rodzin i zabezpieczenie kontraktów, to w tej chwili mamy zabezpieczone ponad 8 mln t. To jest ta liczba, to jest ten wolumen, który był importowany z kierunku wschodniego przez prywatnych przedsiębiorców - jakkolwiek by było, wąski wycinek w ciepłownictwie. Skrócenie łańcucha dostaw oraz usprawnienie funkcjonowania wszystkich możliwych podmiotów czy też właściwie platform ma zapewnić łatwiejszy dostęp do tego surowca, a zakontraktowanie m.in. z Indonezji, Australii czy z RPA ma spowodować, że w Polsce węgla nie zabraknie. To jest wsparcie, które obejmie ponad 7 mln polskich gospodarstw. Co do kwestii dywersyfikacji dostaw gazu, bo ona również była elementem dyskusji, trzeba pamiętać o tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy od początku dywersyfikuje dostawy gazu. Przykładem może być chociażby powstanie Baltic Pipe, projekt, który był krytykowany przez PSL czy przez byłego ministra do spraw gospodarki, czy też chociażby przez środowiska lewicy.

Bardzo dziękuję panu ministrowi za udzielenie odpowiedzi. Drugie pytanie skierowane jest do ministra spraw wewnętrznych i administracji i dotyczy przedłużenia rządowych programów. Proszę bardzo, pan poseł Kopiec.

Ja rozumiem, że to jest także linia rządu, i chciałbym usłyszeć konkretną deklarację ze strony rządu, jak jest naprawdę i czy podtrzymujecie to, że tego węgla w Polsce wystarczy na 200 lat, ponieważ praktyka pokazuje, że wystarczył wam tylko miesiąc embarga na dostawy węgla z Rosji i ten system poległ.

I jaką współpracę międzyresortową i z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak UOKiK, podjęto w celu ochrony cen dla indywidualnych odbiorców? Bardzo dziękuję i przepraszam pana posła za tę nieuwagę. Ozdobę o udzielenie odpowiedzi. Lewica jak zawsze konsekwentna w traceniu przez Polskę suwerenności energetycznej. Po 24 lutego pan uważa, że Polska w energetyce powinna gwałtownie odejść od węgla, i chce pan więcej rosyjskiego gazu. To ja po prostu na tej sali mówię zdecydowanie inaczej. A co do pozostałych kwestii, to jest już punkt trzeci, który będzie w tej dyskusji, więc właściwy minister udzieli odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję. Teraz przystępujemy do zapowiadanego przeze mnie wcześniej pytania kierowanego do ministra spraw wewnętrznych i administracji, w imieniu którego będzie odpowiadał pan minister Paweł Szefernaker, dotyczącego przedłużenia rządowych programów dla pomagających uchodźcom z Ukrainy. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Monika Pawłowska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rząd w połowie marca wprowadził świadczenie 40 zł na dzień dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Potem zmieniły się przepisy, wprowadzono warunek posiadania numeru PESEL i wydłużono czas świadczenia do 120 dni lub więcej, m.in. dla osób chorych. W Polsce kończą się rządowe programy wspierające tych. W Polsce kończą się rządowe programy wspierające tych, którzy przyjęli do swoich domów osoby uciekające przed wojną z Ukrainy, ale pomaganie obywatelom Ukrainy wciąż trwa. Jak będzie wyglądało w lipcu? Pytanie: Jakie rozwiązania planuje rząd, aby rozwiązać problem przyjmowania uchodźców, aby obywatele nie musieli wybierać między sercem i pomocą a własnymi potrzebami?

Dziękuję bardzo, pani poseł. Już zmierza do mównicy pan minister Paweł Szefernaker. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

A więc nic z końcem czerwca się nie kończy, przepisy, które zostały przyjęte w marcu, w dalszym ciągu funkcjonują.

Ta pomoc, której będziemy jako Polska udzielać, ma charakter długodystansowy i dziś rozpoczynamy jej drugi etap. Wychodzimy z takiej pomocy humanitarnej związanej właśnie z pomocą dotyczącą wyżywienia dla wszystkich, noclegów dla wszystkich. W tej chwili będziemy takiej pomocy udzielać przede wszystkim tym, którzy są najbardziej potrzebujący, tzn. osobom niepełnosprawnym, kobietom, które przybyły do Polski z dużą grupą dzieci i nie mają możliwości się usamodzielnić, to będzie też pomoc dla osób starszych, czyli dla tych osób, które rzeczywiście w ciągu 4 miesięcy nie miały możliwości usamodzielnienia się w Polsce.

A więc przyjmujemy wiele różnych rozwiązań systemowych, które zostały zaakceptowane w przyjętej wczoraj przez Sejm ustawie. Ta ustawa w tej chwili jest w Senacie.

One pozostają na 120 dni dla tych osób, które przybywają do Polski. Każdy uchodźca, który przybywa do Polski, ma możliwość otrzymania od polskiej rodziny pomocy, za którą państwo polskie zapłaci. Takie działania podejmiemy w najbliższym czasie. Planujemy także w ciągu najbliższych paru dni we wszystkich województwach rozpisać konkursy dla organizacji pozarządowych, które będą zajmowały się szczególnymi przypadkami, związanymi właśnie z pomocą osobom niepełnosprawnym, z pomocą dzieciom, które potrzebują tej pomocy, a które przybyły do nas z Ukrainy. Staramy się sprawić, aby państwo polskie w swoich rozwiązaniach, procedurach zapewniło pełen wachlarz pomocy osobom, której tej pomocy realnie potrzebują. Ale chciałbym jednocześnie podkreślić, że rzeczywiście jest to taka migracja, która w skali świata, o czym mówią także eksperci, którzy się tym zajmują, chociażby z Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest szczególna, ponieważ rzadko zdarza się, aby tak duża grupa osób chciała się tak szybko usamodzielnić i podjąć pracę w miejscu, do którego dociera. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Jako drugi pytanie zada pan poseł Fryderyk Kapinos. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Uchodźcy wciąż przybywają do Polski. Są ludzie, którzy przyjeżdżają dopiero teraz, bo u nich ten szlak emigracji był bardzo długi, a często zahaczał jeszcze o zjawisko emigracji wewnętrznej. Są ludzie, którzy nie dostali jeszcze żadnej pomocy finansowej, a będą jej potrzebowali, tak samo jak dachu nad głową, edukacji czy dostępu do opieki zdrowotnej. Pytanie, jak przedstawia się sytuacja na granicy i jakie liczby dotyczące przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej odnotowuje teraz Polska. Czy przewiduje się zwiększenie czy zmniejszenie przypływu uchodźców i w jakim czasie? Dziękuję. Dziękuję. Ponownie prosimy pana ministra o udzielnie odpowiedzi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Od 10 maja na polsko-ukraińskiej granicy obserwujemy trend, w ramach którego więcej osób wyjeżdża z Polski, niż do Polski przyjeżdża.

Więc możemy mówić o paru tysiącach osób, które do Polski przyjeżdżają, właśnie uciekając z Ukrainy przed wojną, a jednocześnie więcej osób wyjeżdża na Ukrainę. W rozmowach funkcjonariuszy Straży Granicznej z tymi osobami te osoby deklarują, że chciałyby pozostać już na Ukrainie i że jeżeli tylko będzie możliwy bezpieczny powrót do ich domów, to chcą właśnie wrócić do najbliższych i móc odbudowywać swój kraj. Oczywiście dynamika wojny nie pozwala nam na jednoznaczne stwierdzenie, że taki trend będzie się utrzymywał, aczkolwiek w tej chwili na polsko-ukraińskiej granicy mamy właśnie tego typu sytuację. Codziennie z Polski na Ukrainę przejeżdża około dwudziestu paru tysięcy osób, z czego po rozmowach z tymi osobami zakładamy, że około 1/4 to są osoby, które wracają na Ukrainę, więc można założyć, że ok. 6-8 tys. osób dziennie to są osoby, które wracają na Ukrainę, uchodźcy, którzy wracają na Ukrainę z Polski. Odpowiadając na drugą część pytania, szanowni państwo, powiem, że migracja ma to do siebie, że wiele decyzji, które podejmują uchodźcy, jest bardzo dynamicznych, zmiennych.

Te osoby, myślę, traktują te wizy jako taką polisę na przyszłość, a mimo wszystko w związku z tym, że wiele osób z ich rodzin pozostaje w Europie, czy to w Polsce, czy na Ukrainie, chcą tutaj pozostać jak najdłużej. A więc współpracujemy z innymi państwami, jeżeli chodzi także o pomoc w dotarciu do tych państw osób, które chcą tam dotrzeć w celu poszukiwania bezpiecznego domu. Dziękujemy bardzo panu ministrowi.

Dotyczy ono przyczyn braku węgla i innego opału, drastycznego wzrostu ich cen oraz zysków spółek węglowych. Pierwszy pytanie zada pan poseł Marcin Kierwiński, a w drugiej kolejności pan poseł Krzysztof Gadowski. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Kilka tygodni temu pan premier Morawiecki powiedział, że Polska jest krajem bezpiecznym pod względem energetycznym. No to popatrzmy na kilka liczb, które mają opisywać to bezpieczeństwo. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla ocenia, że deficyt surowca, węgla, w tym roku przekroczy 11 mln t. Cena ekogroszku w ostatnich miesiącach wzrosła trzykrotnie, a może nawet pięciokrotnie.

Do 31% wzrósł odsetek gospodarstw znajdujących się w sytuacji ubóstwa energetycznego. I to jest to wasze bezpieczeństwo energetyczne? O tym mówi pan premier Morawiecki? Doprowadziliście do katastrofy - doprowadziliście do katastrofy na rynku energetycznym. Jesteście grupą rekonstrukcyjną PRL-u. Wprowadziliście tak naprawdę prokuratorów stanu wojennego, Dziennik Telewizyjny, zrobiliście - wy zrobiliście - skrajną inflację, a na sam koniec doprowadziliście do rzeczy, wydawałoby się, nie do pomyślenia - do tego, że nie ma węgla. To zagraża już, panie ministrze, takiemu biologicznemu bezpieczeństwu Polaków. Tu już nie ma co opowiadać tych dyrdymałów, jaką jesteście potęgą, jak wszystko jest świetnie, tylko po prostu należy reagować. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że koszt ogrzewania domku jednorodzinnego, jeżeli w ogóle będzie czym go ogrzewać, w tym sezonie grzewczym będzie wynosił między 15 a 20 tys. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? To jest to wasze bezpieczeństwo? Przecież to jest kpina. Panie ministrze, czy macie jakieś realne, podkreślam, realne rozwiązania tego problemu? Czy jedyne, co macie do zaproponowania, to program chrust+, który swoją drogą jest jakimś skrajnym wyrazem arogancji wobec Polaków? Polacy dziś nie mogą kupić węgla, nie mogą kupić ekogroszku, ceny są rekordowo wysokie, mamy do czynienia ze spekulacją na tym rynku, a wy opowiadacie, mówicie: niech sobie Polacy pójdą do lasu i chrust pozbierają. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Obecnie na rynku węgla energetycznego panuje bardzo trudna sytuacja cenowa i podażowa w efekcie wydarzeń z ostatnich miesięcy. Nastąpiła istotna zmiana sytuacji geopolitycznej, wojna w Ukrainie zaburzyła dotychczasowy ład. Dodam od siebie tylko tyle, że nic, co było jeszcze 24 lutego, już się nie powtórzy, świat będzie inny i jest inny. Wojna zaburzyła dotychczasowy ład, a w konsekwencji pozrywane zostały istniejące łańcuchy dostaw, co wywołało kryzys energetyczny i przełożyło się na ograniczenie importu surowców energetycznych na terytorium Unii Europejskiej i wzrost ich cen. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że z uwagi na zachodzące w Unii Europejskiej procesy transformacji energetycznej wynikającej z celów redukcji emisji

Importem węgla kamiennego zajmowały się głównie podmioty prywatne. Węgiel importowany z Rosji w zdecydowanej większości trafiał do odbiorców indywidualnych, jak również do małych ciepłowni, przedsiębiorstw i ogrodników. Chciałbym tu przypomnieć jedną rzecz: importowano węgiel rosyjski, bo węgiel rosyjski był najtańszy na rynku, a prywatni przedsiębiorcy pracują na własny zysk. Problem niedoborów węgla nie dotyczy dużej energetyki, która jest największym konsumentem tego paliwa oraz największym odbiorcą węgla z polskich kopalń. Energetyka ma zabezpieczone dostawy węgla dzięki temu, że już w poprzednich latach ograniczała wykorzystywanie węgla importowanego na rzecz węgla z polskich kopalń. W najtrudniejszej sytuacji aktualnie są podmioty, które dotychczas korzystały z węgla importowanego, oraz odbiorcy indywidualni zaopatrujący się przez pośredników. Spółki Skarbu Państwa potwierdzają zwiększenie produkcji w bieżącym roku, a pierwsze wyniki wdrożonych działań i zaangażowania górników są już widoczne. Na przykład w marcu bieżącego roku wydobyto o 176 tys. t węgla energetycznego więcej niż w marcu 2021 r., a w kwietniu o 151 tys. t więcej niż rok wcześniej.

Mówię oczywiście o węglu energetycznym. Trzeba jednak podkreślić, że przygotowanie nowych ścian jest procesem czasochłonnym i kosztownym.

Kolejna kwestia.

W efekcie oferta przygotowana przez PGG SA jest atrakcyjna i wzbudza ogromne zainteresowanie wśród klientów, którzy chcą pozyskać ten rodzaj paliwa opałowego. Jednakże zainteresowanie przekracza obecnie możliwości spółki w zakresie podaży surowca, co przekłada się na powstawanie utrudnień i brak możliwości jednoczesnego obsłużenia wszystkich zainteresowanych. Ponadto należy jeszcze raz podkreślić, że węgiel opałowy jest pochodną całości produkcji węgla z kopalń i nie można go w prosty sposób przekierować z innego kierunku do sektora komunalno-bytowego, by w ten sposób zwiększyć dostępność tego paliwa. Podkreślenia wymaga również fakt, że obecna trudna sytuacja nie dotyczy jedynie Polski.

W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy składów węglowych. Są to podmioty prywatne, które działają w celu osiągnięcia zysku. Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także spółki produkujące węgiel nie mogły kształtować cen, po jakich oferowany jest węgiel przez pośredników prowadzących składy węglowe. Przy notowanym obecnie ogromnym popycie naturalną konsekwencją był wzrost cen. Kolejne pytanie zada pan poseł Krzysztof Gadowski. Wysoka Izbo! Rząd nie panuje nad wydobyciem, nie panuje nad sprzedażą węgla, nie panuje nad importem, ba, nie panuje nawet nad chrustem. Polacy, panie ministrze, widzą, że ten chaos, bałagan, ta wasza niekompetencja doprowadziła do czego? Doprowadziła do tego, co mamy dzisiaj, czyli szalejącej drożyzny, 300-procentowego wzrostu cen węgla. Przedsiębiorstwa pod kontrolą Skarbu Państwa generują wysokie marże i generują najwyższe zyski. Polacy generują największe koszty. Panie Ministrze! Opamiętajcie się. Polacy chcą prostej odpowiedzi. Chcą wiedzieć, jaką macie strategię, za ile mogą kupić węgiel, ile będzie kosztowała 1 t węgla importowanego, kto będzie mógł kupić, kiedy, ile będzie kosztowała wiązka chrustu (Dzwonek) na Orlenie. Proszę pana ministra Pyzika ponownie o udzielenie odpowiedzi.

Bardzo dziękuję za to pytanie uzupełniające. Jeśli chodzi o kwestię najistotniejszą, czyli obrony rynku, a dokładnie konsumentów przed tymi cenami, to pracuje nad tym zespół powołany przez panią minister Annę Moskwę. To jest kwestia synchronizacji importu węgla, realnych możliwości wydobywczych. Właśnie o nich przed chwilą Wysoką Izbę poinformowałem. Przeczytam dalej. Wyniki finansowe spółek górniczych: wydobycie węgla kamiennego ogółem, co obejmuje węgiel energetyczny i koksowy, po 4 miesiącach bieżącego roku wynosiło 19 mln t i w porównaniu do 4 miesięcy było wyższe o 153 400 t.

Natomiast cena sortymentów średnich, drobnych węgla energetycznego, czyli m.in. ekogroszku, wzrosła o 68%, a cena sortymentów grubych rok do roku, jeśli chodzi o pierwsze 4 miesiące, wzrosła o 33%. Celowo nie podaję wartości, ponieważ ceny te obejmują sprzedaż zarówno do dużych odbiorców, do odbiorców indywidualnych, jak i do pośredników. Chciałem zobrazować skalę podwyżek w kopalniach i jak to przekłada się na zysk kopalń.

Zauważyć jednak należy, że wyniki obejmują także segment węgla koksowego, który w ostatnich miesiącach także osiąga swoje rekordy. Jeżeli któryś z panów posłów czuje się nieusatysfakcjonowany odpowiedzią, bardzo proszę złożyć zapytanie, a będzie odpowiedź na piśmie. Pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego odpowiadał będzie członek Rady Ministrów pan minister Łukasz Schreiber. Pytanie dotyczy wątpliwości dotyczących prawidłowości oświadczenia majątkowego prezesa Rady Ministrów. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Dariusz Joński, a jako drugi - pan poseł Michał Szczerba. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie szedł do polityki dla żadnej idei. Kłamał, mówiąc takie słowa. Szedł do polityki, aby spekulować na majątku państwowym. Mało mu było, że spekulował na działkach kościelnych, które razem z żoną kupił za 700 tys. zł, a sprzedał za 15 mln zł. Roku temu, kiedy posiadał informacje, których nie przekazał opinii publicznej, cały swój zgromadzony majątek finansowy przerzucił z banków i zakupił obligacje. A więc nie zależy mu na tym, żeby tę inflację zbijać, bo straci. A jak znamy Morawieckiego i jego chciwość, to możemy sobie wyobrazić, że pociągnie nas na dno, żeby zarobić.

Być może gdyby ludzie o tym wiedzieli, stać ich by było dzisiaj na to, by kupić węgiel, a nie palić chrustem w piecu. Dziękuję bardzo panu posłowi.

Proszę bardzo, panie pośle. Właśnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że dwuletnie obligacje o oprocentowaniu stałym nie będą już dostępne.

Pan reprezentuje premiera Morawieckiego, który powinien być w tym miejscu. Na jakich zasadach i kiedy pan premier Morawiecki, nadzorujący ministra finansów, który sprzedawał te obligacje w imieniu ministra Skarbu Państwa. A kto sprzedawał te obligacje? Biuro maklerskie banku państwowego. Na jakich zasadach kupił on te obligacje? Po drugie: Kiedy będzie projekt legislacyjny dotyczący jawności oświadczeń majątkowych rodzin polityków? Zatrzymaliście to rękami Julii Przyłębskiej i do tematu nie wracacie.

Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo pana ministra Łukasza Schreibera.

Wysoka Izbo!

Po pierwsze, to nie jest chyba dla nikogo sensacją, że pan premier posiada majątek, który co roku deklaruje opinii publicznej w oświadczeniu majątkowym. też może warto przypomnieć niektórym na tej sali, jest jawne dzięki działalności posłów III kadencji Sejmu. Jednym z inicjatorów takiego rozwiązania był pan prezes Jarosław Kaczyński, inicjatorami byli także inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, tak jak mówiłem, majątek premiera jest od wielu lat deklarowany w oświadczeniach majątkowych - to sprawa zupełnie jasna.

Idźmy teraz dalej: obligacje skarbowe, obligacje Skarbu Państwa. Państwo uważacie, że to jest coś wstydliwego? Wolelibyście, rozumiem, żeby polski premier inwestował w jakieś fundusze inwestycyjne zagraniczne albo lokował za granicą swoje środki? Myślę, że wręcz przeciwnie.

To chcecie państwo powiedzieć? Zachęcam do minimum przyzwoitości w tych wypowiedziach. Uważam, że nie.

Spójrzcie na Włochy czy na Japonię.

Zresztą to nie jest żadna tajemnica i to, co panowie opowiadacie, jakby to była jakaś tajna operacja czy też operacja dostępna tylko dla, nie wiem, posłów albo członków Rady Ministrów. Nie, dla każdego obywatela.

A więc jest to sprawa absolutnie transparentna.

Państwo macie powód do wstydu za to, w jaki sposób zadaliście te pytania. Dziękuję bardzo. Kolejnym pytaniem także panowie posłowie się podzielą. Tym razem jako pierwszy pan poseł Michał Szczerba. Szanowny Panie Marszałku! To jest kluczowe pytanie, które chcielibyśmy zadać: Czy pan premier Morawiecki ma naturę premiera, czy nadal ma naturę bankstera? Szanowni Państwo! Insider trading jest to wykorzystywanie poufnych informacji, które posiadał rząd, do tego, żeby pomnażać swoje zyski. I na to pan nie odpowiedział, na ten konflikt interesów, który w tej sprawie jest absolutnie oczywisty. Teraz chcielibyśmy powiedzieć o tym, że żyjemy w biedniejącym społeczeństwie. I premier, który ma dostęp do informacji, że będzie inflacja, indeksowane obligacje, indeksowane inflacją, kupuje. Dziękuję bardzo. Pozostało 6 sekund, panie pośle. Być może zostało 6 sekund, ale dla wielu ludzi to jest naprawdę poważny problem, dlatego że tracą swoje oszczędności. Problem polega na (Dzwonek) tym, że Glapiński mówił w zeszłym roku o deflacji. Premier Morawiecki i Glapiński mają pełną informację na temat finansów państwa. I Morawiecki wykorzystał to, wzbogacając się, a nie informując ludzi. Prowadziliście w zeszłym roku różne kampanie billboardowe, informacyjne, łącznie z tym, że wysyłaliście billboardy za granicę, a nie potrafiliście przekazać ludziom informacji, żeby inwestowali m.in. w obligacje, bo nie stracą swoich oszczędności. Pan minister Łukasz Schreiber.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wydaje mi się, że już na wszystkie te pytania odpowiedziałem.

Wiem, że mierzycie ludzi swoją miarą i swoich być może kolegów, swoich ministrów, ale skończcie z tym. Chcecie, tak się domagacie teraz jawności. Niech lider opozycji pokazuje swoje oświadczenia majątkowe. Dlaczego tego nie robi?

Myślę, że to będzie z większym pożytkiem dla opinii publicznej niż takie filipiki jak te przed chwilą, w których tak naprawdę bezpodstawnie obrażacie ludzi. Korzystacie z immunitetu, bo wiecie, że za słowa wypowiedziane tutaj trudno kogoś postawić przed sądem. Jeszcze raz, bardzo proszę, panie pośle.

A odnośnie do obligacji to jeszcze raz powiedzmy to sobie. Państwo mówcie, my będziemy mówili: tak, niech Polacy kupują obligacje, niech inwestują w obligacje Skarbu Państwa. Będzie to z korzyścią i dla obywateli, i dla Polski, i dla zmiany struktury długu publicznego.

Gdybyście mogli powiedzieć, że premier zdobył nielegalnie majątek, gdybyście mogli wskazać takie wątpliwości.

To jest droga, którą kroczycie od 7 lat, droga, którą kroczycie do kolejnej klęski. Teraz pytania będą zadawali, w następującej kolejności, panowie posłowie Ireneusz Raś i Radosław Lubczyk. Sprawa dotyczy komponentu kolejowego CPK. Pytanie skierowane jest do prezesa Rady Ministrów, w którego imieniu głos zabierze obecny już wśród nas pan minister Marcin Horała. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Ministrze! Wysoki Sejmie!

Nasze pytanie w tej chwili, panie ministrze, dotyczy tej sprawy.

Od tego odchodzicie tzw. dziesięcioma szprychami.

Chodzi o pieniądze na inżynierów, na konsultantów.

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana ministra Marcina Horałę.

Panie Marszałku! W jakim stopniu odbiegają do rzeczywistości? Wystarczy nawiązać do tego, o czym pan poseł wspominał, czyli do takiej akcji posłów PSL-u w całej Polsce, zatroskanych o to, że przejęcie.

Natomiast w przypadku przytłaczającej większości lotnisk w Polsce PPL ma taki wpływ jak udziałowiec mniejszościowy, tzn. choćby chciało coś zrobić, udziałowcy większościowi mogą zdecydować inaczej.

Urbanizacja w Polsce postępuje, nowe tereny obejmowane są różnymi kategoriami ochrony środowiska i nie można w prosty sposób powielać rozwiązań sprzed 10 lat, bo one powstały w innych uwarunkowaniach. Ja też ubolewam nad tym, że rząd PO-PSL ten projekt zarzucił, ale skoro już go zarzucił, to nie ma do niego powrotu, trzeba wszystkie analizy i modele zrobić od nowa, w tych realiach, jakie są obecnie. Bardzo dużym nadużyciem jest mówienie, że projekt CPK narusza policentryczny model rozwoju kraju. Jest dokładnie odwrotnie, tzn. jeżeli małe miejscowości są pozbawione komunikacji kolejowej lub tę komunikację mają bardzo słabą, są pozbawione dużej liczby połączeń, to dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą, dla młodych ludzi, którzy chcą planować swoje życie, właściwie pozostaje jedna opcja: wyprowadzić się stamtąd, przenieść się do dużej metropolii. To był model preferowany przez rządy PO-PSL. Natomiast w ramach inwestycji kolejowych CPK, czyli budowy 2000 km nowych linii kolejowych i modernizacji kilku tysięcy kolejnych kilometrów linii kolejowych dokonywanej przez spółkę PKP PLK, o czym też za chwilę, cały szereg miast w Polsce, cały szereg mniejszych miejscowości uzyska dostęp do systemu transportowego kraju. Miejscowości takie jak Sieradz, jak Płock, jak Włocławek, jak Ostrołęka, jak Łomża, jak Jastrzębie-Zdrój uzyskają cały szereg nowych, szybkich połączeń.

W tym programie praktycznie nie ma budowy nowych linii kolejowych, a potrzebujemy budowy nowych linii kolejowych, i to w standardzie KDP.

Więc mówienie o jakichś ośrodkach kompetencji, które zostały wtedy utworzone do budowy linii kolejowych, to jest nieprawda. Były kompetencje najwyżej do zamykania linii. Jeżeli musimy stworzyć nowe centrum eksperckie, nowe centrum kompetencji - bo KDP w Polsce nie mamy - to można to było utworzyć również w nowym podmiocie, który dzięki temu będzie skoncentrowany, jako typowa konstrukcja typu SPV, właśnie na budowie tych linii, i tak się stało. We współpracy chociażby z Instytutem Kolejnictwa CPK opracowało standardy kolei dużych prędkości w Polsce. Pytanie o analizy.

To wszystko funkcjonowało raczej w logice wydawania środków, żeby wydać 100% środków z Unii. Więc zaczynamy bardzo dużo inwestycji - połowa się opóźni, w połowie coś nie wyjdzie, ale na koniec przyjdzie nowa perspektywa, to będzie ich wystarczająco dużo, w miarę zaawansowanych, żeby je zrealizować i wydać środki unijne, natomiast zupełnie bez tej analizy systemowej, którą wprowadziło właśnie CPK.

Te analizy pokazują, że dzięki realizacji programu inwestycyjnego CPK ruch wzrośnie, przykładowo, na stacji Lublin o 200%, w Jeleniej Górze - o 170%, w Nowym Sączu - o 142%, w Sieradzu - o 135%, w Skierniewicach - o 114%, w Gorzowie Wielkopolskim - o 108%, a w Zawierciu - o 99%. Mówimy o stacjach istniejących, bo jak zmierzyć wzrost ruchu pasażerskiego na stacji pasażerskiej Łomża, której obecnie w ogóle nie ma? 60-tysięczne miasto, odcięte zupełnie od komunikacji kolejowej, dzięki realizacji programu CPK taką komunikację zyska.

Ewentualnie inwestycje PKP PLK mogłyby stać w sprzeczności z inwestycjami CPK, bo to CPK odpowiada za główny kręgosłup transportowy, za podstawowe linie, do których linie niższego rzędu muszą się dołączyć, ale oczywiście tak nie jest.

Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Panie Ministrze! Doskonale zdaje sobie pan sprawę, że dzisiaj każdy, kto robi jakąkolwiek inwestycję w firmach, wie, że jest coś takiego jak cena dnia.

Kolejne pytanie o to, co mnie bardzo interesuje: Jak wygląda stan konsultacji społecznych w sprawie wariantów linii kolejowych w poszczególnych województwach i jakie zarzuty najczęściej się pojawiają?

Pan minister mówi o tym, że będzie to połączenie z innymi miastami. Mówicie o szybkiej kolei, która ma osiągnąć prędkość 250 km. Rozumiem, że będzie zatrzymywała się na tych stacjach, gdzie posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą wsiadali do tych pociągów. Bardzo dziękuję panu posłowi. Widzę, że państwo się niczego nie nauczyliście na przykładzie stacji Włoszczowa, która też przez ówczesną opozycję była tak wyśmiewana, że tam pociągi się będą zatrzymywały. A zwłaszcza lokalna społeczność ma możliwość rozwoju, ma możliwość dojazdu w swoich życiowych sprawach.

Źródła finansowania są oczywiste, takie jak przy każdej infrastrukturze publicznej w Polsce, czyli budżetowe środki polskie i środki unijne.

Generalnie w systemie polskich inwestycji infrastrukturalnych obok dwóch dotychczasowych dużych programów, czyli programu budowy dróg krajowych i autostrad i ˝Krajowego programu kolejowego˝, program CPK będzie trzecim dużym programem infrastrukturalnym, jeżeli chodzi o wielkość nakładów, porównywalnym z tymi dwoma wcześniej wspomnianymi. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, jesteśmy w tej chwili w trakcie prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym na całym szeregu odcinków. Na jednym już się zakończyły, na odcinku Warszawa - Łódź trwały rok, to też bardzo sprawne tempo.

W ramach projektu odbyły się dwie tury konsultacji społecznych z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, konsultacje branżowe i spotkania z jednostkami samorządu terytorialnego. W pierwszym etapie konsultowano cztery rozwiązania wariantowe, zebrano ankiety, odbyły się spotkania. W toku uwag i przy uwzględnieniu tych uwag przygotowano trzy nowe przebiegi hybrydowe, składające się z najlepiej ocenionych fragmentów z tamtych poprzednich czterech. Dla nich przeprowadzono uproszczoną analizę wielokryterialną. Warianty te następnie były przeznaczone do ponownej tury konsultacji społecznych.

Po ich wykonaniu będzie trzecia tura konsultacji społecznych, na podstawie których zostanie wyłoniony wariant inwestorski (Dzwonek), co dla tego odcinka jest planowane w III kwartale 2022 r. To była ich wola, pewnie nie wszyscy się wpisali. W 32 gminach, czyli we wszystkich objętych oddziaływaniem inwestycji, w tej turze zebrano również 21 809 ankiet drogą elektroniczną. Tam wszystkie zgłaszane wnioski i rozwiązania są rozważane. Wszyscy chcemy mieć dobre połączenia kolejowe, dobre drogi, miejsca pracy, fabryki, ale mówimy: nie u mnie, tylko we wsi obok, w gminie obok, w dzielnicy obok, tak żebym miał tam blisko, żebym mógł łatwo dojechać, ale żebym nie był bezpośrednim sąsiadem lub nie był wywłaszczany. Wreszcie ostatnia kwestia. To jest też przykład, dlaczego muszą się tym zajmować eksperci.

Natomiast grono lokalnych samorządowców, chcąc właśnie wypchnąć przebieg poza teren ich gmin, niestety wymyśliło sobie taki przebieg, który niszczy tereny chronione. Takich przebiegów niestety nawet nie warto w pogłębionym stopniu analizować, bo one są prawnie zabronione. Wszelkie przepisy ochrony środowiska również jak najbardziej w tym procesie trzeba honorować. Proces przygotowania inwestycji jest bardzo ściśle sparametryzowany przez polskie prawo. Ono jest zakotwiczone w Unii Europejskiej, w prawie unijnym. Są kolejne etapy rozmów, kolejne etapy konsultacji.

Wszystkie konsultacje do tej pory wykonane przez CPK są nadmiarowe i dodatkowe, ponieważ jest to najbardziej transparentny i najbardziej konsultowany w historii polski program inwestycyjny. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Przechodzimy do kolejnego pytania. Będzie ono skierowane do ministra spraw zagranicznych, w imieniu którego udzielać odpowiedzi będzie pan minister Szymon Szynkowski vel Sęk. Dotyczy ono celów dalszego zacieśnienia współpracy w ramach Trilogu. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Barbara Dziuk. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polityka międzynarodowa to jest priorytet każdego państwa, każdego kraju na całym świecie, również Polski. Zauważamy potencjał dalszego zacieśniania współpracy w ramach Trilogu oraz perspektywy rozszerzania tej formuły. Wskazuje to, że format ten udowodnił swoją użyteczność w ciągu 10 lat funkcjonowania tych spotkań. Potencjałem jest niewątpliwie współpraca polityczna, wojskowa tych trzech państw. To są trzy kraje. To one są filarami wschodniej flanki NATO znajdującej się na pierwszej linii Sojuszu i doświadczają bezpośrednich zagrożeń dla swojego bezpieczeństwa ze strony agresywnej polityki Rosji. Celem jest zacieśnienie współpracy między sojusznikami reprezentującymi największe państwa wschodniej flanki NATO oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego. Szefowie dyplomacji trzech krajów wiele uwagi poświęcili sytuacji bezpieczeństwa w regionach. Z zadowoleniem przyjmujemy, że wspólnie poszukujemy możliwości skutecznego reagowania na trudną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie wobec agresji Rosji na Ukrainę i jej implikacji dla Gruzji i Mołdawii. Ministrowie odnieśli się tutaj również do procesu adaptacji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach przygotowań do szczytu NATO w Madrycie. Moje pytanie, panie ministrze, jest takie: Jaki jest cel dalszego zacieśniania współpracy tych państw?

Bardzo dziękuję, pani poseł, za zadanie pytania. O udzielenie odpowiedzi proszę wspomnianego wcześniej pana ministra.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Posłowie! Pani Poseł! Dziękuję bardzo za podjęcie w tym pytaniu tematu współpracy w ramach Trilogu, rzeczywiście bardzo ważnego formatu współpracy, który obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie, zainicjowanego przez Rumunię, natomiast dzisiaj odgrywającego ważną rolę w polskiej polityce zagranicznej, bo stanowiącego doskonałe uzupełnienie innego formatu - bukareszteńskiej dziewiątki, który jest formatem stricte zorientowanym na wzmacnianie bezpieczeństwa naszych krajów, krajów wschodniej flanki NATO w regionie. O ile do formatu bukareszteńskiej dziewiątki należy Rumunia, o tyle nie należy do tego formatu Turcja.

Dwa z tych krajów należą do Unii Europejskiej.

Propozycją turecką jest to, aby takie spotkanie, którego gospodarzem będzie Turcja, mogło się odbyć jeszcze w tym roku.

A więc siłą rzeczy adresatem tego formatu i punktem ciężkości są takie kraje jak dzisiaj Ukraina, ale też Gruzja, jeszcze przed agresją. Ministrowie spraw zagranicznych tego kraju są zapraszani na spotkania tego formatu. Turcja wychodzi również z propozycją, która jest realizowana, aby intensyfikować współpracę przedstawicielstw dyplomatycznych tych trzech krajów przy różnych organizacjach międzynarodowych, przy NATO, przy OBWE. Również ten format i współpraca obejmują wzajemne zwiększenie obecności personelu wojskowego w strukturach NATO ulokowanych na terytorium tychże trzech krajów. Istotnie, tak jak pani poseł już wspomniała, najważniejszą kwestią na agendzie oczywiście był rozwój wydarzeń w kontekście kryzysu na Ukrainie, ale także dyskutowano na temat koncepcji strategicznych w procesie przygotowań do szczytu w Madrycie oraz przyszłości trójstronnej współpracy w ramach Trilogu. Ministrowie oczywiście bardzo jasno odnieśli się do kwestii rosyjskiej agresji, potępiając ją, ale także ocenili możliwość wsparcia militarnego, ekonomicznego i politycznego dla Ukrainy. Omówili kwestię rosyjskiej blokady ukraińskiego eksportu zbóż, olejów i nawozów sztucznych zagrażającej bezpieczeństwu żywnościowemu świata. Zgodzili się także co do tego, że Rosja musi ponieść odpowiedzialność za popełnione zbrodnie. Omówili równocześnie kwestie wzmocnienia jedności Sojuszu przy okazji przygotowań do najbliższego szczytu NATO, nadania priorytetu obronie kolektywnej jako najważniejszemu zadaniu oraz wzmocnienia postawy obrony i odstraszania, zwłaszcza na flance wschodniej, w duchu ścisłej współpracy transatlantyckiej i zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie.

Jak już wspomniałem, strona turecka zadeklarowała gotowość goszczenia pierwszego szczytu Trilogu na szczeblu głów państw w drugiej połowie bieżącego roku, ale jest też przedstawiana, proponowana wizja rozwinięcia współpracy międzyparlamentarnej w formie spotkań na szczeblu przewodniczących parlamentów lub komisji spraw zagranicznych. Takie propozycje pojawiły się już jesienią ubiegłego roku. Dodanie tego formatu parlamentarnego stanowiłoby naturalną konsekwencję i uzupełnienie formuły Trilogu. Jestem zawsze entuzjastą wzmacniania otoczenia polskiej dyplomacji także poprzez aktywność parlamentarną, więc oczywiście liczymy bardzo na to, że ten format parlamentarny również się pojawi. Także w kontekście parlamentarnym sednem współpracy Trilogu pozostałaby problematyka bezpieczeństwa tak w wymiarze NATO, jak i regionalnym, działania na rzecz wzmacniania flanki wschodniej. I tutaj pierwsze wstępne propozycje mówią o możliwym spotkaniu w tym formacie w 2023 r., ale być może będzie przestrzeń do tego, żeby zrobić to jeszcze w tym roku wobec dynamiki sytuacji i ze względu na potrzeby. Podsumowując, panie marszałku, szanowni państwo posłowie, chciałem powiedzieć, że 10-lecie tego formatu pokazuje jego użyteczność i znaczący potencjał rozwoju. Minister Rau podczas majowego spotkania zaprosił już swoich rumuńskich i tureckich odpowiedników do złożenia wspólnej wizyty w Warszawie. A więc najbliższe spotkanie ministrów spraw zagranicznych, bo to jest dzisiaj esencja funkcjonowania tego formatu, odbędzie się w Warszawie w przyszłym roku. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Przechodzimy do kolejnego pytania, które. Pan poseł Jach. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Poprosimy pana ministra. Dziękuję, panie marszałku. Szanowny Panie Przewodniczący!

Niemniej jednak dialog służy właśnie temu, żeby lepiej poznać zastrzeżenia Turcji, żeby starać się też wykonać pracę w zakresie tego, żeby te zastrzeżenia zostały jak najszybciej uchylone, żeby ewentualne wątpliwości zostały rozwiane. Nad tym intensywnie pracujemy w dialogu z naszymi tureckimi partnerami, nie tylko w formacie trilogu, ale również w bezpośrednich kontaktach na różnych szczeblach. Podejmujemy dialog na różnych poziomach, wskazując naszym tureckim partnerom na to, że jest w interesie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale w szczególności w tej chwili w interesie mogących czuć się zagrożonymi krajów północno-wschodniej, tak to bym określił, flanki, czyli krajów bałtyckich i Polski, żeby uzupełnić skład sojuszu o dwóch nowych członków, i że to wzmocni potencjał odstraszania i zwiększy bezpieczeństwo w regionie. Liczymy więc także na wsparcie Turcji. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie i miesiące pozwolą nam dojść do punktu, w którym te zastrzeżenia i wątpliwości Turcji zostaną rozwiane. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Przystępujemy do kolejnej tury pytań. Zadawać je będą panowie posłowie Cezary Tomczyk oraz Marek Rząsa. Skierowane one są do prezesa Rady Ministrów, dotyczą cen paliw oraz zysków i wysokich marż koncernów paliwowych, a odpowiedzi na zadane pytania udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pan minister Jan Kanthak. A teraz prosimy pana posła Cezarego Tomczyka. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedyś chyba poseł Marek Suski powiedział, że to nieprawda, że w całej Polsce drożeje benzyna, bo drożeje tylko na stacjach benzynowych. To jest idealny przykład, który pokazuje, jak jesteście dzisiaj oderwani od rzeczywistości, jak jesteście oderwani od tego, czym żyją Polacy, bo oderwaliście się już jakiś czas temu. Te koncerny paliwowe i energetyczne mają dzisiaj rekordowe zyski, więc dzisiaj chciałbym panu ministrowi zadać pytanie: To na kim oni mają te zyski? Na Szwedach mają te zyski polskie koncerny paliwowe, na Norwegach mają te zyski czy może mają jednak na Polakach? Bo wy dzisiaj próbujecie wyciągnąć każdą złotówkę z kieszeni Polek i Polaków tylko po to, żeby łatać wasz dziurawy budżet. I każdy to wie, bo każdy dzisiaj może stanąć na stacji benzynowej Lotosu i Orlenu i zobaczyć, jak wyglądają ceny. I teraz uwaga: Dlaczego te ceny tak wyglądają? Szanowni państwo, to jest tablica, która pokazuje - myślę, że na wykresie wszyscy zobaczymy to dość łatwo - jak wzrosły marże Lotosu i Orlenu w ciągu ostatnich 4 miesięcy. A więc marża Lotosu wzrosła o 3300%. Trzydziestotrzykrotność tego, co było w styczniu. To jest dzisiaj łupienie każdego kierowcy, który jeździ polskimi drogami. Marże Orlenu - wzrost o 1000%. To jest dzisiaj łupienie każdego kierowcy, który jeździ polskimi drogami. W dodatku zobowiązaliście się w Krajowym Planie Odbudowy do tego, żeby wprowadzić nowy podatek, podatek od aut spalinowych. Czy ktoś na tej sali po prawej stronie w tych ławach rządowych w jakikolwiek sposób jeszcze myśli? Bo wydaje mi się, że nie. Każdy Polak dzisiaj płaci ogromną cenę za waszą nieudolność. Każdy Polak dzisiaj mierzy się z inflacją, z drożyzną, z wysokimi podatkami, które podnieśliście ponadczterdziestokrotnie. I mówię dzisiaj w imieniu kierowców, ale też wszystkich tych, którzy nie mogą wam tego powiedzieć, jak naczelniczka poczty z Pacanowa, bo ją chcecie wyrzucić z pracy, że to musi się skończyć, że drożyzna i inflacja to jest coś, co wy spowodowaliście razem z panem Glapińskim i Narodowym Bankiem Polskim, a Polacy was z tej inflacji i drożyzny rozliczą. Zamiast aut, które palą wiele litrów benzyny, tych limuzyn, do których wsiedliście i zapomnieliście o bożym świecie, pojawi się inny środek transportu, który nazywa się taczka, a wiecie, co politycy robią na taczkach. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana ministra Jana Kanthaka o udzielenie odpowiedzi. Wysoka Izbo! Udany happening, koledzy nagrali, będzie pan miał okazję wrzucić to do mediów społecznościowych, pochwalić się, że jest pan pracowitym posłem. Panie Pośle!

A pana ministra proszę, aby nie oceniał wystąpień posłów, tylko odniósł się do zadanych pytań.

W sposób oczywisty - każdy ma tego świadomość - wynika to z sytuacji geopolitycznej i z tego, że Putin wywołał wojnę, wypowiedział wojnę Ukrainie. O tym najlepiej świadczą, szanowni państwo, liczby. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Rosja odpowiadała za 11 mln baryłek ropy naftowej dziennie, a teraz Polska, Niemcy i cała UE decydują się, aby z tej ropy nie korzystać, to w sposób naturalny i oczywisty ceny rosną. To jest cena naszego bezpieczeństwa i naprawdę czasami klasa polityczna powinna być odpowiedzialna i powinna jak jeden mąż stanąć w prawdzie i powiedzieć: wiemy, że ceny są wysokie. wiemy, że te koszty niestety ponoszą obywatele, ale prawda jest taka, że ta cena ma swoją wartość, wartość bezpieczeństwa i niezależności od Rosji. Chciałbym serdecznie zaprosić, bo jeśli to nie wynika ze złej woli pana posła Tomczyka i posłów Platformy Obywatelskiej, ale po prostu z niewiedzy, to już teraz, jeszcze przed głosowaniami zapraszam na takie godzinne korepetycje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, na których wytłumaczymy. na czym polega modelowa marża rafineryjna. Dlatego dziękuję za możliwość wystąpienia dzisiaj i opowiedzenia o modelowej marży rafineryjnej, która jest takim benchmarkiem, jest algorytmem, który funkcjonuje od wielu, wielu lat i nie został w żaden sposób zmieniony. Z czego to wynika, szanowni państwo?

Ural w porównaniu do ceny baryłki ropy Brent, która jest teraz zakupywana w związku właśnie z działaniami Putina. To pierwszy czynnik. Drugi czynnik to kwestia wartości dolara do złotówki.

Naprawdę nie bądźmy obłudni, spójrzmy, jakie są ceny w Unii Europejskiej. W Polsce jest najtańszy olej napędowy w całej Unii Europejskiej, a jeśli chodzi o benzynę, to jesteśmy, zdaje się, drugim czy trzecim państwem Unii Europejskiej, w którym są najniższe ceny benzyny. Mówimy o rządzie. Jakie rząd ma narzędzia do tego, aby kształtować ceny paliw? Takie, których Donald Tusk nie znał. Mówił: jak ktoś mi pokaże przyciski, które należy naciskać, to ja będę je naciskał. My znaleźliśmy przyciski. Pan poseł Rutnicki, widzę, jest bardzo taki. Panie pośle, trochę spokoju, naprawdę.

A przypomnijmy, jakie były wtedy zarobki. Sytuacja, szanowni państwo, oczywiście nie jest łatwa i nie jest dobra z punktu widzenia obywateli, ale gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdybyście wy rządzili, to ceny już nie mieściłyby się na pylonach na stacjach benzynowych, bo byłoby to powyżej 10 zł. Bardzo dziękuję. I teraz mamy kolejną osobę, która będzie zadawała pytanie. Jest nią pan poseł Marek Rząsa. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

zabijanie kredytobiorców, podnoszenie stóp procentowych, niebotyczne ceny paliw, podnoszone w zasadzie każdego dnia - oto w największym skrócie obraz dzisiejszej Polski rządzonej przez PiS. W zasadzie to nie są rządy, to jest nierząd. Ale Polacy to widzą i doskonale wiedzą, że po prostu łupicie ich bezczelnie, ich portfele. Kiedy byliście w opozycji, mieliście rozwiązania na wszystko. Wszyscy pamiętają słowa pani Szydło, pana Kaczyńskiego, pana Błaszczaka, gdy stali na stacjach benzynowych i mówili, co można zrobić, żeby obniżyć cenę paliwa, które nie kosztowało nawet 5 zł.

Pytanie było proste: Dlaczego są takie duże marże? Bardzo prosimy pana ministra.

Proszę bardzo, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy naprawdę - już o tym wspomniałem - festiwal hipokryzji. Teraz okazuje się, że za inflację na świecie też pewnie odpowiada prezes Glapiński i prezes Jarosław Kaczyński. Jak pan poseł Rząsa pytał o ceny, to ja mogę też zapytać: Jak to jest, że skoro w Polsce są takie wysokie ceny, to mieszkańcy Niemiec, Czech i innych państw sąsiadujących z Polską przyjeżdżają do Polski, żeby zatankować u nas paliwo? Szanowni panowie posłowie, może to ostudzi emocje, jeśli powiem, że naszym obradom przysłuchuje się młodzież z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Gliwic, która przyjechała na zaproszenie pana posła Jarosława Gonciarza. Z pewnością należy ją bardzo serdecznie powitać. A zatem proszę o ostudzenie emocji.

Ale rozumie pan, czym się różni coś modelowego od realnego, i że jeśli uwzględniona jest cena baryłki, tak jak wspomniałem, Ural pochodzącego z Rosji, a teraz jest kupowany Brent, który jest o ok. 30 dolarów droższy za baryłkę niż ten, który jest uwzględniany przy marży, to ta marża będzie się rozjeżdżała z rzeczywistością i nie jest ona odpowiednikiem realnej marży, jaka ma miejsce, ponieważ realna marża jest tajemnicą handlową przedsiębiorstwa, spółki?

To jest naprawdę niecodzienne. Jeśli licealiści się nam przysłuchują, to warto, żeby zwrócili uwagę na to, że Platforma Obywatelska ma pretensje do rządu o to, że spółka Skarbu Państwa przynosi zyski. A jaka jest różnica? W ciągu jednego roku. Panie pośle, naprawdę jest pan tak nadpobudliwy, że obawiam się o pana stan zdrowia o tej godzinie.

To jest naprawdę idealny przykład. A jeśli pan myśli, że sprzedaż paliw na stacjach benzynowych i ogólna sprzedaż na stacjach paliw ma wpływ na zyski osiągane przez Orlen, to chciałbym panu powiedzieć - też zapraszam na korepetycje - że w przypadku zysków Orlenu sprzedaż paliw wynosi wyłącznie 13% udziału w całości zysków osiąganych przez Orlen, ponieważ Orlen osiąga zyski przede wszystkim z działalności rafineryjnej i petrochemicznej. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, jeszcze będzie krótkie sprostowanie, bo pan wielokrotnie odnosił się do pana posła Cezarego Tomczyka. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Panie Ministrze!

A więc strategia Orlenu, o której pan mówił, wygląda mniej więcej tak: dolar się umacnia - paliwo na Orlenie drożeje, dolar traci na wartości - paliwo na Orlenie drożeje, cena baryłki ropy wzrasta - paliwo na Orlenie drożeje, cena baryłki ropy spada - paliwo na Orlenie drożeje. Ostatnie zdanie, panie marszałku. 3300% wynosi wzrost marży w Orlenie i w Lotosie, zyski Orlenu i Lotosu są najwyższe w historii. Panie ministrze, czyim kosztem są te zyski? Przecież one, jeszcze raz powtórzę, nie są kosztem jakiegoś abstrakcyjnego bytu, ludzi, którzy żyją gdzieś w Ameryce Południowej. To są zyski wypracowane na Polakach, którzy płacą na stacjach benzynowych dzisiaj gigantyczne kwoty za benzynę. Ostatni wykres, bo pan przecież lubi dane. Panie ministrze, szanowni państwo, benzyna w Europie, w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich czterech miesięcy gdzie wzrosła najbardziej? W Polsce. To jest pierwszy wynik.

Kolejne pytanie będzie skierowane do ministra funduszy i polityki regionalnej, a zadawać je będą panowie posłowie Mariusz Trepka i Marek Polak.

Proszę teraz pana posła Mariusza Trepkę. Panie Marszałku! Pani Minister! Konkurs wdrażania innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez wdrażanie innowacyjnego produktu lub wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego. Co ważne, innowacja nie musi oznaczać wymyślania produktu od początku, często wystarczy znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących materiałów czy technologii. Innowacje są dostępne dla każdej firmy. Dzięki dotacji przedsiębiorcy będą mogli sfinansować każdy z etapów inwestycji, począwszy od analizy rynku, poprzez zakup licencji, prace dostosowawcze, aż po nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń. Pani Minister! Od kiedy przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do konkursu? Jakie środki europejskie zostały już przekazane w tym obszarze? Jakie zmiany występuję w tej edycji konkursu? Do kiedy firmy będą musiały zrealizować swoje zadania, aby nie utraciły dofinansowania? Ile wynosi maksymalna kwota dotacji? Kontynuacja pytania - kolega Marek Polak. Wysoka Izbo! Pani Minister! Aby przedsiębiorcy mogli realizować projekty do końca 2023 r., do składanych wniosków będą musieli dołączyć wszystkie wymagane decyzje administracyjne, a czas na składanie wniosków to niewiele ponad 3,5 tygodnia, bo od 12 lipca do 5 sierpnia. Dziękuję bardzo. Teraz już poprosimy panią minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Młodzieży! Bardzo dziękuję za to pytanie. Konkurs, który został ogłoszony, wdrażanie innowacji przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dotyczy programu ˝Polska Wschodnia˝ dla perspektywy 2014-2020 i ma to pewne związki z kwestiami terminów. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, od kiedy przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do konkursu, konkurs został ogłoszony 31 maja i od wtedy przedsiębiorcy mają możliwość zapoznania się z dokumentacją konkursową, wnioskiem aplikacyjnym i wymaganymi dokumentami niezbędnymi do przedłożenia razem z wnioskiem.

Jeżeli chodzi o realizację tego działania, czyli wdrażanie innowacji przez MŚP, od początku uruchomienia programu do chwili obecnej na te działania zostało przeznaczone 800 mln zł. Generalnie, szanowni państwo, ten konkurs został ogłoszony po 2 latach jego niebycia w ramach ogłaszanych naborów. Jesteśmy na etapie kończenia perspektywy finansowej 2014-2020.

W związku z tym, że pojawiły się oszczędności w programie ˝Polska Wschodnia˝ i mamy środki, które możemy wykorzystać na pewne działania w ramach tego programu, zdecydowaliśmy o przeznaczeniu puli środków właśnie na te działania, na wdrażanie innowacji przez MŚP, po to żeby wzmocnić ten sektor przedsiębiorczości, który ucierpiał w wyniku pandemii COVID-19 i w wyniku działań związanych z wojną w Ukrainie. A więc chcemy, aby przedsiębiorcy mogli zrealizować te wnioski.

Czyli, po pierwsze, rezygnujemy z działań związanych z pracami budowlanymi, tak aby nie trzeba było stawiać hal produkcyjnych, budować budynków, tylko żeby przedsiębiorcy w ramach tego konkursu mogli zakupić maszyny, urządzenia niezbędne do wdrażania innowacji w swoich firmach, tak aby właśnie zdążyć z tym terminem do 31 grudnia 2023 r.

Nie musi to być innowacyjność na skalę regionalną, wystarczy, że będzie to innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa. Zmniejszono wymogi dotyczące przynależności firmy do powiązania kooperacyjnego, a także wymagania dotyczące ilości dokumentacji niezbędnej do przedstawienia tego warunku. Kwestia związana z uzyskaniem chociażby pożyczki na realizację danej inwestycji jest obligatoryjna na moment podpisania umowy z wnioskodawcą, a nie złożenia dokumentów.

Maksymalna wartość dofinansowania, którą może uzyskać przedsiębiorca, to 10 mln zł. Jeżeli chodzi właśnie o tę maksymalną kwotę dotacji, jest to 10 mln zł. Budżet na konkurs na chwilę obecną wynosi 30 mln zł, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy na etapie zamykania programu, pojawiają się oszczędności w ramach różnych innych działań, które są realizowane w mniejszej skali.

A więc chcemy wybrać projekty do dofinansowania, stworzyć listę rezerwową, tak aby w momencie pojawienia się oszczędności można było podpisywać umowy z innymi wnioskodawcami, którzy zostaną wybrani. Jeżeli beneficjenci przemyślą swoje projekty, jeżeli będą to projekty takie, o których myślimy, czyli zakup urządzeń, zakup maszyn, doposażenie przedsiębiorstwa, niezbędne małe inwestycje w przedsiębiorstwach - tak, wtedy zdążą.

Na chwilę obecną nie ma zgody Komisji na to wydłużenie, więc 31 grudnia 2023 r. to jest termin obowiązujący. Bardzo dziękuję, pani minister. Pani Minister! Bardzo dziękuję za tę informację, bo to jest potrzebna informacja, jeśli chodzi właśnie o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

Może uda się jeszcze więcej, wszystko zależy od tego, jakie będą się pojawiać oszczędności.

Przystępujemy do kolejnych pytań, które są skierowane do ministra infrastruktury. Dotyczą one wprowadzania rozwiązań należycie chroniących bezpieczeństwo dowodów rejestracyjnych samochodów. Pytania będzie zadawał pan poseł Jarosław Gonciarz, a odpowiadał na nie będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Rafał Weber. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych zawiera przepisy określające specjalne wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń, jakie powinny posiadać dokumenty wydawane przez władze publiczne. Dowody rejestracyjne nie spełniają aktualnie ustawowych wymagań. W celu poprawy ich bezpieczeństwa potrzebna jest zmiana technologii, w której wykonywany jest dokument. Według założeń ustawy papier półsyntetyczny powinien być zabezpieczony chemicznie, a w świetle ultrafioletowym nie powinien wykazać luminescencji. Pragnę zapytać, czy ministerstwo zamierza się przygotować na wdrożenie rozwiązań skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa dowodów rejestracyjnych samochodów. Dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana ministra. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Odnosząc się do pytania, bardzo ważnego, które pan zadał, i w ogóle do zagadnienia związanego z bezpieczeństwem dokumentów publicznych, chcę poinformować, że w zakresie właściwości ministra infrastruktury w związku z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych zostało wydane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 maja br., które zmieniło rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. To rozporządzenie weszło w życie 16 maja br. Do 12 lipca br. będą obowiązywać przepisy przejściowe, a od tego dnia już przepisy kompleksowe. Rozporządzenie to wprowadziło nowy wzór dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, to jest dokumentów publicznych kategorii pierwszej. We wzorach oraz opisach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego uwzględnione zostały wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie o dokumentach publicznych. Zmiany ujęte w naszym rozporządzeniu są zgodne z rekomendacjami Komisji do spraw dokumentów publicznych, tak że ta kwestia, o której wspomniał pan poseł Gonciarz, że obecnie dowody rejestracyjne nie spełniają wymagań ustawowych, zostanie rozwiązana tym rozporządzeniem, w sposób pełny od 12 lipca br., bo do tego obligowała nas ustawa, którą wcześniej przytoczyłem. Ponadto informuję, że zmianie uwzględniającej minimalne zabezpieczenia określone w ustawie o dokumentach publicznych uległ również wzór profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 kwietnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów obowiązuje od 1 maja br.

Na koniec wyjaśniam, że ministrem właściwym w zakresie ustawy o dokumentach publicznych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Ponownie prosimy o zadanie pytania pana posła Jarosława Gonciarza. Dziękuję. Pan minister w pierwszej części bardzo wyczerpująco odpowiedział na zadane przeze mnie pytanie, jednak aby tradycji stało się zadość, chciałbym dopytać, czy ministerstwo analizuje potrzebę zmian w odniesieniu do innych dokumentów publicznych, tak aby spełniały wymagania zgodne z ustawą. Dziękuję. Prosimy pana ministra. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Tak, planujemy tego typu zmiany.

Natomiast w odniesieniu do dokumentów kategorii trzeciej zgodnie z ustawą mamy 5 lat od dnia wejścia w życie tych przepisów, czyli 5 lat od 12 lipca 2019 r., aby tę sprawę uregulować, tak więc dokładnie 12 lipca 2024 r. dokumenty kategorii trzeciej będą musiały posiadać zabezpieczenia wskazane w ustawie.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Kolejne pytania będą zadawać panie posłanki Joanna Borowiak i Barbara Bartuś. Dotyczyć będą przygotowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązań systemowych i instrumentów wsparcia dla polskich seniorów. Odpowiedzi na te pytania udzieli pan minister Stanisław Szwed. Zatem proszę panią poseł Joannę Borowiak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rodzina i seniorzy są w centrum uwagi i działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kolejną kadencję przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania systemowe, instrumenty, których ideą jest wsparcie i poprawa sytuacji osób starszych, emerytów, rencistów, wśród których znaczną grupę stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

Tu widać realną różnicę.

Wiemy, że w roku bieżącym to wsparcie będzie jeszcze wyższe, jeszcze bardziej znaczące, ta kwota zostanie zwiększona. Panie ministrze, uprzejmie poproszę o odpowiedź na pytanie: Jakiego rodzaju, w jakiej wysokości wsparcie finansowe zostało zaplanowane dla polskich seniorów, emerytów i rencistów, w bieżącym roku? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy pana ministra. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie dotyczące polityki senioralnej realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że te ostatnie lata to dobry okres dla emerytów i rencistów. Działania, które podejmujemy, mają służyć temu, aby naszym emerytom żyło się lepiej i godniej.

Przypomnę, że tegoroczna waloryzacja jest wyższa niż mogłoby to wynikać z ogólnie przyjętych norm, które przyjmowaliśmy.

Warto też podkreślić, jak wzrastała minimalna emerytura w ostatnich latach, bo przypomnę, że w 2015 r. najniższa emerytura wynosiła 880 zł.

Warto oczywiście to przypomnieć, bo wszyscy o tym doskonale wiedzą, szczególnie emeryci.

Sejm przegłosował już stosowną ustawę, która jest w tej chwili w Senacie. Przypomnę, że jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to ona obejmuje wszystkich ubezpieczonych, tych, którzy są ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w KRUS, mają świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy świadczenia mundurowe.

Czternasta emerytura na podobnych zasadach jak trzynasta emerytura, z tym że wprowadziliśmy limit kwoty uprawniającej do pełnej najniższej emerytury, tj. kwota 2900 zł świadczenia emerytalnego.

O podatku już wspomniałem, zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura zwolnione są od podatku. Pani przewodnicząca o tym wspomniała, ale warto jeszcze przypomnieć, że łącznie w 2020 r. waloryzacja trzynastej i czternastej emerytury to będzie prawie 43 mld zł.

Czas się kończy, ale chcę wspomnieć jeszcze o dodatku osłonowym, który jest zawarty w tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przeznaczamy na to ponad 4 mld zł. Osoby, które mają najtrudniejszą sytuację, a dotyczy to również gospodarstw senioralnych, mogą z tego skorzystać.

To tyle w telegraficznym skrócie, bo oczywiście programów, które realizujemy, jest bardzo dużo, ale czas już minął. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękujemy za początkową odpowiedź, w której pan mówił o przywracaniu godności seniorom, przywracaniu godności emerytom i o waloryzacjach, które realizuje obecny rząd, który jest od 2015 r.

Ale to był efekt tego, jakie rozwiązania przyjął ówczesny rząd.

Warto o tym przypominać, bo dzisiaj, jak żyje nam się coraz lepiej, to zapominamy. Chciałam w tym moim, już (Dzwonek) skończonym, czasie dopytać jeszcze o jedno bardzo, bardzo ważne rozwiązanie - o emeryturę ˝Mama 4+˝

Ile osób, ile kobiet, czy nie tylko kobiet, skorzystało z tego świadczenia? Czy są składane nowe wnioski i jakie to są ewentualnie kwoty - jak pan minister ma te dane - które na ten cel są przeznaczane? Bardzo dziękuję. Prosimy pana ministra. Dziękuję bardzo za te uzupełniające pytania.

I to rozwiązanie, które wprowadziliśmy, zapewnia tym osobom najniższe świadczenie, czyli w tym przypadku kwotę 1388,44 zł.

Oczywiście generalnie to dotyczy matek, ale jest też kilkuset ojców, którzy z tego programu korzystają.

I tak jak powiedziałem, to są te dwa mechanizmy.

Myślę, że to też jest bardzo dobrze przyjęte rozwiązanie, które pomaga tym osobom godnie żyć. Dziękuję bardzo.

Odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani minister Anna Gembicka. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Rolnictwo to jeden z najważniejszych działów naszej gospodarki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości poczynił milowe kroki dla bezpieczeństwa polskiego rolnictwa i rolników. Rewolucyjne zmiany objęły rolniczy system rent i emerytur. Proszę o przedstawienie szczegółów tych zmian. Proszę także wskazać, jak obecnie co do wielkości wyglądają polskie obszary rolnicze na tle innych państw. Chciałbym poprosić jeszcze o przedstawienie, w jaki sposób zmieniła się wysokość emerytur rolniczych z KRUS na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ilu rolników pobiera obecnie to świadczenie? Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Po 30 latach istnienia przepisu w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, który nakazywał zaprzestanie działalności rolniczej rolnikowi, który przechodził na emeryturę, jeżeli chciał otrzymać pełne świadczenie, nasz rząd zaproponował zmiany dotyczące rezygnacji z tego warunku. Od tej pory rolnika, który przechodzi na emeryturę, już nie obowiązuje ten warunek, że musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Był to także jeden z postulatów w naszym programie dla polskiej wsi. Warto podkreślić, że te zmiany są jednoznacznie korzystne dla rolników. Myślę, że o tym świadczy chociażby fakt, że w czasie debaty sejmowej, także w Senacie, wszyscy parlamentarzyści głosowali za tą ustawą. Problem dotyczący warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przy przechodzeniu na emeryturę był zwłaszcza w ostatnich latach stale podnoszony przez rolników indywidualnych, przez samorząd rolniczy, przez związki zawodowe i organizacje rolnicze, oczywiście także przez parlamentarzystów. Ten wymóg był dla wielu rolników niezrozumiały, bo w żadnym innym zawodzie nie było takiej konieczności, żeby przy przechodzeniu na emeryturę, jeżeli chciało się otrzymywać ją w pełnej wysokości, trzeba było swój warsztat pracy sprzedawać, zbywać czy komuś przekazywać. W związku z tym można powiedzieć, że to jest wprowadzenie pewnej sprawiedliwości dziejowej w stosunku do rolników. Oprócz tego nowelizacja ustawy, która już została uchwalona, podpisana przez pana prezydenta i niedługo wchodzi w życie, wprowadziła zmiany dotyczące przepisów, których negatywne skutki obowiązywania powodowały kłopoty dla rolników w ich codziennym funkcjonowaniu.

Jeżeli chodzi o te zbiegi, są to takie sytuacje jak korzystanie ze świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali oni skierowani przez powiatowy urząd pracy, stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne podmioty niż powiatowy urząd pracy, pełnienie czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Chodzi także o osoby, które odbywają służbę zastępczą. Jest to wysokość wynosząca 1% podstawowego świadczenia za każdy rok służby. Oprócz tego kolejną zmianą, która też była postulowana przez organizacje rolnicze, jest umożliwienie KRUS-owi podejmowania działań w celu poprawy stanu zdrowia także emerytów rolniczych. Chodzi o umożliwienie im korzystania z rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji, a także umożliwienie skierowania osób ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne do zakładów rehabilitacji. Chodzi o te osoby, które skorzystają właśnie z możliwości kontynuowania działalności rolniczej przy przechodzeniu na emeryturę, oraz o te osoby, które będą miały doliczane do emerytury również okresy odbywania służby wojskowej. Oprócz tego, jeżeli chodzi o ogólną liczbę świadczeniobiorców, razem z rencistami, mamy ponad 1 mln samych emerytur. I to, co, jak myślę, jest bardzo ważne - te zmiany, o których powiedziałam, to jest, można powiedzieć, pierwsza część zmian, bo w kolejnej nowelizacji chcemy zmienić zasady dotyczące waloryzacji świadczeń emerytalnych. Oprócz tego wspólnie z ministerstwem rodziny pracujemy nad uregulowaniem sprawy zbiegu tytułów emerytalnych w systemie powszechnym i w systemie rolniczym.

Kolejne pytanie, pani poseł Gabriela Masłowska. Bardzo proszę, pani poseł. Korzystając z pani obecności, chciałabym zapytać o sytuację rolników ekologicznych.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Jednym z tych działań jest powołanie w ostatnim czasie polskiej grupy spożywczej.

Ostatnio także w Sejmie procedowaliśmy nad ustawą o rolnictwie ekologicznym, która jest implementacją przepisów unijnych dotyczących funkcjonowania rolnictwa ekologicznego.

Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej, czyli tworzenia tzw. rejestru ciąż, o przedstawienie której wnosił Koalicyjny Klub Poselski Lewicy. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców lub posłów nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 1 minutę. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wysoka Izbo! Zadajemy dziś pytanie na temat rejestru ciąż, rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie włączenia do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących ciąż Polek. Usłyszymy zapewne od pana ministra, że chodzi o proste, techniczne rozwiązanie, wprowadzenie narzędzia, które ułatwi świadczenie lepszych usług medycznych kobietom w ciąży. I rzeczywiście - rejestr ciąż to narzędzie i właśnie dlatego tak ważne jest pytanie, do czego będzie faktycznie używane, bo każdego narzędzia można użyć w dobrym albo w złym celu. Za pomocą siekiery można porąbać drewno na opał, ale można także skrzywdzić. Tak samo jest z rejestrem ciąż. Można go użyć, żeby wzmocnić ochronę ciężarnych kobiet, ale w rękach władzy, która urządziła kobietom piekło, ograniczyła prawo do legalnej aborcji, pozbawiła awaryjnej antykoncepcji, to narzędzie, niestety, może okazać się bardzo niebezpieczne. Bo prawo nie działa w próżni, kontekst ma znaczenie. Tak jak ma znaczenie, czy spis ludności na Krymie przeprowadzałaby Rosja czy Ukraina, tak ma znaczenie, czy rejestr ciąż wprowadza Dania czy Salwador, Szwecja czy Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Jest różnica, czy rejestr ciąż prowadzi państwo opiekuńcze, które kobietom zapewnia prawo wyboru, czy państwo wobec kobiet opresyjne, z niemal całkowitym zakazem aborcji. Niestety, Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest państwem wobec kobiet opresyjnym.

Dalsza część wypowiedzi - pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica. O, przepraszam. Pani Daria Gosek-Popiołek, przepraszam, także Lewica. Wysoka Izbo! Żyjemy w kraju, w którym wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył i tak już bardzo restrykcyjne przepisy antyaborcyjne, zwłaszcza że choć pseudo-Trybunał Konstytucyjny teoretycznie stwierdził, że możliwe jest przerwanie ciąży, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest skutkiem czynu zabronionego, to jednak prokuratura ministra Ziobry ma inne podejście. Dowodem na to jest to, co wydarzyło się w Białymstoku. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przerywania ciąży prokuratura sprawdzała, czy w szpitalu przeprowadzono aborcję i dlaczego. Wystąpiono o dane pacjenta. Dopiero doniesienia medialne i nacisk opinii publicznej sprawiły, że śledczy zrezygnowali z dalszych działań. I takiej prokuraturze dał pan minister dostęp do wrażliwych medycznych danych pacjenta, prokuraturze, która gotowa jest ścigać kobiety, które w desperacji chcą wyjeżdżać za granicę, by w godnych, bezpiecznych warunkach przeprowadzić zabieg przerywania ciąży, prokuraturze, która gotowa jest ścigać bliskich, partnera, koleżanki. Nie ma co się dziwić, że brak zaufania do państwa, obawa przed prokuraturą, brak wiary w to, że ktokolwiek pomoże w tej sytuacji, sprawia, że niechęć, lęk kobiet przed zajściem w ciążę w Polsce wzrasta. Dalszy ciąg - pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, klub Lewicy. Wczoraj Sejm zdecydował kolejny już raz, że nie będzie dawał prokuratorom 7-dniowego terminu na wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej na przerwanie ciąży pochodzącej z gwałtu. Zgwałcone kobiety nie zgłaszają, że są w ciąży ze swoim oprawcą, bo prokuratorzy ze względu na terminy prowadzenia śledztw wydają te decyzje po 3-6 miesiącach, uniemożliwiając legalne przerwanie tych ciąż. Te skrzywdzone kobiety polskie państwo zmusza do czynów nielegalnych, mówiąc: radźcie sobie same, a teraz będzie je inwigilować. Nie do gwałciciela przyjdzie prokurator, ale do zgwałconej kobiety - z pytaniem, co zrobiła pani z ciążą. Uderzacie także w matki, których dzieci urodziłyby się obarczone śmiertelnymi wadami, w te Polki, dla których od wyroku pseudo-Trybunału Konstytucyjnego ważniejsza jest miłość i współczucie, w te kobiety, które dotknęła tragedia, a ich wyczekane dzieci będą skazane na cierpienie i śmierć, bo te Polki przerywają ciążę, zanim płody i dzieci zaczną odczuwać ból. Teraz te kobiety będziecie inwigilować. W chwili największej życiowej tragedii naślecie na nie policjantów z pytaniem, co zrobiła pani z płodem obarczonym wadą letalną. I trzecia grupa kobiet - kobiety, które poroniły swoje upragnione dziecko, będziecie pytać: A może jednak nie chciała pani dziecka i dlatego nie jest pani w ciąży? Zgwałcone, przeżywające żałobę, przeżywające tragedie osobiste - w te kobiety pod płaszczykiem rejestru medycznego uderzacie.

Teraz proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Waldemara Kraskę. Bardzo proszę, panie ministrze.

Wysoka Izbo! Na wstępie chciałem powiedzieć, i podkreślić to z wielką mocą, że wprowadzenie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej nie tworzy rejestru ciąż. Państwo wielokrotnie powtarzali już w swoich wystąpieniach, że stworzyliśmy rejestr ciąż. Takiego rejestru nie tworzymy, a także nie tworzymy żadnego innego rejestru. Powtórzę to jeszcze raz, po raz trzeci powtórzę: nie tworzymy żadnego rejestru ciąż. Chcemy, aby dane zawarte w Systemie Informacji Medycznej zapewniały pracownikom medycznym jak najszerszy dostęp do danych konkretnego pacjenta, tak aby udzielanie świadczeń medycznych odbywało się na jak najwyższym poziomie i bez szkody dla zdrowia pacjenta. Na pewno padną pytania, kto jest uprawniony do dostępu do takich danych. A więc, po pierwsze, pracownik medyczny, który wytworzył daną dokumentację elektroniczną, po drugie, pracownik medyczny, który pracuje w danej placówce i będzie odpowiadał za dalszą prowadzoną diagnostykę lub proces leczenia. Trzecią osobą, która jest uprawniona do dostępu do tych danych, czyli do Systemu Informacji Medycznej, jest lekarz, pielęgniarka lub położna pracujący w POZ, lekarz rodzinny. I czwartą osobą, która będzie miała dostęp do tych danych, jest każdy pracownik medyczny - wtedy kiedy jest stan zagrożenia życia pacjenta, który się zgłasza, np. z wypadku, na SOR. Proszę państwa, nie muszę chyba przekonywać lekarzy, którzy znajdują się na tej sali, jak ważna jest informacja o tym, czy osoba jest w ciąży, czy też nie.

Wprowadzamy informację o wyrobach medycznych zaimplantowanych pacjentowi, czyli tzw. implantach.

To jest bardzo ważne dla lekarza, który będzie tego pacjenta kierował.

Też nie muszę nikogo przekonywać do tego, że w stanach nagłych ta informacja jest bezcenna.

Przyjeżdża młoda osoba z wypadku, nieprzytomna.

Po raz czwarty powtarzam: takiego rejestru nie wprowadzamy. To nie wzięło się znikąd.

Ta komisja zakończyła pracę w roku 2013. Także Polska w roku 2013 nie wnosiła żadnych zastrzeżeń co do tego rozporządzenia, które zacznie obowiązywać już w przyszłym roku. W tej chwili Unia Europejska kończy prace nad tym rozporządzeniem. Szanowni Państwo!

Wręcz odwrotnie, to jest dla ich bezpieczeństwa.

Jeżeli nie, to oczywiście czekam na pytania i ewentualne odpowiedzi. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Informuję, że zgłosili się posłowie do dyskusji. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zapisać się do głosu? Otwieram dyskusję. Jako pierwsza pani poseł Anna Kwiecień, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Niestety z przykrością wysłuchałam tych wystąpień szanownych koleżanek z uwagi na to, że są one obarczone kłamstwem. Wiecie doskonale, drogie panie, że nie ma czegoś takiego jak rejestr ciąż.

I w sytuacji, kiedy, nie daj Boże, Polka pojedzie za granicę.

Natomiast ważne jest to, że gdy kobieta, nie daj Boże, trafi np. w Grecji w sytuacji stanu zagrożenia życia do szpitala, to żeby lekarz wiedział, że np. nie może jej zlecić tomografii komputerowej, która jest niczym innym jak jednorazową dawką 100 zdjęć tradycyjnych rentgenowskich, w sytuacji kiedy ona jest w ciąży.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ze zdumieniem słuchamy, jak bardzo pan nie rozumie, o czym jest ta rozmowa. Otóż doprowadziliście Polskę do stanu takiego, że Polki, młode kobiety, boją się zachodzić w ciążę - waszym zakazem aborcji, zabraniem Polkom in vitro.

Prowadzicie politykę antykobiecą i antydemograficzną i nawet wasza pani Otóż ma to służyć temu, żeby ciążę wraz z lekarzem prowadził prokurator pana Ziobry. I do tego chcecie doprowadzić, żeby młode kobiety bały się jeszcze bardziej. Stosujecie język pogardy i nienawiści do Polek (Dzwonek), których nie rozumiecie i nie chcecie zrozumieć.

Najpierw Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło całkowity zakaz aborcji, potem domagało się od innych krajów, by zakazać aborcji Polkom. Na szczęście rząd Czech odmówił wprowadzenia takiego zakazu. Teraz PiS chce rejestrować każdą ciążę. Nic dziwnego, że Polki się boją, czują się osaczone i kontrolowane. Nie chcą być nękane przez policjanta pytaniami o dalszy przebieg ciąży. Boją się zachodzić w ciążę, a gdy zajdą, to boją się iść do lekarza, by ciąża nie została zarejestrowana. Dlatego pytam w ich imieniu: Po co wam, po co prokuratorowi informacja na temat każdej ciąży? Czy będzie prowadzone śledztwo, jeśli dziecko się nie urodzi? Czy prokuratura zamierza stworzyć specjalny wydział do kontrolowania stanu i losów każdej ciąży? A ciąż było znacznie więcej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim ta informacja o ciąży znajdzie się w tzw. rejestrze, to najpierw kobieta musi mieć dostęp do ginekologa. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2018 r. pokazał, jaka jest smutna rzeczywistość w Polsce, jak fatalny dostęp do opieki ginekologiczno-położniczej mają Polki w naszym kraju - tej refundowanej, finansowanej z budżetu państwa. Szczególnie zły dostęp mają kobiety spoza dużych aglomeracji. Wiejska droga do ginekologa jest wybrukowana wielkimi wybojami. Więc zanim pan minister zacznie zajmować się takimi szczegółami, które teoretycznie do niczego nie są potrzebne i przez nikogo nie są oczekiwane, warto zająć się podstawowymi sprawami dotyczącymi opieki ginekologiczno-położniczej. Także i tymi paniami, tymi parami i małżeństwami, które czekają na dzieci.

Szczęść Boże! - polskim dzieciom, zwłaszcza narodzonym, nienarodzonym. To jest oczywiście groteska, że państwo, którzy popieraliście projekty rejestru szprycowanych, teraz oburzacie się na rejestrowanie ludzi wedle innych kategorii.

Ja akurat nie popieram centralizacji i odzierania ludzi z prywatności pod pretekstem spieszenia im z pomocą. Skorzystam z obecności ministra Kraski. Chcę zapytać pana, panie ministrze, bo ministerstwo pańskie nie odpowiada na piśmie: Co pan robił, zanim zaczął się pański oficjalny życiorys w Wikipedii?

Jest pan poseł Suchoń? Bardzo proszę. Nie ma pana posła.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chcę przypomnieć, że bycie w ciąży to jest normalny stan, jaki przeżywa kobieta. Mówię to jako kobieta, która przeżyła cztery ciąże, i z tego jestem dumna. Trzeba mówić o opiece nad kobietą w ciąży, a nie o aborcji. Chcę przypomnieć, że zbieranie danych nie jest niczym nowym. Tu mam pytanie do pana ministra. Czy przypadkiem nie jest tak, że we wszystkich krajach europejskich będą takie same standardy, że kobieta będzie zarejestrowana, tak aby zająć się nią w tym stanie, w którym ona przeżywa poczęcie nowego życia? Bo życie jest najcenniejszym darem, o który winniśmy wszyscy zadbać, a przede wszystkim politycy.

Trzeba przyznać, że PiS jest konsekwentny w działaniu przeciwko kobietom. Dziś do zakazów dokłada Polkom rejestr ciąż. więc dziś skupię się na tym, co my, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, zrobimy, kiedy PiS trafi na śmietnik historii. Otóż całościowo rozwiążemy kwestie zdrowotne kobiet. Zapewnimy bezpłatne badania prenatalne. zagwarantujemy łatwy dostęp do bezpłatnej antykoncepcji, dostęp do tabletki dzień po bez recepty, wrócą lekcje edukacji seksualnej w szkołach i stałe wsparcie finansowe oraz opieka medyczna w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego. Wrócimy też do bezpłatnego in vitro. Wprowadzimy także nową umowę społeczną, w której zagwarantujemy każdej Polce prawo do podjęcia przez nią po konsultacji z psychologiem i lekarzem indywidualnej decyzji o przerwaniu ciąży do 12. tygodnia w bezpiecznych warunkach, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej. Kobiety muszą mieć prawo do podejmowania osobistej decyzji dotyczącej macierzyństwa w zgodzie z własnym sumieniem, muszą mieć zapewnioną kompleksową opiekę (Dzwonek), muszą być bezpieczne i mieć zagwarantowane prawo wyboru. Wysoki Sejmie!

Ale przyszedł taki czas, kiedy Lewica rządziła i ustąpiła w tych sprawach, poszukując kompromisu. Ten kompromis został zawarty. To dla Lewicy było za mało, ale chcieliśmy uszanować wszystkie poglądy, nie tworzyć państwa wyznaniowego, które będzie nakazywało wszystkim. Bo dzisiaj to jest kwestia ciąży, przerywania ciąży, ale jutro pójdziemy dalej, pójdziecie dalej. To jest błąd.

Pani poseł Urszula Pasławska, Koalicja Polska. Ja mam pytanie: Po co PiS-owi rejestr ciąż? Po to, żeby ukryć inflację, po to, żeby odwrócić uwagę od drożyzny, od wysokich rat kredytów? Bo chyba nie po to, żeby wesprzeć kobiety, bo to nie ma nic wspólnego ze wsparciem kobiet. Jeżeli chcecie państwo wspierać kobiety, to w Polsce miliony kobiet niewidzialnych dla systemu potrzebują wsparcia, kobiet, które pragną dzieci, a nie stać ich na in vitro, kobiet po depresjach poporodowych, po poronieniach. Czy będzie miała prawo niewyrażenia takiej zgody? Po trzecie, co z naszymi prawami obywatelskimi, osobistymi?

Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050.

Wysoka Izbo! Pewnie w normalnym kraju elektroniczny rejestr byłby dobrym pomysłem, ale w Polsce? W Polsce system opłat za drogi śledzi kierowców nawet wtedy, kiedy jeżdżą po drogach bezpłatnych. W Polsce urzędy skarbowe od lipca będą mogły wchodzić na konta Polek i Polaków bez żadnej przyczyny, według swojego widzimisię. W Polsce do każdego cyfrowego rejestru mają dostęp np. Wojska Obrony Terytorialnej, bo taką ustawę sobie uchwaliliście. W Polsce do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych ostatnio dostały dostęp trzy czy cztery kolejne organy, zupełnie nie wiadomo po co. Baza PESEL w Polsce i nasze numery telefonów zostały przekazane rachmistrzom spisowym pod pozorem ułatwienia narodowego spisu rolnego.

Pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2023 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywać jednolity system informacji medycznej, w tym o zdarzeniach medycznych. Zawarte w systemie informacji medycznej dane nie są czymś wyjątkowym. Zgodnie z obowiązującymi standardami każda porada lekarska obejmuje wywiad oraz, jeśli nie jest to teleporada, badanie fizykalne. Udzielający porady medyk pyta o wszystkie istotne sprawy, o alergie, przebyte zabiegi operacyjne, sposoby zaopatrzenia, choroby w rodzinie, przyjmowane leki, kobiety są pytane o pierwszą, ostatnią miesiączkę, ilość porodów, poronienia, również o ciąże czy grupę krwi. Nie tworzy się oddzielnych katalogów złamanych nóg leczonych operacyjnie ze wstawieniem implantów, alergii na sierść kota, osób z określoną grupą krwi czy kobiet będących w ciąży. Dlaczego zatem do e-dokumentacji wpisuje się te dane? Bo są bardzo ważne z punktu widzenia możliwej diagnostyki i zastosowanej terapii.

No to przypomnijmy, standardem europejskim jest in vitro, standardem europejskim jest aborcja dla kobiety zgodnie z jej wolą do 12. tygodnia ciąży, standardem europejskim jest to, że antykoncepcja awaryjna jest bez recepty. Wy tego wszystkiego zabraniacie polskim kobietom. Powiem więcej, zabroniliście im również aborcji w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu, w dramatycznej dla nich sytuacji. Natomiast tak chętnie zajmujecie się rejestrem ciąż. do którego dostęp poza lekarzami będą mieli również prokurator i sąd w ramach artykułu Kodeksu karnego. Ja bym chciała, żebyście wy się zajęli innym rejestrem. Polska była na czele rankingu, najbardziej czarnego rankingu dotyczącego dodatkowych zgonów w czasie pandemii. Średnia europejska - 12,5%, jeśli chodzi o te nadmiarowe zgony.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pomysł Ministerstwa Zdrowia, żeby w Systemie Informacji Medycznej przechowywać kolejne informacje, np. o alergiach czy ciążach, w normalnym państwie nie wzbudziłby aż takich emocji, jakie mamy obecnie w Polsce. Proszę państwa, ministerstwo ignoruje głosy kobiet, które w obecnej sytuacji prawnej i politycznej, od jesieni 2020 r., po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, boją się zachodzić w ciążę i mają uzasadnione obawy przed nadmierną ingerencją państwa w ich prywatność. Pan minister doskonale wie, że oprócz pracowników medycznych dostęp do tego systemu będą mieli także, zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sędzia i prokurator. Polki nie ufają państwu ani państwa rządom, Polki obawiają się prokuratury. Polki boją się, że nie uzyskają pomocy, kiedy znajdą się w kryzysowej sytuacji. Panie Ministrze! Czy pacjentki będą wiedziały, kto, kiedy i w jakim celu sprawdzał ich dane medyczne?

W Polsce musimy przywrócić normalność. Polskie kobiety nie mogą się bać zachodzić w ciążę. Zamiast cieszyć się dziś z poczęcia, kobiety boją się, idąc na pierwszą wizytę do lekarza, czy będzie dobrze, bo jak nie, to co dalej. Dziękuję. Wysoka Izbo! Szanowne Panie! Pani się nie śmieje, mamy normalne Ministerstwo Zdrowia, normalny rząd, taki, który dba o zdrowie kobiet.

Przed chwilą pan minister wyraźnie wytłumaczył, że to jest wymóg Unii Europejskiej, to jest rozszerzenie katalogu gromadzonych danych i przełoży się na zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej.

Panie Ministrze! Nasza reakcja na rejestr ciąż ma po prostu bardzo polski kontekst. Jest to kontekst strachu wobec zakazu aborcji w Polsce. Jest to kontekst strachu wobec niedostępności ginekologa dla Polek, zwłaszcza tych z małych miejscowości i ze wsi. Niektóre Polki muszą dojeżdżać 50 km do lekarza ginekologa. Opieka okołoporodowa jest na dramatycznie niskim poziomie. Wzrastają umieralność i skala poronień. Kobiety z niepełnosprawnościami - dramatyczny dostęp do opieki lekarskiej, ginekologicznej. Dostęp do ginekologa dla nastolatek tylko pod opieką osoby dorosłej. Nastolatka ma prawo pójść do ginekologa, porozmawiać o swoich problemach, niekoniecznie pod opieką osoby dorosłej czy rodzica.

Panie Ministrze! W krajach, gdzie aborcja jest europejskim standardem, a o tych europejskich standardach było dzisiaj tutaj bardzo dużo, czyli wszędzie poza Polską i Maltą. Bardzo proszę o uciszenie. Ten rejestr to zwykła procedura w ramach cyfryzacji procedur medycznych i z tym się absolutnie zgadzamy. Ale mamy obawy, że w Polsce będzie to straszak na kobiety i źródło prześladowania tych, które przerwą ciążę. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej pacjentki, które są w ciąży obarczonej wadą letalną, słyszą dzisiaj pytanie, czy mają pieniądze, i słyszą dzisiaj sugestię, żeby wyjechały za granicę. Mamy prawo podejrzewać, że prokuratura ministra Ziobry może używać tego rejestru, aby urządzić polowanie na kobiety, które przerwały ciążę. Chciałabym zapytać, czy w obliczu poszerzenia tego rejestru - mamy pełną świadomość, że ten rejestr funkcjonował - będzie także instrukcja dla lekarzy i być może przypomnienie o tym, że dzisiaj kobiety w Polsce mają prawo przerywać ciążę same, że jest to legalne, a ci lekarze nie mają prawa zadawać pytań (Dzwonek), gdzie to zrobiły, w jaki sposób i dlaczego. Wysoka Izbo! Wsłuchując się w głosy oponentów, na pewno należy potwierdzić jedno: ciąża to nie choroba, a stan niekiedy bardzo wyczekiwany przez kobietę czy małżonków. Dlaczego temat ciąży poruszany w Sejmie budzi zawsze tyle emocji? Przecież od tego, ile się dzieci urodzi, zależy demografia i nasza przyszłość w wielu wymiarach społecznych. Obowiązkiem państwa jest opieka nad kobietą w ciąży, zarówno pomoc socjalna, jak i opieka zdrowotna, a ważnym czynnikiem jest szybka i skuteczna pomoc medyczna w sytuacjach skrajnych czy zagrażających życiu matki i dziecka. Dziś młode kobiety od początku potwierdzenia faktu, że zostaną matkami, szukają dobrego lekarza położnika i informacji, gdzie znajdą najlepszą opiekę. Czemu więc nie rozszerzyć katalogu informacji medycznej o tę tak istotną informację o ciąży, skoro jest to jeden z czynników wspomagających procedury medyczne, a jednocześnie wynika to z zaleceń zespołu powołanego przez Komisję Europejską? Panie ministrze, komu przysługuje dostęp do zbierania informacji i danych w SIM? Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj wyjątkowo nie będzie o polityce, bo ciąża to nie polityka. Dostęp do darmowej antykoncepcji to nie polityka. Decydowanie o swojej płodności to nie polityka. Wysoki standard opieki okołoporodowej to nie polityka. Dostęp do ginekologa, który nie ocenia wyboru kobiet, to nie polityka. Bezdzietność to nie polityka. Legalne zamrażanie komórek jajowych na życzenie to nie polityka. Legalna aborcja to nie polityka. Prawo do surogatki to nie polityka. Każdy mężczyzna korzysta z usług surogatki, bo przecież sam nie rodzi. In vitro to nie polityka. Małżeństwo to nie polityka. Nawet seks to nie polityka.

Pośmialiście się państwo? Ale, pani poseł, czas mija. Ja jeszcze nie zaczęłam, panie marszałku, bo czekam, aż państwo się wyśmieją. Wysoka Izbo! Prawicowa mentalność to nakazy, zakazy, inwigilacja i nadzwyczajne zainteresowanie seksualnością innych. To wynik waszego światopoglądu, kompleksów, fobii i obsesji. Angielska prawica dawno wyzwoliła się z wiktoriańskiej pruderii. Polska z dulszczyzny - nie, bo to waszej prawicowej władzy na rękę. Zamiast logiki - cuda. Ciąża dla was to nie naturalne następstwo połączenia komórki jajowej i plemnika, ale cud poczęcia. Cuda też musicie inwigilować. Zakazując aborcji, doprowadziliście do tego, że kobiety muszą wyjeżdżać ze swojego kraju, teraz chcecie, żeby kobiety w swoim kraju bały się pójść do ginekologa. Dramatów przybędzie, ale co was to obchodzi? Nic.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Panie Posłanki z Opozycji! Polskie kobiety, które zachodzą w ciążę, nie boją się chodzić do ginekologa, a poczęcie to cud i każda jedna kobieta stara się w najwyższym stopniu zadbać o ten cud i wyeliminować każde zagrożenie. A niestety są środki medyczne, które stwarzają zagrożenie. Panie Ministrze! Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Jakie medykamenty, jakie lekarstwa mogą przyczynić się do skutków ubocznych dla ciąży? Czy to tylko kwestie badań rentgenowskich, czy są być może też inne środki medyczne, które zagrażają ciąży?

Też nie ma pani poseł. Pan poseł Jerzy Paul, Prawo i Sprawiedliwość. Też nie ma pana posła. Pani poseł Jagna Marczułajtis-Walczak, Koalicja Obywatelska. Wasze rządy to ograniczanie praw kobiet. Ograniczyliście dostęp do tabletki dzień po i dostęp do legalnego przerywania ciąży. W Zakopanem od kilku lat kobiety mają ograniczony dostęp do porodówki, muszą jeździć do innych miast i tam rodzić dzieci.

Ograniczacie również opiekę wytchnieniową.

Pan poseł Zdzisław Wolski, Lewica. Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra zdrowia o możliwości przestępczego korzystania z Systemu Informacji Medycznej, konkretnie chodzi mi o możliwe cyberataki, o możliwości stosowania przepisów RODO w praktyce w zmodyfikowanym Systemie Informacji Medycznej. Wiemy, że jeżeli chodzi o placówki służby zdrowia, są one pod tym względem dużo gorzej zabezpieczone niż inne branże, nie tylko bankowość. Wiemy, że gwałtownie rośnie ilość ataków hakerskich, na przykład w roku 2020 ofiarą tych ataków padło 18 mln kartotek pacjentów.

Nie ma pana posła. Pan poseł Jarosław Wałęsa, Koalicja Obywatelska. Przepraszam, nie zauważyłem. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jeżeli kobieta trafia w stanie bez kontaktu na jakiś oddział w dowolnym kraju, może to być obcokrajowiec z Unii Europejskiej w Polsce, czy ta informacja jest potrzebna lekarzowi, który podejmuje decyzje diagnostyczne czy lecznicze w sposób pilny, natychmiastowy i błyskawiczny? Wszyscy pytają, kto trafia.

Od zarania dziejów mężczyźni uzurpowali sobie prawo do decydowania o kobietach i o tym, co się z nimi dzieje.

Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej zasadzie: rząd ma sprawować władzę, a to nie jest rząd dusz. Zostawcie w spokoju nasze sumienia i niech każdy decyduje za siebie, jak powinno wyglądać jego życie, szczególnie kobiety. Dlaczego musimy wracać do tego i dyskutować na ten temat w zasadzie codziennie albo bardzo często? Dlaczego nie możemy raz na zawsze potwierdzić tego, co jest rzeczą oczywistą?

Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Pan ma zaufanie do siebie jako lekarz i człowiek o określonej wiedzy. My mamy zaufanie do lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych.

Stąd nie dziwmy się, że Polki obawiają się zapytać: Jakie przesłanki prawne zdecydowały o wprowadzeniu danych o ciąży do Systemu Informacji Medycznej? Drugie pytanie: W jaki sposób Policja, prokuratury i sądy mają dzisiaj dostęp do tej informacji medycznej? Trzecie pytanie: Ile było oficjalnych wniosków złożonych przez organy państwa o dostęp do Systemu Informacji Medycznej?

Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! My mamy normalne państwo, my mamy w tym kraju nienormalną opozycję.

Tą receptą jest totalna aborcja. I tutaj słowo do panów posłów: panowie posłowie, zadecydujcie o sobie, nie o kobietach, o sobie - wazektomia jest też dostępna.

Dlatego zwracam się też do posłów i posłanek z lewej strony, nie majstrujcie panie, panowie (Dzwonek) swoją propagandą przy życiu i zdrowiu kobiet i dzieci, bo wasza propaganda może zabijać. Pani poseł Iwona Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Inwigilacja i kary to kolejny pomysł rządu PiS skierowany do kobiet i do lekarzy. Nadzór i kontrola, a 10-latki do poprawczaka, rodzice dzieci z chorobami SMA muszą poradzić sobie sami. Co roku rodzi się w Polsce ok. 50 dzieci chorych na SMA. Zamiast zapowiadanego rejestru ciąż może wreszcie rząd zajmie się refundacją leków na SMA i możliwością leczenia tych dzieci? Dzieci cierpią, rodzice błagają o pomoc. 10 mln na dziecko to jest ogromna kwota i naprawdę trudno ją zebrać. Mała Zosia, mały Krzyś walczą o życie, walczą o zdrowie, czekają na refundację.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Jak zwykle, wiele hałasu o nic. Gromadzenie danych, w tym danych osobowych, a szczególnie danych wrażliwych, zazwyczaj budzi, a przynajmniej powinno budzić, zainteresowanie osób, których dane są lub będą agregowane i dalej przetwarzane. Dane dotyczące zdarzeń medycznych bez wątpienia do takich danych wrażliwych należą. A osobami uwzględnianymi przez system będziemy my wszyscy. Standardy przetwarzania danych opierają się m.in. na zasadzie ograniczenia celu przetwarzania. W świetle prawa dane muszą być zbierane w konkretnych, wyrażanych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W związku z tym mam pytanie: W jakim celu będą zbierane dane dotyczące (Dzwonek) zdarzeń medycznych, w tym dane o ciąży? Wysoka Izbo! Kobiety w Polsce traktowane są bardzo przedmiotowo i nie mają prawa decydować same o sobie, są dyskryminowane, nie mogą dokonywać same wyborów dotyczących ich ciała i życia. Dlatego każdy nowy pomysł, który się pojawia, każda inicjatywa rządowa od razu budzi podejrzenia. Po co jest rejestr ciąż? Gdzie jest drugie dno? Po co? Statystyki to są dane wyjątkowo wrażliwe. Zbieranie informacji o kobiecie i jej stanie, ciąży, jest niebezpieczne i wbrew konstytucji i RODO. To są dane wyjątkowo wrażliwe, raz jeszcze powtarzam. W naszym prawie nie ma takiej sytuacji, żeby można było się uchronić przed inwigilacją. To jest kolejna inwigilacja społeczeństwa, kolejny rejestr, który może wyłapywać kolejne ofiary dla Ziobry.

Wysoka Izbo! Mam kilka pytań do pana, panie ministrze, jak i do opozycji, której rozum przysłania ideologia w tej dyskusji, to widać jak na dłoni. Panie ministrze, po pierwsze, czy te zapisy, o których mówimy, to jest ewenement w skali Europy, czy one też obowiązują w Holandii, będą obowiązywać w Holandii, w Niemczech i we Francji?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata o tzw. rejestrze ciąż jest tak naprawdę debatą o tym, na ile Polki mogą ufać państwu polskiemu i jego instytucjom; na ile mogą ufać, że państwo chce chronić ich zdrowie i życie, a nie przejąć totalną kontrolę nad ich ciałem; na ile mogą ufać, że zajście w ciążę lub wizyta u lekarza nie skończą się w przypadku poronienia wizytą prokuratora. Niestety odpowiedź na to pytanie jest jedna. Państwu pod rządami Zjednoczonej Prawicy Polki nie mogą w żadnym względzie ufać. To zaufanie zostało pogrzebane przez PiS w październiku 2020 r., kiedy na polityczne zlecenie tzw. trybunału Przyłębskiej wprowadzono niemalże całkowity zakaz przerywania ciąży. A teraz chcecie gnębić kobiety rejestrem ciąż.

Wysoka Izbo! Nie dajmy tych informacji do lekarza. Państwo tego nie chcecie. Weźmiecie odpowiedzialność za tę śmierć? Weźmiecie za to odpowiedzialność? Dobrze tylko pokrzyczeć z tej mównicy. Panie Marszałku! XXI w. System elektroniczny ma ratować życie ludzkie, ułatwiać ratowanie tego życia. Mam takie pytanie: Z jednej strony - kto ma dostęp do tych informacji oprócz zespołu medycznego? A z drugiej strony - może utworzymy rejestr odlotów intelektualnych i kłamstw opozycji? Pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Oczywiste jest, że rząd PiS boi się kobiet. bo odkąd rządzi, utrudniacie im życie i pozbawiacie je wielu praw, o których tu już dzisiaj była mowa. Teraz wykorzystujecie zalecenia Komisji Europejskiej i dajecie dostęp do dokumentacji medycznej prokuratorowi Ziobrze. Po co? Prokurator Ziobro udowodnił nie raz, że nie powinien mieć żadnego dostępu do danych niejawnych, bo sam stanowi zagrożenie. Dlaczego kłamiecie, że rozporządzenie w obecnym kształcie wynika z zaleceń Komisji Europejskiej, w których nic nie ma o konieczności udostępniania dokumentacji medycznej prokuratorom? Dlaczego tę zmianę wprowadzacie rozporządzeniem, a nie ustawą?

Pani poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Dulszczyzna to właśnie ukrywanie informacji o tym, że kobieta jest w ciąży, a poza tym panie ubezwłasnowolniłyście mężczyzn, bo oni nie mają nic do powiedzenia na temat poczęcia.

Jest to informacja, która w tej chwili jest w systemie e-informacji, jaką posiada podstawowa opieka zdrowotna i nie tylko podstawowa opieka zdrowotna. Wiedza na temat ciąży dotyczy pewnych ryzyk w ocenie potrzeby leczenia i stosowania leków, gdyż większość leków praktycznie ma przeciwskazanie do stosowania w ciąży. Pytanie do pana ministra: Jakie informacje o ciąży będą przekazywane do Systemu Informacji Medycznej? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z majowego badania Ipsosu wynika, że 66% Polek i Polaków jest za prawem kobiet do przerywania ciąży do 12. tygodnia. 66%, czyli 7 na 10 osób w Polsce, jest za. W związku z tym nie będę do państwa apelowała. Nie będę pytała, czy w antykobiecym państwie rejestr ciąż czy - jak mówicie - System Informacji Medycznej może powodować nadużycia, bo to jest oczywiste, że może. Zaapeluję do kobiet, żeby zachowały spokój. W świetle obowiązującego w Polsce prawa za własne aborcje kobiety nie mogą być karane. Niezależnie więc od zagrożeń, jakie przynoszą kolejne projekty Prawa i Sprawiedliwości, większość Polaków jest za zmianą tego antykobiecego prawa. Pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość. W ramach wieloetapowej procedury stanowienia prawa przewidziano instytucję komisji prawniczej, która funkcjonuje w ramach Rządowego Centrum Legislacji, która ma charakter pomocniczy. To przede wszystkim weryfikacja pod kątem poprawności struktury aktu względem ˝Zasad techniki prawodawczej˝ itd. Dlaczego rozporządzenie, o którym dzisiaj dyskutujemy, panie ministrze, zostało zwolnione z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą?

A swoją drogą to jest to zgroza, kiedy słyszę dyskusję kobiet z opozycji, które w każdych warunkach, w każdej sytuacji domagają się takich przepisów prawa, które pozwalają matkom mordować własne dzieci. To jest po prostu zgroza. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dewotki i dewoci polityczni zgotowali polskim kobietom piekło. W Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Ukrainie, Bułgarii, na Słowacji, we Włoszech, Szwecji, Norwegii, Hiszpani, Niderlandach, Finlandii, Rumunii, Chorwacji, Danii, Grecji, Belgii, na Litwie, Łotwie, w Szwajcarii aborcja jest legalna i bezpieczna.

Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, mam do pana prośbę, aby pan jeszcze raz wytłumaczył paniom siedzącym po tej stronie, że to nie jest rejestr ciąż, że jest to System Informacji Medycznej, który funkcjonuje od dawna, zawierający dane, które są niezbędne do ratowania życia i zdrowia kobiet, jak również dzieci. Bardzo mi przykro, że panie traktujecie kobiety przedmiotowo i że mówiąc o zdrowiu kobiet, zdrowiu dziecka, mówicie tylko o aborcji i o tabletce ˝dzień po˝ Czy prawdą jest, że obecny rząd wprowadził standard opieki okołoporodowej, gdzie określamy wiele świadczeń należnych kobietom, m.in. wsparcie psychologiczne?

Panie Ministrze! Cóż takiego się stało w naszym kraju, że w tym momencie wprowadzacie tzw. rejestr ciąż? Dla państwa to jest śmieszne, ale dla obywateli nie. A więc trzeba to wszystko przykryć. Co się robi? Wprowadza się rejestr ciąż.

Szanowni Państwo! Pani poseł Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo trudno przysłuchiwać się tej dyskusji. Sprowadziliście ją państwo do jednego: do aborcji. Tabletka po˝ - to jest dla was najważniejsze.

Gdyby nie moja wielka wiara i doświadczenie wyniesione z mojego domu rodzinnego, nie byłoby mojej pierwszej córki. Zapamiętajcie to sobie. I nie doprowadzajcie do takich stanów młodych kobiet. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Chciałbym zapytać pana ministra, czy dane wrażliwe dotyczące rejestru ciąż i stanu zdrowia milionów kobiet w Polsce będą gromadzone zgodnie z dyrektywą o ochronie danych osobowych wydaną przez Unię Europejską. Chciałbym przypomnieć, że w przypadku gdy dane te będą gromadzone wbrew woli zainteresowanego i zostaną zapisane w tym rejestrze, to prawo unijne nakłada na administratora takiego systemu obowiązek ich usunięcia na wniosek osoby, której te informacje dotyczą. W każdym innym przypadku na instytucje gromadzące te dane będą nakładane milionowe kary. Chciałbym zapytać pana ministra, czy Polska jest przygotowana w związku z tym na taką ewentualność. Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Panie Ministrze! Podpisano rozporządzenie, które zgodnie z zapewnieniem ma wpłynąć na polepszenie stanu zdrowia kobiet. Tworzy się kolejny rejestr danych wrażliwych, który, jak się zapewnia, nie jest rejestrem związanym z systemem karnym, sądowym, skarbowym czy też policyjnym. Czy pan, panie ministrze, jest przekonany, że dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia milionów kobiet w Polsce będą gromadzone zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej? Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią Anitę Kucharską-Dziedzic. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Jestem zbudowana dzisiejszą dyskusją, zwłaszcza tym, że po jednej i po drugiej stronie sali plenarnej wszyscy się powoływaliśmy na standardy europejskie. To jest coś, co może nas rzeczywiście połączyć. Przypominam, że standardy europejskie to przy opiece nad ciężarną wizyty w domach położnej, a nie dzielnicowego.

Przypominam, że standardy europejskie to także właśnie ta nieszczęsna aborcja do 12. tygodnia ciąży, to in vitro i wszystkie inne kwestie, które są ważne dla zdrowia reprodukcyjnego kobiet, a które w Polsce są pomijane, zakłamywane, przemilczane i kobietom odbierane.

Wanda Nowicka jest na sali. Przypominam, że działania Parlamentarnej Grupy Kobiet wasza koleżanka z Prawa i Sprawiedliwości zablokowała i grupa nie zebrała się ani razu. Przypominam także państwu, że standardem europejskim jest godność i podmiotowość człowieka. Człowieka - kobiety i mężczyzny. I pewnie nie byłoby dzisiaj tej dyskusji, gdybyście państwo, planując stworzenie rejestru, whatever jak go nazwiemy, uwzględnili godność i podmiotowość kobiet i ich prawo do podejmowania decyzji, czy chcą, by w owym rejestrze znalazła się informacja o ich ciąży. Jeżeli to będzie decyzja na życzenie, to będziemy naprawdę ukontentowani tym, jak panie chcecie przywracania standardów europejskich w opiece zdrowotnej nad kobietą w Polsce. Pani poseł Daria Gosek-Popiołek. Pan minister twierdzi, że dostęp do tych danych o ciąży kobiety będą mieć jedynie pracownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, ratownicy. Ale nie jest to prawdą. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego dostęp do tej dokumentacji ma również prokurator. I to, co zmienia to rozporządzenie, jest fundamentalne, bo będzie to teraz możliwe na bardzo szeroką skalę. Obawy związane z tą właśnie skalą były zgłaszane już na poziomie konsultacji przez organizacje pozarządowe, proponujące bezpieczniki do tego rozporządzenia, ale zostały one całkowicie zignorowane. Więc te wszystkie obawy podnoszone przez nas są absolutnie uzasadnione. A teraz proszę panią poseł Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Panie Ministrze! Czy państwo się słyszą? Stajecie tutaj i mówicie, że chcecie dać dostęp do informacji o ciąży Polek Zbigniewowi Ziobrze, żeby dbać o ich zdrowie. Zbigniew Ziobro ma dbać o zdrowie Polek w ciąży. To przypomnijmy, jak dbacie o zdrowie Polek. Pani Izabela z Pszczyny, pani Agnieszka z Częstochowy, pani Anna ze Świdnicy. Tak dbaliście państwo o zdrowie Polek, o zdrowie tych kobiet, że tych kobiet, tych matek nie ma dzisiaj już z nami. Takie skutki ma zakaz aborcji, który wprowadziliście decyzjami politycznymi. Lewica jest po to, żeby powiedzieć: Ani jednej więcej. Lewica jest po to, żeby uspokoić kobiety, które boją się waszego rejestru ciąż. Pamiętajcie: przerwanie ciąży przez kobietę nie jest w Polsce karalne. Nie jesteście same, nie będziecie same. A już za 2 tygodnie - głosowanie w sprawie legalnej aborcji bez kompromisów. Proszę teraz o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Waldemara Kraskę. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z wielką uwagą przysłuchiwałem się dyskusji, jaka przetoczyła się dzisiaj przez salę obrad polskiego Sejmu.

Państwo dzisiaj wielokrotnie, pewnie dziesiątki razy mówiliście o rejestrze ciąż. To jest ewidentne kłamstwo. Powtórzę to jeszcze trzeci raz: nie tworzymy żadnego rejestru ciąż. Państwo to kłamstwo powtarzacie wielokrotnie, aby przestraszyć polski naród, polskie kobiety. Na takich samych zasadach jak do tej pory miał dostęp do dokumentacji medycznej. Proszę państwa, w tej chwili dane, które są w systemie informacji medycznej, czyli także te dotyczące wizyty kobiety u lekarza ginekologa, u lekarza położnika, odnotowanie, że jest w ciąży.

Grupa krwi, czy jest w ciąży czy nie, czy jest uczulona, czy ma w sobie jakiś implant - to są kluczowe informacje, którymi ja jako lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego będę się posługiwał. I muszę mieć do tego szybki dostęp. W stanie zagrożenia życia i zdrowia tego czasu nie mamy. Państwo mówicie tutaj naprawdę kłamstwa. Jeszcze raz powtórzę: Izba, jaką jest Sejm, nie jest miejscem, aby wprowadzać Polaków w błąd.

Mówiliście państwo o sądach, o prokuraturze. Ten dostęp do informacji medycznej jest taki sam jak był do tej pory. Proszę państwa, nie kłamcie, nie mówcie Polakom nieprawdy. Ten dostęp jest na tych samych zasadach co do tej pory. Proszę państwa, wprowadzamy ten rejestr, który będzie dostępny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale za kilka miesięcy tak się stanie we wszystkich krajach. To także jest dla bezpieczeństwa Polaków, Polek, które wyjeżdżają za granicę, niekoniecznie na wakacje, na wczasy, bo wyjeżdżają np. do pracy, wyjeżdżają w innych celach.

Państwo tego odmawiacie Polakom. Wiemy, proszę państwa, że wiele leków, które są przepisywane przez lekarzy, nie może być stosowanych u kobiet w ciąży.

Już od wielu, wielu lat mamy elektroniczną receptę i jak do tej pory żadne dane nie wyciekły, więc, proszę państwa, ten system jest dobrze chroniony.

Bardzo proszę państwa posłów o zajmowanie miejsc. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2312 i 2337. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków, - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2338 i 2336. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 2334. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Szanowni państwo posłowie, czy mogę prosić, wzorem poprzedniego dnia, o obniżenie. Bardzo proszę państwa posłów o zajmowanie miejsc.

Witamy razem z opiekunami. Bardzo proszę, panie premierze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Powiem o inflacji. Szanowni państwo, Polska przeżywa festiwal solidarności po raz drugi. O Polsce dawno nie mówiono tak dobrze, i to we wszystkich językach świata.

I rzeczywiście za to wszystko, przede wszystkim za wspaniałe przyjęcie Ukraińców w Polsce, chciałbym w pas się pokłonić naszym rodakom. Dziękujemy wszystkim naszym rodakom. Nad Polską zawisła czarna, ruska chmura. Dzisiaj, Wysoka Izbo, jest taki czas, że musimy ze sobą jak najbliżej współpracować, także przy tym bardzo ważnym głosowaniu, które jest przed nami. Potrzebujemy tej jedności. Dzisiaj można powiedzieć, że Polska jest na ustach całego świata. Rzeczywiście, jak rozmawiam z przywódcami z całego świata, to tak właśnie jest. Mógłbym ten pierwszy punkt podsumować swoimi słowami, ale podsumuję go słowami pana przewodniczącego Schetyny: Polska jest na pierwszej linii frontu w pomocy humanitarnej, Polska jest na pierwszej linii polityki i Polska jest na pierwszej linii w staraniu o sankcje. Dziękujemy, panie przewodniczący. Szanowni Państwo! Otóż jest to program, który po pandemii ma pomóc krajom członkowskim wyjść z zapaści gospodarczej. Pamiętamy te recesje, które były wszędzie, pamiętamy kłopoty na rynkach pracy. My sobie z tym inaczej poradziliśmy, ale tego było bardzo dużo w Europie. Co jest dzisiaj Polsce najbardziej potrzebne?

Polsce potrzebna jest promocja eksportu, Polsce potrzebne są oszczędności - i wszystkie te elementy zabezpiecza również krajowy program odbudowy. A więc mamy program, który na ten czas jest niezbędny, i dlatego głosowanie za nim uważam za bardzo ważne.

Szanowni Państwo! Po długich rozmowach, zbyt długo trwających, blisko rok, bo już rok temu powinny być one zamknięte. Dyskutowaliśmy o różnych kwestiach związanych z krajowym programem odbudowy, za chwilę jeszcze o tym powiem. Ale najwięcej czasu, właściwie 100% czasu, prawie 100% czasu poświęciliśmy tzw. reformie wymiaru sprawiedliwości, którą i tak planowaliśmy od dłuższego czasu. Tak zwanej z punktu widzenia Unii Europejskiej i problemów z tzw. praworządnością. Otóż, szanowni państwo, tak, w Polsce są problemy z praworządnością, ale właśnie ze względu na to, że nie ma równego traktowania obywateli przez sądy, także dzisiaj. Dlatego jest potrzebna reforma. A przede wszystkim praworządności nie było w czasach waszych rządów. Czy pamiętacie regułę Neumanna? Sąd zasądzi tak, jak Platforma sobie życzy. Albo pamiętacie regułę Milewskiego? Będzie sądził ten sędzia, którego wybierze ktoś z kancelarii premiera. Albo regułę Pietrzkowskiego? Nie mówiąc już o strzelaniu do górników albo o brutalnej akcji ˝Widelec˝ Taka była praworządność w waszych czasach. Ale, szanowni państwo, my nie ustępujemy przed Komisją Europejską. My wypracowujemy to, co i tak zamierzaliśmy zrobić, m.in. zmiany w Izbie Dyscyplinarnej. My nie jesteśmy traktowani przez Unię Europejską tak, jak do tej pory, do waszych rządów, dawniej to bywało, czyli jak niepiękna panna na wydaniu albo gorzej, jak Rafał Trzaskowski traktuje kobiety. My jesteśmy. Nie, tu proszę nie klaskać, to naprawdę nie ma tutaj. Należy się tylko nad tym ze smutkiem pochylić. My, szanowni państwo, jesteśmy dumnym krajem, dlatego negocjowaliśmy jak równy z równym.

Mogę też powiedzieć, że rzeczywiście to trwało miesiącami, to była mitręga, mnóstwo dokumentów. Czasami się zastanawiam, po co tyle tych dokumentów jest tworzonych.

Otóż są tam urzędnicy tacy jak Donald Tusk, którzy brali ogromne pieniądze - ogromne pieniądze - za to, że był wróg w Brukseli. Tak. I, szanowni państwo, właśnie za co on brał te pieniądze? Ja wiem, że was boli i dręczy. Szanowni państwo, ja wiem, że was boli i dręczy to, że ja zostawiłem za sobą złote trony i 100 albo więcej milionów złotych. Zostawiłem to wszystko dla służby publicznej. A wasz lider zostawił zaszczytną funkcję premiera dla kasy w Brukseli i pojechał do Brukseli. Zostawił was, przyczynił się do waszej klęski. Szanowni Państwo! Otóż tak: sam namawiam od dłuższego czasu, nakłaniam Polaków nie od wczoraj, nakłaniam od wielu miesięcy, od wielu lat, do tego, aby inwestować, aby kupować polskie obligacje. Namawiam do tego Polaków, ponieważ jest to inwestycja transparentna, bezpieczna dla wszystkich i propaństwowa. Jeśli sam robię to, do czego namawiam, to chyba dobrze, jeśli za moimi słowami idą czyny. Czyż nie tak? Gdybym tego nie zrobił, jestem przekonany, że krzyczelibyście, że trzymam pieniądze na depozytach i lokatach w tych strasznych bankach. Tak to już z wami jest, przyzwyczaiłem się do tego. Jeszcze jedno, szanowni państwo. Chciałbym też powiedzieć, ponieważ widzę tutaj zainteresowanie z tej strony sali, że mniej więcej 10 do 30 tys. zł średnio miesięcznie przeznaczam na różne działania charytatywne (Oklaski), na wspieranie różnych domów dziecka, na wspieranie warsztatów terapii zajęciowej, na kolonie, na wyjazdy dzieci w różne miejsca w Polsce i na Litwę, wspieram także osoby z niepełnosprawnościami. i od niedawna otaczam opieką również kilkanaście rodzin z Ukrainy po to, żeby się jak najszybciej zasymilowały w Polsce. Ale wracam do KPO po tej krótkiej dygresji. Otóż KPO, szanowni państwo, to jest program dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zawiera on kamienie milowe, wskaźniki w liczbie dla całej Unii Europejskiej ok. 5200. Włosi mają ich ponad 500, Rumunia ma ponad 500 tych wskaźników, tych kamieni, Rumunia ponad... przepraszam, Hiszpania - ponad 400, cztery razy mniejsza od nas Portugalia - ponad 300. My mamy 283. Ogromna większość tych kamieni milowych jest i tak ujęta w już istniejących dyrektywach albo tych, które są procedowane. Ogromna większość z nich służy naszym interesom, jest w naszym interesie, jest dla nas dobra lub neutralna. Śmiem twierdzić, że z wyjątkiem tych, które twardo negocjowaliśmy, które są związane z reformą wymiaru sprawiedliwości, po prostu wszystkie. Za chwilę powiem o tych fake newsach, na których się koncentrujecie, bo dzisiaj jest ważne głosowanie. Dzisiaj jest ważne głosowanie, szanowni państwo, drodzy rodacy, w przypadku którego Platforma Obywatelska chce głosować przeciw krajowemu programowi odbudowy, przeciw pieniądzom dla Polaków. Przynajmniej, drodzy rodacy, będziemy wiedzieli, komu trzeba podziękować za to, że te pieniądze cały czas do nas nie docierają, za to, że jest jakaś zwłoka. Nie wiem tego dokładnie. Liczę na to, że będzie to na przełomie tego i przyszłego roku. Też rzeczywiście na to liczę. To są ważne środki w wychodzeniu z kryzysu. Ale, drodzy rodacy, patrzcie na to, co mówi Platforma Obywatelska i opozycja na rożnych forach międzynarodowych, w tych europejskich trybunałach i na mównicach. Dzisiaj chcą zakrzyczeć to, że będą głosować przeciwko krajowemu programowi odbudowy. To wielki błąd. To jest wielki błąd, który mógłby bardzo dużo Polskę kosztować. Szanowni Państwo!

To nie jest żart, to jest rzeczywiście wstyd. To jest rzeczywiście skandal.

I że on jest dobrej myśli, że będą kolejne warunki narzucane przez Komisję Europejską. Niesamowite. Czy wy to rozumiecie? Szanowni państwo, jak słyszę takie rzeczy, to się zastanawiam, czy to jest jeszcze polska opozycja, czy to jest opozycja wobec Polski.

Czy Polsce służy traktowanie projektu Nord Stream 2 jak projektu biznesowego, czy służy Polsce raczej budowanie gazociągu do Norwegii, bałtyckiego gazociągu? Czy Polsce służy budowanie zapory na granicy z Białorusią, aby nie było prowokacji ze strony Łukaszenki i Putina, czy służy bieganie z reklamówką, obrażanie funkcjonariuszy i opowiadanie, że wpuścimy tutaj wszystkich? Wy mówiliście: Co powie na to Rosja? Tak się należy zastanawiać. I niech sobie wszyscy na to dzisiaj odpowiedzą. Szanowni Państwo! Trzeci punkt: inflacja. Inflacja jest dzisiaj problemem na całym świecie. Mamy jednego przeciwnika.

Zadziałała. Jak był kryzys, jak były początki kryzysu inflacyjnego, wdrożyliśmy tarczę inflacyjną, która częściowo również zadziałała.

Potrzebujemy konfiskaty majątków oligarchów rosyjskich, Federacji Rosyjskiej, tego, czego nie chcecie poprzeć. W tych działaniach antyinflacyjnych kluczowa jest także wiarygodność, bo polityka musi polegać na dotrzymywaniu umów.

Po pierwsze, obiecaliśmy zerowy VAT na żywność, co jest działaniem także zapobiegającym skutkom inflacji, bo zostawia pieniądze w kieszeniach Polaków. Obiecaliśmy trzynastą i czternastą emeryturę. Zrobione.

Dopłaty do nawozów - zrobione. Do 8%, bez zgody Unii Europejskiej. Obniżka VAT-u i akcyzy na energię elektryczną, na ciepło, na paliwo, na węgiel - to wszystko zrobione. To jest wiarygodność. To jest dotrzymywanie umów. A po waszej stronie? Miały być oszczędności, a wyszedł zabór OFE. I jeszcze Tusk niedawno mówił, że zrobiłby to samo. Zabierze drugą część OFE. Tak, skandal. Miała być, szanowni państwo, dobra polityka senioralna, a wyszła podwyżka wieku emerytalnego. Podniesienie ZUS-u w ich czasach - o tym zapominamy. Otóż rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, z 13% na 6%. To są nasze działania, które mają zapobiegać skutkom inflacji. To są nasze działania antyinflacyjne. Walczymy z inflacją tak, jak walczy cała Europa. Jest to jasne dla wszystkich, że inflacja jest dzisiaj wielkim problemem. Wielkim społecznym i gospodarczym problemem dla wszystkich rodzin. nie tylko w Polsce. Wie o tym prezydent Biden, prezydent Macron, premier Johnson, kanclerz Scholz, premier Republiki Czeskiej, prezydent Litwy, tylko jakoś Platforma Obywatelska nie wie o tym, bo tu.

To próbują zrobić.

Szanowni Państwo! Ale też w takim czasie jak ten prócz walki z inflacją... tu przejdę do ostatniego punktu, do czwartego punktu. Czwarty punkt to jest to, co chcemy zrobić, aby złagodzić ból Polaków związany z wysokimi cenami węgla, z wysokimi cenami paliw. Otóż, po pierwsze, prowadzimy program zakupu węgla i zwiększenia wydobycia węgla w polskich kopalniach (Oklaski) bo, owszem, Polska jest w awangardzie organizacji procesu sankcji na Rosję po to, żeby skutecznie walczyć o suwerenność Ukrainy. To jest potrzebne, ale to, zdajemy sobie z tego sprawę, dotyczy bardzo mocno polskich rodzin.

Pracujemy dzisiaj nie tylko nad zakupami, ale także nad mechanizmami dystrybucji, po to żeby ominąć łańcuszek pośredników, po to żeby nie zarabiali na tym pośrednictwie, tak żeby po prostu Polacy mieli jak najtańszy węgiel. Trzecia.

Dlatego powiem o tym, co już zrobiliśmy. Obniżenie VAT na paliwo kosztem ok. 7 mld zł dla budżetu - a wy się dziwicie, że ciągle ten budżet daje sobie radę, prawda?

Ale tak, paliwo cały czas jest za drogie. Będziemy starali się robić wszystko, aby było jak najtańsze, także poprzez umocnienie złotówki. A co umacnia złotówkę? Krajowy Plan Odbudowy umacnia złotówkę i nasza polityka fiskalna oraz nasza polityka regulacyjna umacniają złotówkę. To jest jedna, kompleksowa polityka makroekonomiczna - spójna, logiczna i dobra dla Polaków. Co jeszcze zrobiliśmy, szanowni państwo. aby ulżyć Polakom, aby zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków? Ok. 15 mld zł pozostanie w kieszeniach Polaków, i to po 18 mld, które od początku roku zostały w kieszeniach Polaków. Pewnie, że cały czas bolą te ceny w sklepach, bolą Polaków, ale pomyślcie, szanowni państwo, co byłoby, gdyby nie te proobywatelskie, prospołeczne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dalej, wśród różnych cen nośników energii bardzo ważne są ceny ciepła.

Bo rynek komercyjny to jedno, a działania społeczne to jest druga sprawa. I my zrobimy wszystko, aby ulżyć Polakom w tym zakresie.

Czy można zaufać takim ludziom, którzy mylili się w tych zasadniczych sprawach? Którzy uważali, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy, a rosyjscy inwestorzy, tak Tusk mówił, to są normalni inwestorzy i nie można ich traktować jako jakichś ideologicznych inwestorów? Albo jeszcze jeden cytat. Mówił, że mamy tutaj gaz z gazociągu jamalskiego i niepotrzebny jest nam ten gaz norweski. Gdzie byśmy byli dzisiaj, szanowni państwo? Można im miłosiernie wybaczyć, ale nie zaufać, drodzy rodacy. Czy rację mieliśmy my, budując tę zaporę z Białorusią, czy wy, którzy chcieliście wpuszczać? Czy rację miał prezes Jarosław Kaczyński, który mówił o tym, że Rosji nie można zaufać za żadne skarby (Oklaski), czy wy, którzy próbowaliście robić politykę razem z Rosją, a Niemców i niemiecką politykę nazywaliście, i to jeszcze niedawno, błogosławieństwem dla Europy? Ręce opadają, wstyd. Ale nic dziwnego, bo chcę jeszcze o jednej rzeczy przypomnieć.

Otóż on przyjmował bardzo wiele nagród, niemieckich nagród, z rąk Niemców, ale przyjął jedną szczególną, którą łatwo będzie zapamiętać wszystkim Polakom. To jest minister spraw zagranicznych, Niemiec, ten, który negocjował Rapallo.

A więc zapamiętajmy wszyscy. Szanowni Państwo! Dzisiaj na koniec chcę powiedzieć, że potrzebujemy współpracy, potrzebujemy walki, wspólnej, razem, aby zdusić inflację, aby walczyć o lepszy los Polaków. Dzisiaj nie potrzebujemy wroga wewnętrznego. Nie szukajcie wroga wewnętrznego, poproście wasze media, żeby nie szukały wroga wewnętrznego. gdzieś tam jakieś mównice europejskie okupować. Dla nas najważniejsze jest to, co się tutaj dzieje, tu, w Polsce, w Augustowie, w Krośnie, w Rzeszowie, w Gorzowie, wszędzie tutaj, właśnie w Polsce, w Gorlicach, nie mylić z Goerlitz. I dlatego, szanowni państwo, nie idźcie tą drogą. Wszyscy razem powinniśmy pracować na rzecz Rzeczypospolitej, na rzecz wyjścia z tego ogromnego kryzysu. Nie proponujcie swoich rozwiązań inflacyjnych, bo one prowadzą nas prostą drogą do inflacji jak w Turcji - dzisiaj 73,5%. Dzisiaj mamy jednego przeciwnika, jednego wroga, jest nim Kreml, jest nim straszna, straszliwa wojna na Ukrainie, którą Ruscy zaczęli. Jest wojna z rosyjskim reżimem. To wojna o to, żeby pokojowo zakończyć te straszne zmagania, ale utrzymać suwerenność Ukrainy. Pomagajcie Polsce i pomagajcie nam pomagać Ukrainie, a będzie dobrze.

Dziękuję bardzo. Proszę państwa.

To prawda, różnimy się między sobą. Nie, pan nie pozwala, oczywiście. Proszę państwa, czuję się zażenowana. Czuję się zażenowana wobec tej młodzieży, która siedzi na galerii i patrzy na polityków, którzy decydują o losach naszego państwa. Państwo uważacie, że wam wolno, a tej stronie nie wolno. Do wniosków formalnych zgłosili się posłowie. Proszę. A pani nie powinna krzyczeć z ławki, a inna posłanka nie powinna odwracać się tyłem, wtedy kiedy ktokolwiek z tej mównicy przemawia. Przypominam tylko.

Wysoki Sejmie! Zwracam się z wnioskiem o przerwę w celu zwołania Konwentu Seniorów i uzupełnienia porządku obrad o normalną debatę nad 280 zobowiązaniami, tzw. kamieniami milowymi, do których premier zobowiązał się w ramach kapitulacji przed Komisją Europejską. Dziękujemy, panie premierze, za wystąpienie - kompletnie nie na temat. Tu powinna się odbyć normalna debata, każdy klub powinien mieć prawo normalnie usłyszeć, co sprzedaliście, jak obiecywaliście, że będziecie wstawać z kolan, a zdecydowaliście się pełzać przed Brukselą. Wzrost cen ogrzewania, wzrost cen prądu, wzrost cen posiadania aut, zakazy wjazdów do centrów. Gdzie jest granica obrony suwerenności, której nie przekroczycie? Gdzie jest ta granica? Dlaczego boicie się normalnej debaty? Nieprawda, panie premierze? Dziękuje, panie pośle. Bardzo proszę, pan premier chce zabrać głos. Panie premierze, ale jeszcze chwilę. Panie premierze. Przepraszam bardzo. Proszę państwa, oprócz uczniów, których powitałam, są jeszcze uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza ze Strzyżowa oraz stypendyści gminy Boguchwała. Witamy.

Teraz się do tego czwartego też odniosę. Pierwsza kwestia, która jest często podnoszona, to jakobyśmy mieli nałożyć dodatkowe opłaty za korzystanie z dróg ekspresowych, druga - o opłatach na samochody, trzecia - o wieku emerytalnym i czwarta związana teraz z tym, co usłyszałem, o wjazdach do centrów miast. Zacznę może od tej pierwszej.

Budujemy drogi ekspresowe. za pieniądze i europejskie, i coraz więcej za pieniądze polskiego podatnika, dlatego na ciężarówki, tak jak jest to dzisiaj, będziemy również nakładali obowiązek uiszczania opłat na tych drogach ekspresowych, które znakomicie budujemy w ekspresowym tempie - dziękuję panu ministrowi Adamczykowi. Czy to źle? Chyba to dobrze? To punkt pierwszy. Punkt drugi to opłaty od samochodów. To jest kolejny fake news, nie mamy zamiaru nakładać żadnych opłat od samochodów.

Na samochód, który ma wysoką pojemność skokową silnika, jest wyższa akcyza. Jeżeli jest samochód niskoemisyjny albo elektryczny, to mamy dopłaty. Wy myślicie, że można tylko nakładać podatki, tak jak robiła Platforma Obywatelska. Nie, można zwalniać z podatku i w ten sposób promować czyste powietrze (Oklaski) i promować w sumie też innowacyjność, bo zależy nam na tym, żeby rzeczywiście rozwijał się ten sektor, rozwijał się ten przemysł, to jest nasz model rozwoju Polski. Punkt trzeci to wiek emerytalny, szczególnie forsowany przez opozycję. Z tej mównicy. Platforma Obywatelska i PSL podwyższyły wiek emerytalny: dla kobiet o 7 lat i dla mężczyzn o 2 lata, a dla rolników, dla kobiet - o 12 lat.

Oczywiście mamy historycznie niskie bezrobocie, nigdy nie było tak niskiego bezrobocia. Więc jeśli ktoś chce, to chociażby przez zerowy PIT dla emerytów zachęcamy do pracy dłużej tego, kto ma ochotę pracować. Bo my dajemy wybór, jesteśmy partią, która daje wolność, partią wolności.

Proszę bardzo, z wnioskiem formalnym. Proszę. Pani Marszałek! Wnoszę o przerwę, by pan premier mógł ochłonąć i przestać kłamać.

Chce pan porozmawiać o dokonaniach rządu? 14-procentowa inflacja - zrobione. Zielone światło dla mafii węglowej - zrobione, gigantyczny wzrost rat kredytów - zrobione, drastyczny wzrost cen żywności - zrobione, rekordowe zyski Orlenu - zrobione. To są wasze prawdziwe dokonania. Chce pan porozmawiać o prawdzie i solidarności? Dziś będziemy głosować nad poprawkami Senatu, które zbliżają nas do wypełnienia kamieni milowych, które pozwolą, by pieniądze europejskie przypłynęły do Polski. Proszę, pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Koalicja Polska.

Gdy premier poprosił o głos, myślałem, że chce przeprosić panią Agnieszkę z Pacanowa, naczelniczkę poczty, za to, że próbowaliście ją dyscyplinarnie zwolnić za mówienie prawdy. Ale co? Premier duby smalone bredzi z tej mównicy. Jako polityk mogę pana oceniać, ale jako lekarz muszę pana zdiagnozować: pan jest patologicznym kłamcą. Proszę o odroczenie obrad, dopóki premier Morawiecki nie podda się terapii. Nie ma dzisiaj głosowania nad KPO. Dzisiaj jest głosowanie nad praworządnością, nad pieniędzmi dla Polski, za Polską.

Nie, to są uwagi, które są absolutnie niedopuszczalne, panie przewodniczący, absolutnie. Sugerowanie czegoś takiego jest niedopuszczalne. Wam wolno, prawda? Wam wolno ubliżać, upokarzać.

Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Ten stek kłamstw, te manipulacje, które przed chwilą usłyszeliśmy, i te obelgi z pana strony wobec opozycji są najlepszym dowodem na waszą arogancję i pogardę dla ludzi. Gardzicie ludźmi. Bo jak to jest, że premier Rzeczypospolitej wychodzi na mównicę i kłamie? To jest pogarda. Ta pogarda zeszła na dół. Wasi aparatczycy, partyjniacy gardzą ludźmi, wyrzucają ich z pracy w Pacanowie, a pan tu wychodzi i opowiada te wszystkie kłamstwa. Dziękuję panu prezesowi za trafną diagnozę i w pełni ją podzielam, chociaż nie jestem lekarzem. Prosiłbym jeszcze, panie prezesie, o wypisanie recepty, która pomoże Polsce.

Kiedy pan poseł Kaczyński kazał panu premierowi przebiec maraton, on źle zrozumiał.

Sam sprzedał nieruchomości tylko po to, żeby uciec przed podatkiem z Nowego Ładu, który pan zafundował, a jedynymi osobami, które głosowały przeciwko Funduszowi Odbudowy, byli Ziobro, Kaleta, Kanthak, byli pana ministrowie. To są właśnie pana oszustwa.

To nie był żaden wniosek formalny.

Ostatni wniosek formalny. Wysoka Izbo!

2 lata temu na tej sali zdarzył się cud.

Byliśmy na tej sali zgodni, że trzeba stanąć po stronie ofiar przemocy domowej. Dzisiaj na tej sali znów możemy stanąć przed analogiczną sytuacją, analogicznym wyborem, i czekam na rewanż strony rządowej, która może poprzeć opozycyjny projekt ustawy, który staje po stronie ofiar przemocy seksualnej, a o gwałcie mówi, że to nie jest byle jaki (Dzwonek) występek, tylko zbrodnia.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2315? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie pośle, wniosek był nie o przerwę, tylko o przerwę, żeby zwołać Konwent, żeby pan premier. Nie ma warunku, panie pośle. Proszę bardzo, panie pośle, bez głosowania ogłaszam 2 minuty przerwy.

Przypominam, że jesteśmy w trakcie głosowania.

Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2315? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

451 - za, 2 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2278. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2278? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2277 i 2277-A) - trzecie czytanie. Proszę pana posła Piotra Babinetza o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2121. Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedzeniu w dniu 26 maja rozpatrzyła poprawkę i wnosi, aby Wysoki Sejm raczył tę poprawkę przyjąć. Ponadto przypominam, że na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu komisja rekomendowała Wysokiej Izbie, aby przyjąć nowelizację ustawy o tej instytucji, tak aby była to nowa instytucja: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Żeby otworzyła się na Ukrainę, na Gruzję, na Mołdawię i inne kraje, a szczególnie narody Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2277. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia również poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2277, wraz z przyjętą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ˝Polskie Koleje Państwowe˝ (druki nr 2204, 2280 i 2280-A) - trzecie czytanie. Proszę pana posła Jerzego Polaczka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Wysoki Sejm oraz Komisja Infrastruktury procedowały nad rządowym projektem zmiany ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ˝Polskie Koleje Państwowe˝ Jest jedna poprawka.

Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2280? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ˝Polskie Koleje Państwowe˝ Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2245, 2279 i 2279-A) - trzecie czytanie. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo!

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2279. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 2. i 5. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 4. i 8. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Kto jest za przyjęciem 4. poprawki?

Sejm poprawkę przyjął. 5. poprawka jest bezprzedmiotowa. Kto jest za przyjęciem 8. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto jest za przyjęciem 10. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 12. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto jest za przyjęciem 14. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2279, wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (druki nr 2133, 2187 i 2187-A) - trzecie czytanie.

Dziękuję. Komisja przedstawia jednocześnie wniosek mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Kto jest za przyjęciem wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem 14. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad całością projektu ustawy z druku nr 2187. Kto jest za przyjęciem projektu ustawy w całości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Proszę pana posła Władysława Kurowskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!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 Sejm na 55. posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r., zgodnie z regulaminem, skierował ponownie projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu.

przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2246? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2260-A. Proszę pana posła Grzegorza Matusiaka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2205. Podczas drugiego czytania zgłoszono pięć poprawek. Komisja te poprawki odrzuciła. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2260. W dodatkowym sprawozdaniu przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem poprawki 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2260? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2283-A. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw w trakcie drugiego czytania, które odbyło się 8 czerwca, zostały złożone trzy poprawki. Ustawa została ponownie skierowana do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W dniu dzisiejszym połączone komisje rozpatrywały przedstawione poprawki.

Połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie odrzucenie tej poprawki i co oczywiste, głosowanie nad całością projektu.

Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2283? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2311. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość wniosków mniejszości 4. i 5. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest za przyjęciem 9. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 10. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 11. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 13. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 14. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 15. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 16. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest za przyjęciem 17. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest za przyjęciem 18. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 19. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 20. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2318-A. Proszę pana posła Marcina Porzucka o przestawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje głosowanie przeciw wszystkim dziewięciu poprawkom. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2318. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 2. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 3. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 7. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 6. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 7. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2318? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2316. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Sejm podjął decyzję o przystąpieniu do trzeciego czytania bez ponownego kierowania projektu ustawy do komisji. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu ustawy. W przypadku jego odrzucenia przystąpimy do głosowania nad całością projektu ustawy. Głosujemy nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy z druku nr 2316? Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2316? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2309 i 2312) Proszę pana posła Krzysztofa Lipca o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pragnę poinformować, że w dniu wczorajszym komisja rozpatrzyła 29 poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo. Chciałam przywitać gości z województwa lubuskiego. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Kto jest za odrzuceniem 4. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest za odrzuceniem 17. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 18. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2333 i 2337) Proszę panią poseł Gabrielę Masłowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem Sejmu skierowała w dniu 9 czerwca uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 - za, przeciw - 440, 1 się wstrzymał. Sejm poprawkę przyjął. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za odrzuceniem 3. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy.

Sejm poprawki przyjął. Kto jest za odrzuceniem 13. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za odrzuceniem 16. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

te krzyki? No i po co te krzyki?

Głosujemy. Kto jest za odrzuceniem poprawek 17. i 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 - za, przeciw - 451, nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawkę przyjął. Kto jest za odrzuceniem 20. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druki nr 2332 i 2338) Proszę pana posła Artura Szałabawkę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków, druk nr 2332, Senat zaproponował pięć poprawek.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest za odrzuceniem 4. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2331 i 2336) Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani marszałek Sejmu skierowała uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2331, do Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głosujemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Kto jest za odrzuceniem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Huberta Dominika Massalskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Niemirowicza-Szczytta z dnia 31 lipca 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Jacka Lisieckiego. Na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Jacka Lisieckiego. Na podstawie art. 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Jacka Lisieckiego. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Huberta Dominika Massalskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Niemirowicza-Szczytta z dnia 31 lipca 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Jacka Lisieckiego za czyn określony w tym wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Zieloni o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań, które zamierza podjąć Rada Ministrów w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które oddala wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Głosujemy nad wnioskiem w sprawie uzupełnienia porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy nad wnioskiem w sprawie uzupełnienia porządku dziennego o punkt obejmujący informację Prezesa Rady Ministrów na temat działań związanych z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw?

Prezydium Sejmu, na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Nikt się nie zgłasza. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 2334? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Proszę przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa panią Dagmarę Pawełczyk-Woicką o przedstawienie informacji. Bardzo panią proszę. Wysoki Sejmie! Powołanie Krajowej Rady Sądownictwa wynikało z ustaleń okrągłego stołu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa poszerzył zakres kompetencji rady m.in. o współdecydowanie o budżecie wymiaru sprawiedliwości. Do kompetencji rady przekazano także uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Zaowocowało to systematycznym wzrostem nakładów na sądownictwo powszechne. Rada jest strażnikiem niezależności sądów i niezawisłości sędziów - art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest także jedynym organem państwa uprawnionym do przedstawiania prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie na urząd sędziego, na wszystkie stanowiska sędziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa jest samodzielnym, centralnym organem państwowym, którego funkcje powiązane są z władzą sądowniczą. Krajowa Rada Sądownictwa wykonuje swoje zadania przy pomocy biura rady. Ustrój, zakres, działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Istotne zmiany dotyczące funkcjonowania i zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wprowadziła ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 17 stycznia 2018 r. Ustawą tą zmieniono sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów. Przedmiotowa ustawa przyznała możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa grupie co najmniej 2 tys. obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, mają pełna zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych, lub grupie co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ostateczny wybór przyznano zaś Sejmowi, który wybiera 15 sędziów spośród zgłoszonych kandydatów na wspólną 4-letnią kadencję. Wspólna kadencja dla członków rady, którzy są sędziami, została wprowadzona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. uznającym za niekonstytucyjne rozumienie kadencji członków rady wybranych spośród sędziów w ten sposób, że ma ona charakter indywidualny. Kwestia wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm stanowi źródło sporu politycznego.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ustrojodawca zasadnicze kwestie związane z funkcjonowaniem rady przekazał do regulacji ustawowej, pozostawiając w tekście konstytucji jedynie pewien minimalny standard konstytucyjności Krajowej Rady Sądownictwa. Zarówno na etapie prac nad tekstem konstytucji, jak i współcześnie sam fakt istnienia Krajowej Rady Sądownictwa umocowanej konstytucyjnie nie jest immanentnie wpisany w istnienie demokratycznego państwa prawa. Fakt bycia reprezentacją środowiska prawniczego wynika bowiem nie ze sposobu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale z tego, że z dużą przewagą wybierani są do jej składu sędziowie, co jest objęte gwarancją konstytucyjną.

Zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa członek rady potwierdza udział w innych niż posiedzenie plenarne pracach na rzecz rady złożeniem podpisu w karcie pracy i wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy. Po § 8 ust. 1 Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa dodano ust. 1a, w myśl którego członek Krajowej Rady Sądownictwa może brać udział maksymalnie w pracach dwóch komisji problemowych powołanych w radzie. W § 26a ust. 1 dokonano zmiany umożliwiającej komisjom rady odbywanie posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie w trybie obiegowym w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Uprzednio taki tryb pracy był dopuszczalny w przypadku rady, prezydium rady i zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa. Art. 179 konstytucji wskazuje, że Krajowa Rada Sądownictwa posiada wyłączną kompetencję do przedstawiania prezydentowi wniosków w sprawie powołania sędziów. Art. 186 ust. 2 konstytucji stanowi podstawę do występowania przez Krajową Radę Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy apelacyjne i wojskowe sądy okręgowe, w ramach prowadzonych przez nie postępowań. Proszę państwa, w dalszej części sprawozdania omówię te poszczególne kwestie, jak to wyglądało w 2021 r.

Rada wewnętrznie jest podzielona na komisje. Są to komisje stałe, co wynika z ustawy: Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, Komisja budżetowa, Komisja do spraw wizytacji i lustracji, Komisja do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych.

W skład Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wchodzi również członek wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa.

W dniu 30 listopada 2021 r. rada wskazała sędziego Jarosława Dudzicza jako swojego przedstawiciela w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dodam, że wygaśnięcie mandatu w radzie nie powoduje jednoczesnego wygaśnięcia tego mandatu. W skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. jako przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa powołano sędzię Katarzynę Chmur. Proszę państwa, w Krajowej Radzie Sądownictwa działa wspólna komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Krajowa Rada Sądownictwa odbyła 20 posiedzeń plenarnych w 2020 r., które trwały łącznie 77 dni. Rada rozpoznała 1792 zgłoszenia do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, administracyjnych oraz w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkich sądach administracyjnych, które pochodziły od 1713 osób, celem przedstawienia wyłonionych kandydatów prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie. Rada podjęła 1626 uchwał w sprawach indywidualnych, w tym 556 uchwał w przedmiocie przedstawienia prezydentowi wniosków o powołania na stanowiska sędziowskie i asesorskie.

Zespoły członków krajowej rady.

Jakby mogła pani w przeciągu 30 sekund podsumować, toby było bardzo, bardzo miło. Rok 2021 był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o działalność rady poprzedniej kadencji, właśnie w zakresie rozpoznania spraw indywidualnych konkursowych. Oprócz tego rada wydała 66 opinii o projektach aktów normatywnych i przedstawiła 18 stanowisk w sprawach dotyczących sądownictwa i sędziów. Rada podjęła 17 uchwał stwierdzających brak podstaw do podjęcia czynności wizytacyjno-lustracyjnych, wniosła odwołania czterech nieprawomocnych wyroków sądów dyscyplinarnych.

Bardzo dziękuję, panie marszałku. Bardzo proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie stanowiska komisji. Widziałem pana posła, widzę.

I też, panie profesorze, etyka. Wysoka Izbo!

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2022 r. zapoznała się z powyższą informacją oraz przeprowadziła dyskusję. Mnie pozostaje zrelacjonować, że dyskusja w dużej mierze miała merytoryczny charakter, co mnie cieszy.

Ze strony pani przewodniczącej padły odpowiedzi na pytania, a na te pytania, na które odpowiedzi nie padły, być może padną one w trakcie debaty sejmowej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie informacji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r., zawartej w druku 2115.

Myślę, że nie trzeba tego powtarzać. Chciałbym skupić się na tych działaniach związanych z posiedzeniami plenarnymi, o których pani przewodnicząca mówiła w ubiegłym roku. Tych posiedzeń było 20, a rok wcześniej było 16 posiedzeń. Rada rozpoznała 1792 zgłoszenia do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, a w poprzednim roku było ich 879, więc był to znaczny wzrost. Rada podjęła 1626 uchwał w sprawach indywidualnych, a rok wcześniej było to 920 uchwał.

Rada wydała również 66 opinii o projektach aktów wykonawczych i podjęła 17 uchwał stwierdzających brak podstaw do podjęcia czynności wizytacyjnych. Wniosła także odwołania do Sądu Najwyższego od czterech nieprawomocnych wyroków sądu dyscyplinarnego, sądu pierwszej instancji.

Myślę, że na szczególne podkreślenie zasługuje działalność rady na arenie międzynarodowej. Rada utrzymywała bieżące kontakty z innymi organizacjami międzynarodowymi, prowadziła dialog z Europejską Siecią Rad Sądownictwa. Brała udział.

W związku z tym myślę, że da pan sobie radę.

Rada utrzymywała kontakt ze sprawozdawcami komisji monitorignowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Spotykamy się dzisiaj na debacie, której tak naprawdę nie powinno być, bo rozmawiamy o sprawozdaniu organu widmo, organu, który de facto nie istnieje.

To jest pseudoinstytucja, która prześladuje polski wymiar sprawiedliwości, prześladuje demokrację. Niesie to ze sobą tylko kłopoty i szkody. Tę ocenę potwierdził niedawno Sąd Najwyższy, który uchwałą siedmiu sędziów orzekł, że Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana w tym trybie z 2017 r. nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym, którego skład został opisany w konstytucji, w art. 187.KRS-u nie ma. Jest za to neo-KRS, taka tandetna podróbka instytucji, którą niegdyś była. KRS została wyrzucona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa właśnie dlatego, że nie istnieje jako organ, który jest niezależny od polityków, i nikt poza Kaczyńskim i Ziobrą jej nie uznaje. Jednak jest to jedna z najdroższych podróbek w historii Polski.

W stosunku do 2020 r. zauważalny był znaczny wzrost pobranych diet, np. sędzia Styrna w 2020 r. pobrał z neo-KRS-u 68 tys., rok później już 169 tys. zł, czyli o 100 tys. zł więcej. Tyle samo otrzymał sędzia Mitera. Za ile dni pracy? Pani przewodnicząca mówiła - 77.

I to są dodatkowe pieniądze poza zasadniczą pensją. Rozumiecie państwo? Tak wygląda właśnie ta walka Jarosława Kaczyńskiego z tłustymi kotami. Te koty puchną z roku na rok, setki tysięcy złotych za taką polityczną wierność. Wstydu nie macie. Jakby tego było mało, te ciepłe posadki są także maszynką do szybkich, niesamowicie dziwnych awansów członków neo-KRS-u i ich rodzin.

Standardem powinno być nieubieganie się o awans w trakcie zasiadania w radzie, gdyż nad takim kandydatem muszą głosować jego koledzy z rady, a zatem działają nieobiektywnie. Zabiegają właśnie o własne awanse, aby zabezpieczyć sobie byt na przyszłość i mieć coś z tego, że poparło się niszczenie niezależności polskiego sądownictwa. Pani Dagmara Pawełczyk-Woicka - awans, Grzegorz Furmankiewicz - awans, Rafał Puchalski - awans, Dariusz Drajewicz - awans, Joanna Kołodziej - awans, Maciej Nawacki - awans, nawet podwójny, bo najpierw do sądu okręgowego, potem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wysoka Izbo! To jest sprawozdanie z działania organu, który uzurpuje sobie konstytucyjność, działa rozrzutnie. Sposób jego funkcjonowania naraża Polaków na blokadę środków z Krajowego Planu Odbudowy i kolejnego budżetu Unii Europejskiej. To sprawozdanie przyda się absolutnie do jednego - w trakcie postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej (Dzwonek) Ten papier nie zasługuje na rozpatrywanie przez Wysoką Izbę. Jest niepotrzebny, tak jak niepotrzebny jest neo-KRS. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ex iniuria non oritur ius, z bezprawia nie rodzi się prawo - mawiali Rzymianie. Nie znano jeszcze wtedy koncepcji państwa według PiS. Państwo PiS, zamiast strzec praworządności, strzeże swoich politycznych interesów - rządzącej formacji. W państwie bezprawia i niesprawiedliwości dobra zmiana może wszystko. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 186 przeczytamy, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Tymczasem neo-KRS nie jest organem niezależnym. Mianowani przez neo-KRS sędziowie zostali powołani w procedurze, która nie jest wolna od nacisków politycznych, nie dają więc rękojmi niezawisłości. Orzekły to już rok temu europejskie trybunały, orzekł to polski Sąd Najwyższy i mówiliśmy już o tym nie raz, i w tej Izbie, i podczas prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Neo-KRS nie jest organem niezależnym, nie gwarantuje obiektywnej i bezstronnej procedury wyborów sędziów i w konsekwencji dyskwalifikuje wszelkie sędziowskie nominacje do KRS. Jak co roku mamy tutaj omawiać informację z działalności Krajowej Rady Sądownictwa, tym razem za kolejny rok - 2021. Ale jak tu oceniać działalność tworu, którego zarówno powołanie, jak i funkcjonowanie stają w rażącej sprzeczności z konstytucją czy wręcz są złamaniem konstytucji i konstytucyjnych zasad: prawa obywatela do niezawisłego sądu, praworządnego i demokratycznego państwa prawa. Tworu, który w tej Izbie głosami państwa z prawej strony po raz kolejny został niedawno wybrany z naruszeniem konstytucji, a konkretnie art. 187 ust. 3. Po raz kolejny na kolejną kadencję wybrali państwo nową starą neo-KRS. W grzechu poczęta i reprodukowana neo-KRS produkuje owoce zatrutego drzewa - kolejne podważalne sędziowskie nominacje. Neo-KRS stała się kluczem dla autorytarnej władzy do przejęcia sądownictwa. Pycha - bo brak autorytetu i dorobku zawodowego nie jest tu wadą i nie przeszkadza z politycznego nadania wejść do neorady. Chciwość - podwójne diety za udział w posiedzeniach i komisjach, głównie zdalnych, stały się dla tej rady sprytnym sposobem na dorobienie. Nieczystość - grzech pierworodny nielegalnego przejęcia kontroli i upolitycznienia KRS przez obecną władzę. Łakomstwo - funkcje, awanse, finansowe frukty, dodatki mieszkaniowe i funkcyjne. Nepotyzm - intratne posady dla członków rodzin.

Lenistwo i znużenie - to, proszę państwa, grzech, który grozi nam wszystkim, obywatelom i obywatelkom, zmęczonym deformą polskiego wymiaru sprawiedliwości i demolką praworządności w naszym kraju. Rys historyczny, skład, lista kompetencji, wykaz komisji, formułki jak przepisane z podręcznika. Wszystko to, co można znaleźć w internetowej przeglądarce, jeśli to kogoś interesuje, wszystko, z czego nie wynika nic. Czy merytoryczna wartość i treść informacji odpowiadają jakości i ilości pracy, liczbie dni przepracowanych w tej radzie, przez tę radę? Cóż, jaki KRS, taka informacja i takie wystąpienie.

Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Dzisiaj mamy taką bardzo wymowną koincydencję. Głosowania przed niespełna 2 godzinami nad poprawkami Senatu, które miały na celu ratowanie praworządności w Polsce, pokazanie zarówno tu, w kraju, jak i na zewnątrz, że mamy wolę naprawienia praworządności. Niestety ten egzamin większość sejmowa oblała. Mam nadzieję, że jest świadoma konsekwencji dzisiaj, jutro i w kolejnych miesiącach czy latach swojej decyzji. Dzisiaj po niespełna 2 godzinach obradujemy nad sprawozdaniem Krajowej Rady Sądownictwa i na tym dzisiaj przede wszystkim się skupiamy. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, różnie oceniane, przeze mnie niezwykle krytycznie, były tym sztandarowym krokiem, etapem Zbigniewa Ziobry i jego reformy na drodze do naprawy wymiaru sprawiedliwości. Jak Zbigniew Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim dochodzili do władzy w 2015 r., zarzekali się, że te wszystkie elementy, zmiany w instytucjach wymiaru sprawiedliwości dadzą obywatelom wymiar sprawiedliwości sprawiedliwy, dostępny dla każdego obywatela, tańszy, działający w sposób przyjazny, dający gwarancję rozwiązania spraw obywatelom w sposób znacznie lepszy niż dotychczas. Dzisiaj, pani przewodnicząca, mija za chwilę 7 lat od czasu, kiedy też w sumie postać pani dosyć bliska, minister Ziobro wziął się do pracy. Dzisiaj w tym sprawozdaniu wypadałoby właśnie wykazać z ramienia Krajowej Rady Sądownictwa, co w kontekście 7-letniej działalności bliskiej pani politycznie osoby, jego obozu politycznego, tych kilkuset zmian legislacyjnych zrealizowano z tych obietnic, które państwo złożyliście. Terminy w sądach biją kolejne rekordy, rozpatrywanie kolejnych spraw budzi obawy, budzi niepokój Polaków. Mizernie działający wymiar sprawiedliwości ma swoje przełożenie również na życie gospodarcze Polski. Nie ma dynamicznie rozwijającej się gospodarki z kulejącym sądownictwem, to jedno z drugim się wyklucza. Zapewnialiście, że w tym względzie też będzie rewelacyjnie.

Zabrakło w tym wystąpieniu jakiegokolwiek dowodu na to, że te wielkie reformy, w których wprowadzaniu pani, chcąc nie chcąc, uczestniczyła, przyniosły jakikolwiek wymierny efekt. Ja powiem, pani przewodnicząca, że wiele osób dało się zwieść 7 lat temu tym hasłom, że będzie lepiej, że będzie sprawiedliwiej. Dzisiaj jasno o tym mówią. Bardzo często z tej mównicy przytaczam przykład pana Marka Kubali, jednego z tych, którzy tworzyli stowarzyszenie osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. On bardzo często pisze do mnie, jak rozmawiamy, to też wspomina: proszę przypomnieć moją sprawę, proszę przypomnieć, że zaufałem i Ziobro i jego sprzymierzeńcy mnie oszukali. 4 lata oczekiwania na rozpatrzenie skargi nadzwyczajnej.

Przed nami wreszcie będzie wielki problem, prędzej czy później, co z tym dorobkiem iluś lat funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa zrobić, bo państwo zmienicie, mam nadzieję, swoją lokalizację, jeśli chodzi o usytuowanie w Sejmie. Będzie wielki problem, jak to przywrócić na normalne tory, z wielkimi konsekwencjami dla Polski, bo to nie z PiS-owskiej kasy będą wypłacane odszkodowania za błędy w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, tylko państwo polskie będzie płaciło odszkodowania za wadliwie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. Ten całokształt - kończąc, panie marszałku - skłania nas do przyłączenia się do wniosku o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Sądownictwa za 2021 r. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, koło Konfederacja.

Szczęść Boże! - sędziom i podsądnym. Mam osobiste doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości, głębsze, można powiedzieć wielopokoleniowe tradycje sięgające jeszcze poprzednich reżimów. Sam stawałem przed sądami postpeerelowskimi w charakterze i podsądnego, i świadka, i jako obserwator, dokumentalista. Dokumentowałem, jak czyni się zadość niesprawiedliwości w tym resorcie, ponieważ to jest oczywiście bardzo smutny pejzaż, to jest tragiczny obraz. Właśnie ta chwila, ta debata, która powinna ogniskować uwagę opinii publicznej i angażować wielu parlamentarzystów, tu, przy pustawej sali, to już sprawa przebrzmiała. Wszyscy wiedzą, że i tak się nic nie zmieni, bo pozostaje zachowana podstawowa zasada ustrojowa w Rzeczypospolitej III i pół sformułowana, zdefiniowana i zdiagnozowana przez znakomitego pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Zasada ta brzmi: wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. I tej zasady trzymacie się wszyscy - i lewica z lewej, i lewica z prawej - i kopiecie się, ale nie powyżej kostek.

Gdzie był ten KRS, kiedy przez poprzednie 2 lata łamano prawo na wszystkich szczeblach i poziomach, kiedy pozbawiano Polaków ich praw konstytucyjnych, pozbawiano ich zdrowia, życia pod pretekstem walki z mniemaną pandemią? To jest rzeczywiście szopka, groteska, to jest tylko ewentualna przepychanka, wymienianie nie naszych i nielojalnych wobec naszej centrali partyjnej na naszych i nic się nie zmienia. Tu łamano prawo aż do zbrodni, a milczał KRS, który ma wiele do powiedzenia w innych sprawach, wtedy kiedy to jest w głównym nurcie, kiedy to jest poprawne politycznie. Oczywiście 40 już.

Można powiedzieć, że perfumujecie ten zbiornik nieczystości, wielopokoleniowe kadry sądownictwa postpeerelowskiego, nowe złogi, bo to się już wychowały nowe pokolenia. Przecież to są całe klany, żeby nie powiedzieć szajki sędziowskie, prokuratorskie, przerośnięte te złogi z nieprawością w różnych służbach i resortach.

Witam was, dzieci, witam was, wychowawcy, witam dziewczynki i chłopców. Cieszę się, że jesteście i patrzycie na naszą ciężką pracę. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Dlaczego krytycznie oceniła pani kilka dni temu uchwałę Sądu Najwyższego, który uważa, że KRS nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym? Czy według pani skład rady jest reprezentatywny? Jak wytłumaczyć częste roszady w Krajowej Radzie Sądownictwa? Liczyłem na to, że inaczej niż w poprzednich latach przedstawi pani informację o działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Po raz kolejny to ponad 100-stronicowa informacja, która powstała na zasadzie: kopiuj - wklej. Mówiłem już o tym na posiedzeniu komisji. Przyznam, że mile mnie pani zaskoczyła dzisiejszym mailem, bo zapowiedziała pani, że kopiowania w informacji w następnym roku raczej nie będzie. Nie odpowiedziała pani jednak ani przed sejmową komisją, ani w tym mailu do mnie na pytania, dlatego stawiam kolejne. Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła 1792 kandydatury na sędziów, przedstawiła prezydentowi 920 wniosków nominacyjnych, a odbyła jedynie 261 rozmów z kandydatami i dwie z wizytatorami. W orzeczeniach międzynarodowych trybunałów znajdują się krytyczne opinie o KRS. Dlaczego brak nawet pół zdania na ten temat w informacji dla Sejmu? Dlaczego stanowisko KRS w sprawach przed międzynarodowymi trybunałami jest zawsze zgodne ze stanowiskiem obozu rządzącego? Dlaczego ani słowa w tej informacji o sprawie Grzęda przeciwko Polsce? Przecież Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prawo do odbycia pełnej kadencji członka KRS znajduje oparcie w fakcie, że KRS jest organem przewidzianym w konstytucji do ochrony niezawisłości sądów i sędziów. Na stronie 102 czytamy: pomimo zawieszenia członkostwa KRS w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa prowadziła dialog. Pani sędzio, przecież KRS ostatecznie straciło status członka, bo uznano, że nie jest niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a przecież musi gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa. Przejrzałem wszystkie ubiegłoroczne opinie i stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa. Dlaczego niemal zabrania się sędziom udziału w akcjach społecznych, charytatywnych, a przykładowo nie ma żadnego zastrzeżenia, choćby w przypadku opinii na temat projektu ministerstwa dotyczącego resocjalizacji nieletnich. Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z konstytucją musi stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nie siedziała pani, siedział przewodniczący Styrna. Ale pytanie jest aktualne: Dlaczego Krajowa Rada Sądownictwa boi się stanąć w obronie wielu sędziów? Pani sędzio, solidarność - jedno z najpiękniejszych słów. Wystosowała pani pismo w obronie sędziów odsuniętych od pracy? Milczenie w tym przypadku nie jest złotem, jest wstydem. Bezduszność wyparła słowo: solidarność. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, do zadania pytań zapisało się 18 posłów. Czy ktoś jeszcze chciałby się zapisać? Zamykam listę.

Czytając niniejsze sprawozdanie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że najbardziej doniosłym osiągnięciem Krajowej Rady Sądownictwa w roku 2021, oczywiście poza trwaniem w swoim składzie i przekonywaniem Polaków, że nic się nie stało, była likwidacja rady bibliotecznej tej instytucji składającej się z pięciu osób, w tym czterech z tytułami doktorskimi. Poza tym w sprawozdaniu Krajowej Rady Sądownictwa mamy opis jej walki z pandemią. Ani słowa o kontrowersjach, które budzi rada swoim składem wśród sędziów, prawników i naukowców związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości oraz międzynarodowej społeczności. W zasadzie nie ma takiego pytania, na które można byłoby się spodziewać satysfakcjonującej odpowiedzi. Pozostaje więc jedynie życzyć radzie trwania w błogostanie, a Polakom życzyć szybkich i nieuniknionych zmian. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Przewodnicząca! Wiem, że 3 tygodnie na stanowisku to niewiele, ale chciałbym zapytać, czy podjęła pani problem organizacji pracy rady w kontekście tych diet, o których mówi Najwyższa Izba Kontroli, o których donoszą media, w wysokości blisko 2900 tys. zł. Wiceprzewodniczący rady otrzymał 244 tys. To blisko drugiej osoby w państwie, o 60 tys. więcej niż wicemarszałkowie Sejmu. Kolega wiceprzewodniczący, poseł Mularczyk, zarobił tyle, co szeregowi posłowie w całym roku. W związku z powyższym chciałbym zapytać, czy pani przewodnicząca chce to przeorganizować, aby było to bardziej przejrzyste. Druga kwestia dotyczy udziału KRS-u w pracach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Państwo w sprawozdaniu piszecie, że ta decyzja była bezprawna, niezgodna ze statutem tejże sieci. Wobec powyższego chciałbym zapytać, jakie działania, jakie kroki prawne podjęła nasza KRS, żeby udowodnić, że decyzja Europejskich Sieci Rad Sądownictwa dotycząca zawieszania KRS-u była bezprawna. Dziękuję. Pan poseł Rafał Adamczyk. Czy jest? Nie ma. Zapraszam. Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Europejski Trybunał Praw Człowieka i TSUE jednoznacznie orzekły, że upolityczniony neo-KRS jest organem niekonstytucyjnym i tak naprawdę po prostu nie istnieje. Nawet pani przewodniczącej tutaj nie ma. Eksperci są zgodni, że dopóki nie zlikwidujemy neo-KRS-u i nie powołamy go w konstytucyjnym trybie, dopóki wszyscy nominaci neo-KRS-u nie stracą swoich posad, a awansowani sędziowie nie wrócą na swoje poprzednie miejsca, absolutnie wszyscy, od osób powołanych na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, administracyjnych czy NSA, kończąc w Sądzie Najwyższym, dopóty nie będziemy mogli w Polsce mówić o przewróceniu praworządności. Nie możemy też mówić o przywróceniu praworządności dzisiaj po tym, jak odrzuciliście wszystkie poprawki Senatu dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. Polacy przez to cierpią i będą cierpieć dalej, bo pieniądze z Unii, które nam się należą, a nie wam, Polkom i Polakom, nie przypłyną (Dzwonek) Ale przyjdzie czas, że przywrócimy praworządność w Polsce. Odwrócimy wszystkie wasze złe ustawy. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Krystyna Skowrońska. Nie ma. Pani posłanka Wanda Nowicka, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Stąd te ogromne diety, stąd te ogromne uposażenia - bo takim ludziom po prostu trzeba słono zapłacić.

Piszecie w raporcie, że ta decyzja jest niezgodna ze statutem i nie wywołuje skutku prawnego.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! KRS to fundamentalny problem wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej 15 członków wybierali sędziowie spośród swojego grona. Co ciekawe, jednym z autorów takiego rozwiązania był sam Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w pracach podstolika ustrojowego w ramach okrągłego stołu. Przez wiele lat nie budziło to wątpliwości, aż do czasów dobrej zmiany. Polski wymiar sprawiedliwości cierpi na systemową dysfunkcję związaną z procesem nominacyjnym sędziów, którą trzeba naprawić. To musi być zmienione. Kiedy ten haniebny czas się skończy? Jeszcze tylko słowo o wyborach w Hiszpanii. To prawda, że członków naczelnej rady sądowniczej wybierają Kortezy, czyli parlament, ale sam wybór poprzedzony jest selekcją i oceną kandydatów dokonywaną wyłącznie przez sędziów. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Panie Marszałku! Neo-KRS - nielegalnie, niezgodnie z konstytucją powołany organ, organ widmo, ghost ship. Tylko że w legendach żeglarskich taki statek widomo to była kara boska, a tutaj jest działanie z premedytacją, zmierzające do zniszczenia systemu sądownictwa. W waszym sprawozdaniu też są same kwiatki. 17 grudnia ub.r. neo-KRS uznała, że wspieranie działalności charytatywnej jest wprawdzie co do zasady słuszne, ale może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. Skoro mamy już na sali przedstawicieli tego organu, to proszę wyjaśnić, skąd tak absurdalne i abstrakcyjne stanowisko. Czy np. polski sędzia może wesprzeć zbiórkę Caritas Polska?

Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Bardzo uprzejmie dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam do szanownych pań sędzi takie dwa pytania. Po pierwsze, do której tradycji nawiązywał pan sędzia Radzik, nazywając biuro rzecznika katownią? Panie powinny to wiedzieć, to jest to samo biuro. I drugie pytanie: Czy Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, której zadaniem jest przecież składanie wniosków do rady (Dzwonek) w przedmiocie żądania podjęcia czynności dyscyplinarnych, zauważyła w tej podłości pana sędziego Radzika coś nagannego i czy podjęła jakiekolwiek czynności wobec tej czarnej owcy, która hańbi imię środowiska sędziowskiego, nazywając siedzibę rzecznika dyscyplinarnego katownią?

Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oto ważny fragment tej rezolucji: Od wybuchu wojny w Ukrainie polskie władze podjęły szereg działań wprost sprzecznych z trzema warunkami postawionymi przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Po pierwsze, 25 lutego zawieszono polską sędzię Annę Głowacką za stosowanie prawa europejskiego oraz wyroków sądów europejskich. Po drugie, polski prezydent wręczył nominacje ponad 200 nowym, nieprawidłowo powołanym na wniosek neo-KRS tzw. neosędziom, w tym cztery nominacje do Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo! Ten raport nie jest raportem o działalności Krajowej Rady Sądownictwa, tylko jej atrapy, neo-KRS. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Słuchając tej informacji, mam wrażenie, że osoby zasiadające w neo-KRS żyją w jakimś matriksie. Zgodnie z konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Tymczasem neo-KRS nic nie robi i biernie przygląda się prześladowaniom sędziów za wybryki polegające na stosowaniu prawa unijnego i konstytucji. Niby sędzia Juszczyszyn wraca do orzekania, ale po to, byście go znów szykanowali przeniesieniem do innego wydziału. Ale co z pozostałymi, których represjonujecie? Kiedy przestaniecie prześladować takich sędziów jak Olimpia Barańska-Małuszek, Bartłomiej Przymusiński, Piotr Gąciarek, Monika Ciemięga czy Igor Tuleya? Ten twór, którego dotyczy dzisiejsza informacja, nie ma kompletnie nic wspólnego z prawdziwym KRS. Póki Krajowa Rada Sądownictwa nie stanie się niezależna i póki wszyscy sędziowie nie przestaną być przez was prześladowani, póty obywatel nie będzie mógł liczyć na niezależny sąd w każdej sprawie. Żadne kłamstwa i żadne pudrowanie syfu tego nie zmienią.

Do pana adresowany był projekt, poprawka, w istocie ustawa, która rozcinałaby ten węzeł gordyjski - to zbyt szumnie brzmi - właśnie tę plątaninę niepięknych powiązań, zależności, zaszłości. To jest projekt naszego kolegi Jakuba Kalusa - nasze biuro prawne - przez nas prezentowany i formalnie złożony, i jako ustawa, i jako poprawka. Ławnicy losowani, wybierani do tej roboty z szeregów istniejących ławników, tworzący sądy przysięgłych, które byłyby obligatoryjnie powoływane do każdej sprawy dyscyplinarnej. To pozwoliłoby wyjść z tego zaklętego kręgu przepychania się między waszymi a naszymi.

Co pan osobiście na jego temat uważa? Czy nie jest prawdą, że najważniejsze jest, żeby zachować wpływ, możliwość zdalnego sterowania stanem sędziowskim? Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Otóż art. 186 konstytucji mówi, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Pytam: Co zrobiliście w tej sprawie? Jakie działania podejmowała KRS w ostatnim roku i ostatnich latach, żeby wykonywać ten podstawowy, konstytucyjny obowiązek? Jak broniliście sędziów, którzy byli karani dyscyplinarnie? Czy zabieraliście głos w tej sprawie? Czy zwracaliście się do rzecznika dyscypliny o jakieś stanowiska, o to, na jakiej podstawie karze sędziów? Co zrobiliście, żeby bronić sędziów i niezawisłości sędziowskiej? Czy tylko dbaliście o własne etaty? Bo o to mam kolejne pytanie. Ilu z was ubiega się o awanse? Ilu z was wnioskuje samych siebie do siebie, żeby poprawić sobie byt i awansować do sądu wyższego szczebla? Ilu z was chce być w sądzie okręgowym, apelacyjnym czy w Sądzie Najwyższym? Bo to jest granda, że sędziowie, członkowie KRS-u ubiegają się sami u siebie o to, żeby awansować. Ile jest wakatów sędziowskich? Co zrobiliście w aferze hejterskiej? Co zrobiliście, żeby bronić godności sędziów? Wysoka Izbo! Pytam jako wieloletni członek Krajowej Rady Sądownictwa pod przewodnictwem najwybitniejszych prawników: pana Stanisława Dąbrowskiego, legendy ˝Solidarności˝, Romana Hausera, Dariusza Zawistowskiego, gdy standardem były wyraźne kryteria awansów, m.in. stabilność orzeczeń, terminowość uzasadnień. Ale pytam też o standardy, ponieważ sam broniłem sędziego, który został posądzony przez jednego z policjantów o to, że może być pod wpływem alkoholu. Nie podano wtedy alkomatu, w związku z tym nie był oskarżony, obwiniony o to, że odmówił, ale o to, że sam z własnej inicjatywy nie doprowadził do wyjaśnienia wątpliwości.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Ast, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Pytanie do pani przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa: Czy prawdą jest, że do tej pory w postępowaniach nominacyjnych, od 2019 r., uczestniczyło kilka tysięcy sędziów, adwokatów, prokuratorów, asesorów, że wynikiem tych postępowań było ponad 3 tys. wniosków nominacyjnych do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że ponad 2 tys. nominacji pan prezydent wręczył sędziom? Czy przypadkiem nie oznacza to, że jednak zdecydowana większość środowiska sędziowskiego uznaje status ustrojowy Krajowej Rady Sądownictwa? Bo chyba nie ma lepszego na to dowodu.

Widzicie państwo, jak się miło zrobiło. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do pani przewodniczącej: Czy to prawda, że Europejska Sieć Rad Sądownictwa to jest prywatna organizacja, że nie jest w żadnej strukturze Unii Europejskiej i że do tej sieci nie należą Austria, Czechy, Cypr, Finlandia, Estonia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja?

Proszę słuchać. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Zimoch, koło Polska 2050. Wysoki Sejmie!

To tak w największym skrócie. Proszę mnie utwierdzić w przekonaniu - mówię to oczywiście z przymrużeniem oka - że chodzi o sędziów hejterów. A tak na poważnie, proszę zdradzić, jakie jest stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa właśnie w sprawie tych sędziów hejterów. Czy czuje się pani komfortowo, kiedy w prezydium rady, obok pani znajduje się obecnie sędzia, który podczas zebrania sędziów podarł projekty uchwał podjętych przez innych sędziów, a dzisiaj niezgodnie z przepisami wysyła na urlop przywróconego do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna, ba, niezgodnie z przepisami przesuwa go do innego wydziału? A do pana posła Smolińskiego: panie pośle, gdzieś jest granica absurdu. Czy to, że w wielu krajach nie skacze się na nartach, oznacza, że nie będziemy doceniali sukcesów polskich skoczków narciarskich? Pani posłanka Katarzyna Maria Piekarska, Koalicja Obywatelska. Wielce Szanowny Panie Marszałku! Pani Sędzio!

Dzięki temu można sobie zarobić spokojnie drugą pensję. Pani sędzia Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor udzieliła bardzo ciekawego wywiadu. Czy pani się zgadza z panią prezes Manowską, że obok likwidacji Izby Dyscyplinarnej trzeba także zreformować Krajową Radę Sądownictwa? Czy pani zdaniem to, że prokuratura czwarty rok, to już blisko 4 lata, wyjaśnia aferę hejterską nie jest po prostu skandalem? Czy nie ma pani takiego poczucia, czy ja wiem, absmaku, że została pani szefową KRS w sytuacji, gdy jest pani koleżanką ministra sprawiedliwości?

Być może to jest zbieg okoliczności, ale ja w zbiegi okoliczności nie wierzę, bo już za długo żyję. Dziękuję. Panie pośle, odpowiem panu, bo chciał pan, żebym skrócił wypowiedź. Nie skróciłem tej wypowiedzi dlatego, że pani przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa przedłużyłem wypowiedź o 4 minuty. Niech pan sobie wyobrazi, że próbuję i staram się prowadzić te obrady w sposób sprawiedliwy.

Czy poseł sprawozdawca pan. Ale to króciutkie było to pytanie, panie pośle. Dobrze, to już mi się zaczyna podobać. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tych pytań było tak wiele, że nie sposób na wszystkie odpowiedzieć, ale część z nich dotyczyła kwestii, które nie są związane ze sprawozdaniem, więc pozwolicie państwo, że nie odpowiem na wszystkie pytania, które tu padły.

Proszę państwa, Krajowa Rada Sądownictwa nie jest ani sądem dyscyplinarnym, ani organem powołanym do zarządzania sądami, czyli te wszystkie uwagi dotyczące sprawności postępowań sądowych, jakości tych postępowań nie dotyczą nas bezpośrednio. Tutaj nie będę się wypowiadać.

Tak najprościej można to ująć. Proszę państwa, w związku z tym, że to właśnie sędziowie, którzy zostali powołani na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, są najbardziej atakowani - z przykrością stwierdzam, że mówi się, że wyrzuci się ich z zawodu czy wrócą, skąd przyszli - Krajowa Rada Sądownictwa. To jest naturalne, ponieważ oni podlegają atakowi. Jeżeli chodzi o sędziów, którzy występują w mediach i często są wymieniani jako obrońcy niezawisłości, niezależności, to przynajmniej co do niektórych mogę powiedzieć, że ich odsunięcie od czynności, od obowiązków było spowodowane szkodami, które czynili obywatelom. Bo proszę państwa, jeżeli sędzia odmawia nadania klauzuli wykonalności, która jest czynnością. którą ma wykonać referendarz sądowy - nie jest czynnością orzeczniczą, nie jest rozstrzyganiem niezawisłych spraw - tylko demonstracyjnie odmawia nadania klauzuli wykonalności, bo w sądzie niższej instancji uznał, że nie będzie uznawał sądu apelacyjnego, który notabene oddalił apelację. Pani Poseł! Ci dzielni sędziowie, jeden z tych dzielnych sędziów wysyła mi kartki, już chyba ze 20 wysłał, to są otwarte kartki.

Bo proszę państwa, nawet z tej uchwały siedmiu sędziów Izby Karnej. nie wynika, że ktoś nie uznaje statusu tych sędziów w sensie prawa do wynagrodzenia, w związku z czym to nie były działania podejmowane w interesie tych sędziów w sensie ich wynagrodzenia. Mam ją tutaj, ale nie będę jej odczytywać, bo szkoda czasu. Tutaj złożę skargę na posła Asta, wkręcił mnie, powiedział, że mam czas dowolny. Bardzo przepraszam. W związku z tym to sprawozdanie nie było ułożone w takiej formule, jak powinno być, bo może były istotniejsze elementy, ale ono jest pisemne. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia członków rady, to wszystko leży w gestii Sejmu, parlamentu.

Natomiast. Przepraszam, to jest nieporozumienie. Komisje zdalne działały podczas. Ja nie mam pojęcia, bo. Teraz jest wprowadzony taki zeszyt i trzeba szczegółowo pisać, co poszczególny członek rady robił.

Przepraszam bardzo, pani przewodnicząca. Proszę państwa! Mówię do panów. Proszę nie ruszać głową, bo dobrze pan wie, jak są obrady prowadzone. Możemy od tego momentu uznać, że jedni w trakcie przemówień drugim nie przerywają. Jeśli tak uznamy, to taką zasadę wprowadzimy. Nie wprowadziłem tej zasady, bo jedni byli warci drugich. Więc jeżeli państwo tak prosicie, to proszę i jedną, i drugą stronę o rozsądek. Pani przewodnicząca, proszę bardzo. Dysponujemy kontrolą Najwyższej Izby Kontroli, która była pozytywna, jeżeli chodzi o finanse rady za 2021. Jeżeli więc są wątpliwości co do rzetelności tej kontroli, to trzeba się zwrócić do Najwyższej Izby Kontroli, bo ja za tę instytucję nie odpowiadam. Proszę państwa, jeżeli chodzi o tzw. podwójne diety, to nie było niczego takiego.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o awanse sędziów, to też wszystko w rękach państwa. Możecie zmienić przepisy ustawy w ten sposób, że członkowie Krajowej Rady Sądownictwa nie będą mogli się ubiegać o wyższe stanowiska sędziowskie. W poprzednich kadencjach rady również były takie wnioski do prezydenta, część spotkała się z akceptacją głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, część nie. W poprzedniej kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, jak już mówiłam, jeżeli chodzi o członków rady, tak naprawdę awansowały dwie osoby. Wśród tych dwóch osób jestem ja. Nie jesteśmy też, panie pośle Braun, instytucją do oceny prawidłowości ustaw ogłaszanych przez parlament czy rozporządzeń ministrów we wszystkich sprawach.

Tak troszeczkę tylko. Postaram się króciutko. Jeżeli chodzi o system wyłaniania najlepszego kandydata w konkursach, to oczywiście - oprócz konkursu do Sądu Najwyższego - nie ma tam obligatoryjnych wysłuchań kandydatów. Działamy w oparciu o dokumenty. Te dokumenty są zebrane wcześniej, na etapie tej procedury jeszcze przed prezesami sądów.

A więc możemy zwiększyć tę ilość wysłuchań. Jeżeli chodzi o Europejską Sieć Rad Sądownictwa, proszę państwa, to nie zdradzę chyba jakiejś tajemnicy najwyższej rangi, jeśli powiem, że w momencie kiedy zaczęliśmy działalność, odwiedziła nas delegacja z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i ta rozmowa przebiegała w taki sposób, że bardzo szybko zorientowałam się, że nas w ciągu jakiegoś spodziewanego czasu usuną z tej sieci. Zapytałam kolegę z jednego z krajów bałtyckich, który był, czy nas z tej sieci usuną.

Trwał dialog. W końcu stało się tak, że zawieszono nas w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. My nie uznawaliśmy tego zawieszenia, ponieważ nie było to przewidziane w statucie.

Na szczęście - bo na początku wszyscy byli przeciwko nam - ta decyzja akurat, z tego, co wiem, nie zapadła tak gremialnie, jednoznacznie przeciwko nam. Rzeczywiście trwa w dalszym ciągu wymiana korespondencji z Europejską Siecią Rad Sądownictwa i utrzymywany jest dialog. Nie jesteśmy obrażeni, nie zamierzamy pozywać tej sieci przed. Chyba że rada in gremio zobowiąże przewodniczącego do wystąpienia w takiej sprawie. Jeżeli chodzi o stanowisko rady w sprawie działalności charytatywnej, to już mówiłam na posiedzeniu komisji, że to jest wielkie nieporozumienie, ponieważ nie zabraniamy sędziom, broń Boże, działalności charytatywnej. Zwracaliśmy tylko uwagę, żeby nie zajmować się dobroczynnością z wykorzystaniem statusu sędziego, żeby nie nabijać sobie tym punktów wśród obywateli. Stanowisko to zostało przyjęte na skutek skargi obywatela, a nie z naszej własnej inicjatywy. Po prostu rozpoznaliśmy całokształt tej sprawy i komisja etyki zaproponowała radzie uchwałę o treści, którą państwo znacie, bo jest stanowiskiem rady. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o działalność w mediach społecznościowych sędziów, to jeżeli chodzi o tzw. aferę hejterską, to ja nic nie mogę na ten temat powiedzieć. To są materiały, dla mnie jako sędziego, medialne. A ja nigdy nie wypowiadam się na temat, nie osądzam sprawy w oparciu o materiały medialne, których prawdziwości nie mogę zweryfikować. Nie prowadzę takiego postępowania ani dochodzenia. Jeżeli miały miejsce działania o charakterze mowy nienawiści, to oczywiście to stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa dotyczy wszystkich, w tym takich zachowań. Bo nie wiem, czy paniom posłankom by się podobało to, że sędzia do prezesa, kobiety prezesa. Na Twitterze pod jakąś tam publikacją, linkiem prasowym: cała ona, kocham ją, serduszko. Proszę państwa, jeżeli chodzi o inne poruszone kwestie, to tutaj państwo posłowie, członkowie rady wskazywali na ilość kandydatów, którzy zgłaszali się do rady.

W całej kadencji to było 2411 wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Już mówiłam pani poseł, że po prostu nie wypada. Natomiast, jeżeli mogę coś dodać, to z pewnością nie należy do katalogu praw człowieka prawo, żeby sędziowie wybierali sędziów, którzy wybierają sędziów. Nie ma takiego prawa (Dzwonek) w katalogu praw podstawowych. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! To ja może jeszcze raz powtórzę.

Niektórzy członkowie neo-KRS-u zamiast pracować w komisjach w dniach, w których wypadają posiedzenia plenarne, zaczęli się spotykać w innych terminach. W efekcie zamiast jednej diety były im wypłacane dwie. Co ważne, jak podawała prasa, posiedzenia komisji odbywały się bardzo często w formie on-line i zazwyczaj trwały bardzo krótko. Te spotkania trwały od 31 minut do 109 minut, średnio 66 minut, i tysiączek wpadał. Pan poseł Ast w sumie zarobił ile? Obecny tu pan Smoliński - 43 tys. zł. Sprawozdawca komisji pan poseł Marek Ast. Zapraszam pana posła. Panie Marszałku! Na początek taka uwaga. Ze zrozumieniem przyjąłem zaproponowany przez pana marszałka sposób prowadzenia tej debaty, polegający na wchodzeniu przez posłów w interakcje z salą, natomiast jeżeli chodzi o przedstawicieli organów konstytucyjnych państwa, którzy występują na sali sejmowej, to oni raczej nie mają możliwości przerywania posłom ich wystąpień.

Bardzo proszę.

Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana posła Brauna, to powiem, panie pośle, że absolutnie jesteśmy za zwiększeniem czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, ale projekty ustaw, które są zgłaszane przez Konfederację, powinny też być zgodne z polską konstytucją.

Zamykam dyskusję.

czasie treningu, oraz udziału w pozorowanej akcji ratowniczej czy też udziału w akcji ratowniczej. Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu na petycję, którą komisja uznała za zasadną. Aktualne przepisy zawarte w obu zmienianych ustawach zakazują wprowadzania bądź puszczania psa luzem w czasie treningu w lesie oraz w miejscach przyrodniczo chronionych. Proponowana zmiana w ustawie Kodeksu wykroczeń eliminuje ryzyko sankcji za puszczenie psa ratowniczego luzem podczas szkolenia i działań ratowniczych. Wysoka Izbo! W akcjach poszukiwawczo-ratowniczych uczestniczą ratownicy wraz ze swoimi psami. Zwierzęta te muszą być przez kilka lat szkolone. Jednym z elementów egzaminu certyfikowania jest poszukiwanie osoby zaginionej w terenie leśnym. I tutaj pojawia się problem, ponieważ pies tropiący podczas treningu w terenie leśnym według obecnych przepisów musi być trzymany na smyczy przez swojego przewodnika. Czyli zdaje on egzamin z poszukiwania osoby zaginionej bez żadnego skrępowania, a ćwiczony jest na krótkiej smyczy przy nodze przewodnika. Podczas akcji ratunkowej pies odbiega od swojego przewodnika nawet na kilkaset metrów, dlatego również podczas treningu powinien biegać i szukać w sposób nieskrępowany. Psów certyfikowanych do poszukiwań jest w Polsce ok. 100, a zatem treningi będą sporadyczne i zazwyczaj będą odbywać się pojedynczo, dlatego nie ma zagrożenia, że zmiana ustawy doprowadzi do atakowania czy straszenia dzikiej zwierzyny przez psy trenujące w terenach leśnych. Projekt zmiany ustawy, który mam zaszczyt przedstawić, popiera m.in. Państwowa Straż Pożarna oraz kilkanaście stowarzyszeń i grup poszukiwawczych z całej Polski. Zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie likwidacja istniejącego od wielu lat dysonansu pomiędzy stanem prawnym a potrzebą jak największej skuteczności działań ratowniczych podejmowanych z wykorzystaniem psów ratowniczych. Ze względu na swój charakter i ograniczony zasięg ustawa nie wywoła skutków gospodarczych, jak również skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Wysoka Izbo! Panie Marszałku! W imieniu Komisji do Spraw Petycji, którą mam zaszczyt reprezentować, proszę o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w komisji. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę pana posła Dariusza Bąka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zabranie głosu. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko odnośnie do projektu ustawy z druku nr 1971. Wysłuchaliśmy przed chwilą uzasadnienia tego projektu ustawy, ale chciałbym zwrócić uwagę na niektóre sprawy, które zostały tu poruszone.

Kodeks wykroczeń, mających na celu umożliwienie psom ratowniczym udziału w treningach w lesie poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie psów ratowniczych w czasie treningu, udziału w pozorowanej akcji ratowniczej czy też udziału w akcji ratowniczej.

Pani posłanka Katarzyna Maria Piekarska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Kodeks wykroczeń. Ten projekt ustawy to efekt petycji skierowanej do Sejmu. Widać, że warto podejmować inicjatywy legislacyjne w ważnych dla danych grup kwestiach.

Historycznie po raz pierwszy zauważono te zdolności w XVII w. Jeśli chodzi o poszukiwanie ludzi np. pod lawinami, to był to XVII w. Były to bernardyny hodowane przez mnichów na Przełęczy Św. Wysoka Izbo! Aby te psy mogły być wykorzystywane do poszukiwań osób zaginionych, muszą, co oczywiste, jak wspominał pan poseł sprawozdawca, przejść odpowiednie szkolenie. Musi to być szkolenie w różnych terenach, w tym także w lesie, aby pies nauczył się wykorzystywać te swoje niezwykłe zdolności w służbie człowiekowi.

W projekcie postuluje się zmianę art. 30 ust. 2, aby możliwość puszczania psa luzem dotyczyła również psa ratowniczego w trakcie szkoleń i akcji ratowniczych. W obecnym stanie prawnym istnieją jedynie nieliczne wyjątki od zakazu puszczania psa luzem. Chodzi o dopuszczenie do organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników górskich i psów ratowniczych na terenie parku narodowego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, ale to jest zdecydowanie za mało. Projekt przewiduje też zmianę art. 166 Kodeksu wykroczeń, która eliminuje ryzyko sankcji za puszczanie psa ratowniczego podczas szkolenia. Wysoka Izbo! Naszym zdaniem ten projekt zasługuje na poparcie, dlatego jesteśmy za dalszym skierowaniem go do prac w komisjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Szejna. Nieobecny.

Szczęść Boże!

I oczywiście z pewną ulgą przyjmuję taki miły projekt. Jedna jest taka, że wpłynęła petycja. Oto Sejm pochylił się nad nią. Ona aż tutaj do nas dopłynęła. Wręcz przeciwnie, cieszy nas choćby wycinkowa, choćby tylko do terenów leśnych ograniczona tendencja powrotu jakiejś normalności. Bywałem w lesie, bywałem i z psami. Miewałem oczywiście do czynienia również z nieodpowiedzialnymi ludźmi, którzy źle wychowali swoje psy. Wiemy wszyscy, że to jest problem. W związku z tym norma prawna, która zobowiązuje właścicieli psów do tego, żeby poważnie traktowali możliwe zagrożenia wynikające ze złego ułożenia zwierzaka, nie powinna być uchylona, ale jednak bądźmy poważni, bądźmy normalni.

Szanowni państwo, nie traktujmy tego projektu jak jakiegoś tam drobnego, nieważnego, jak jednego z michałków, które tutaj, w Sejmie, się trafiają.

Może skoro nie chcemy, chwała Bogu, mam nadzieję, że do tego się wszyscy przychylą, stawiać świata na głowie i ścigać myśliwych, ratowników i strażaków, którzy z psami robią to, co im kunszt, przeszkolenie i tradycja nakazują, to może przestańmy też ścigać ludzi. Może przestańmy ścigać i czołgać myśliwych, którzy zabierają do lasu swoje świadome i wychowywane w pięknej tradycji dzieci. A Sejm tej kadencji przecież właśnie zabrał się za penalizowanie i delegitymizację tradycji myśliwskich. Wróćmy do normalności nie tylko w tym wąskim zakresie, także w sprawie dostępu do broni palnej, bo przecież to się łączy z tym procederem polowania. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo uprzejmie dziękuję. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Wysoka Izbo! Celem projektu ustawy jest dokonanie zmian w ustawie o lasach i w Kodeksie wykroczeń, które mają na celu generalnie dopuszczenie do możliwości szkolenia psów ratowniczych, udziału w treningach na terenach leśnych poprzez wyłączenie tego procesu szkolenia z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie, psów ratowniczych w trakcie treningu, udziału w pozorowanej akcji ratowniczej czy też udziału w akcji ratowniczej.

Kiedy jest to zasadne, parlament również opracowuje projekt ustawy i ta ustawa jest procedowana w Wysokiej Izbie. Nie trzeba być posłem, nie trzeba zebrać 100 tys. podpisów, ale właśnie taką drogą petycji skierowanej do parlamentu również można wpływać na zmiany w prawie.

W związku z tym celowe jest wprowadzenie różnego rodzaju szkoleń w warunkach terenowych, ponieważ tylko takie szkolenia są w stanie zapewnić odpowiedni poziom wyszkolenia psa, a to warunkuje niesienie szybkiej i skutecznej pomocy.

Niemniej jednak Koło Parlamentarne Polska 2050 widzi potrzebę dalszych prac nad przedstawionym projektem. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Aktualne przepisy zawarte w obu zmienianych ustawach zakazują bądź wprowadzania psów do lasów, bądź też puszczania ich luzem na terenach lasów oraz obszarów objętych ochroną ścisłą i czynną. Nieliczne wyjątki od tej zasady występujące w prawie nie dotyczą szkoleń i działań podejmowanych przez psy ratownicze. Jednym z nich jest dopuszczenie organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników psów górskich i psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, na obszarze parku narodowego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody na zasadach uzgodnionych z dyrektorem parku narodowego. Tak więc przeprowadzanie szkoleń psów ratowniczych jest obecnie możliwe na określonych warunkach na terenie parków narodowych, ale nie jest możliwe w lasach. Chciałbym w imieniu klubu Lewica z zadowoleniem przyjąć zaproponowane przepisy i regulacje i zagwarantować, że klub Lewica z zadowoleniem weźmie udział nad procedowaniem nad dobrymi rozwiązaniami w ramach tej ustawy. W imieniu ratowników oraz przewodników psów ratowniczych chciałbym bardzo serdecznie podziękować autorom projektu za potrzebne i, jak się wydaje, bardzo oczywiste regulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby się dopisać do listy? Jeżeli nie, zamykam listę. Ustalam czas zadawania pytania - 1 minuta. Zapraszam pana posła Jana Szopińskiego, który skończył przed chwilą swoją przecudną przemowę i zacznie teraz drugą. Bardzo proszę. Obawiam się że dotychczasowe przepisy bardziej ograniczały pracę formacji ratowniczych, niż wpływały na swobodne wypuszczanie psów na terenach leśnych. Problem wypuszczanych, a często porzucanych psów wymaga szeregu dodatkowych regulacji w polskim prawie. Ale biorąc pod uwagę osiągnięcia obecnej władzy w reformowaniu naszego życia, będzie chyba lepiej dla czworonogów, gdy tym problemem zajmie się już kolejna ekipa rządząca. Z tego miejsca, korzystając z okazji, tej debaty, chciałbym podziękować wszystkim schroniskom, domom tymczasowym dla zwierząt, prywatnym ludziom wspierającym taką działalność oraz samorządom za ich wkład pracy w opiekę nad wszystkimi zwierzętami. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dzisiaj rozpatrywana ustawa jest ważnym elementem obywatelskości, czyli możliwości wpływania obywateli na tworzenie prawa przez petycje. Ta petycja zmierzająca do realizacji możliwości szkolenia psów ratowniczych luzem w lesie dzisiaj ma szansę uzyskać naszą rekomendację w czasie prac parlamentarnych. Korzystając z obecności na sali pana posła, pana ministra Edwarda Siarki, który na co dzień również nadzoruje Lasy Państwowe, chciałbym może zapytać, w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi mówiących o tym, że w parkach narodowych można to już czynić, ale po uzgodnieniu z dyrektorem parku.

Dziękuję. Pan poseł Rafał Adamczyk. Nie ma. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana posła, który jest przedstawicielem komisji. Chciałem zapytać, czy wnioskodawca tego projektu ustawy pojawił się na posiedzeniu komisji i czy przedstawił również osobistą motywację dotyczącą podjęcia tego typu projektu ustawy? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Nie mogę się jednak oprzeć, żeby nie skorzystać z pańskiej obecności tutaj - zwracam się do pana ministra Siarki, pełnomocnika rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa. Pytanie przy okazji, wykraczające rzecz jasna poza materię tej ustawy. Jaka będzie jej cena? Jaka będzie jej dostępność? Czy może przez Pocztę Polską można by je rozprowadzać? Panie ministrze, wiązka chrustu+ od Lasów Państwowych - za pośrednictwem rozmaitych innych molochów.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Wanda Nowicka, Lewica. Szanowna Pani Marszałkini! Wysoka Izbo!

Ale moje pytanie jest takie. Ta ustawa tego nie obejmuje. Jeżeli tak, to z mojego punktu widzenia jest to w porządku.

Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu tego projektu jest mowa wyłącznie o potrzebie i prawie zwolnienia ze smyczy psów na obszarach leśnych w czasie ich szkolenia i akcji ratowniczych.

Dziękuję bardzo. O odpowiedź na pytania proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pana ministra Edwarda Siarkę.

Wysoki Sejmie!

Niejednokrotnie środowisko ratowników i specjalizujących się w tym strażaków, którzy prowadzą specjalne grupy ratowniczo-poszukiwawcze. Na terenie Małopolski jest ich kilka.

Z naszego punktu widzenia - mówię o Ministerstwie Klimatu i Środowiska - jest pełne poparcie dla tego pomysłu, dla tego rozwiązania.

Chcielibyśmy rozdzielić samą kwestię szkolenia.

Myślę, że w pełni dojdziemy do porozumienia w tych kwestiach i rzeczywiście rozwiążemy ważny temat, istotny z punktu widzenia ratowania życia ludzkiego, temat dostępności dla służb ratowniczych.

Natomiast rzeczywiście, jeśli spacerujemy po lesie, a tam luzem biegają często, powiedzmy sobie.

Myślę, że to jest kwestia oznakowania tych psów.

Tu nie o to chodzi. Proszę państwa, pan poseł Braun wraca do sprawy, która. Nie wiem, dlaczego pan poseł akurat przy tej okazji to porusza, ale muszę powiedzieć - i to bardzo wyraźnie - że w ostatnich dniach rzeczywiście pojawiły się różnego rodzaju memy na temat tego, jakoby był uruchomiany jakiś specjalny program chrust+. Proszę państwa, chcę bardzo wyraźnie z tej trybuny powiedzieć: nigdy w tej sprawie się nie wypowiadałem, nie znajdziecie państwo mojej wypowiedzi, mimo że w środkach przekazu, zwłaszcza w mediach społecznościowych, przypisano mi słowa, których nigdy nie powiedziałem.

Nic więcej. Tylko tyle.

To dzieje się od lat.

Nic takiego nie ma miejsca, tym bardziej że - tak jak mówię - program jest dostępny dla ludzi od lat i wszyscy ci, którzy korzystają z drewna w Polsce, rozumieją ten problem.

Do tego jeszcze dochodzi 500 tys. kominków, gdzie też drewno jest wykorzystywane. Nie rozumiem więc, dlaczego, że tak powiem, robimy wokół tego hejt, skoro przecież z tego drewna korzystamy. Co więcej, Komisja Europejska wszystkie te elementy związane z biomasą traktuje jako zeroemisyjne. To jest w naszym interesie, żebyśmy korzystali z tego surowca.

Przepraszam, że być może za długo na ten temat mówię, ale ponieważ padło to pytania przy okazji tego, o czym dzisiaj mówimy. Jeśli panu się udało. Nie unikam tego tematu. Panie pośle, wie pan, ten temat ma duże wzięcie w mediach społecznościowych, nawet ostatnio oglądałem ciekawe materiały, które ukazały się gdzieś tam w radiu czy w telewizji, bardzo ciekawe intelektualnie, wie pan, na wysokim poziomie.

Dziękuję, pani marszałek. W trybie sprostowania pan poseł Braun. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pan mówi, że nie wiadomo, skąd ta fala memów. Pan minister Kowalczyk ostatnio wszedł nawet w taką polemikę medialną. Mówił, że chrust, patyczki to może nie, ale konary - proszę bardzo. Nie lekceważę tego, wręcz przeciwnie, nawet mam się za wykwalifikowanego w tej dziedzinie.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Kodeks wykroczeń, zawarty w druku nr 1971, do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 56. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczanie? Zamykam listę. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Wanda Nowicka. Szanowna Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Chciałabym złożyć wyrazy ubolewania, że Prawo i Sprawiedliwość nieustannie zajmuje się dwiema grupami społecznymi i najczęściej to zajmowanie się nie wychodzi tym grupom na dobre. Przede wszystkim mam na myśli w tym przypadku kobiety i dzieci, młodzież. Jeśli chodzi o kobiety, dużo już było dzisiaj mowy o represyjnej ustawie antyaborcyjnej i jej skutkach, także o rejestrze ciąż, który stwarza kolejne zagrożenie i wywołuje niepokój wśród kobiet, że prokurator może się interesować ich ciążami, i to akurat niekoniecznie z najlepszych pobudek, tylko po to, żeby ścigać je w przypadku, gdyby okazało się, że z tej ciąży nie urodziło się dziecko.

Mam nadzieję, że to nastąpi.

Jeśli chodzi o młodzież i dzieci, znowu to jest kwestia edukacji, kwestia szkół.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Wszyscy mamy świadomość, że krew to dar życia, a oddawanie krwi jest aktem solidarności. Dlatego chcę dziś zwrócić uwagę na wielką rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa w ratowaniu życia, na to, jak wpływa ono na wzmacnianie solidarności w społecznościach lokalnych. Wszystkim krwiodawcom dziękuję za to, że poświęcają cząstkę siebie, aby nieść pomoc innym ludziom. Życzę wam zdrowia oraz tego, abyście w każdym miejscu i czasie cieszyli się ludzką wdzięcznością i szacunkiem, bo z pewnością na to zasługujecie. W tym dniu pragnę również podziękować całej społeczności aktywnej w ruchu honorowego krwiodawstwa. Dzięki waszemu zaangażowaniu możliwe jest zapewnianie krwi osobom potrzebującym. Dlatego na ręce społeczników i pielęgniarek Polskiego Czerwonego Krzyża i jednostek publicznej służby krwi składam dziś najlepsze życzenia pomyślności i satysfakcji z prowadzonej działalności i pełnionej służby. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie! Nestor polskich historyków - też z Piotrkowa. Jest taka ulica w moim Piotrkowie, niedługa, wzdłuż dawnych murów miejskich, wychodzi wprost na kamienicę z dużą, pamiątkową tablicą. W tym domu mieszkał, pracował i zmarł Kazimierz Stronczyński. Tylko nieliczni historycy znają to nazwisko, a szkoda. Bo był to człowiek, który tworzył zręby nowoczesnych polskich nauk historycznych. Urodził się w 1809 r. Ciekawe, że dokładne daty zarówno urodzin, jak i śmierci nadal budzą wątpliwości. Edukację zaczął w kolegium pijarskim w Piotrkowie i kontynuował ją na Uniwersytecie Warszawskim. Był nauczycielem i urzędnikiem, walczył w wojnie z Rosją w latach 1830-1831. Realizował ją, zarówno stojąc na czele komisji rządowej, przeprowadzając pierwszą tak gruntowną inwentaryzację zabytków w Królestwie Polskim, jak i po pracy zajmując się sfragistyką i swoją ukochaną numizmatyką. Jego opus magnum to ˝Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim˝, dziś nazywane albumami Stronczyńskiego. W pięciu tomach, zrealizowanych z benedyktyńską cierpliwością, ujęte zostały ówczesne znane zabytki z dokładnym opisem, umiejscowieniem i wieloma akwarelami i gwaszami. Publikował także doskonałe prace o tematyce numizmatycznej, zbierając informacje o monetach w średniowiecznej Polsce oraz o pieczęciach, w czym był pionierem. Jego prace do dziś są ważnymi opracowaniami dla historyków, tym bardziej że dziś wiele zabytków, które opisał Kazimierz Stronczyński, już nie istnieje. Był bezsprzecznie prekursorem rozwoju nauk pomocniczych w historii. Zmarł w Piotrkowie w roku 1896, gdzie został także pochowany, na Starym Cmentarzu. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł. Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wszyscy chwalą ludzki rząd, który wprowadził ułatwienia w zbieraniu chrustu. Tą sprawą żyje cały kraj, bo oddaje ona dosyć dobrze absurdalne podejście do ekonomii obecnej ekipy. Efekt, jaki wywołali swoją wypowiedzią, jest jak zwykle odwrotny do tego, co sobie zaplanowali. Wcześniej leśniczy przymykali oko, gdy ktoś zabrał kilka gałęzi, a teraz poprzez narodową zbiórkę chrustu leśniczy będą brać kasę za każdą wiązkę. Ludzie na wsi, także elektorat PiS-u, są wściekli, bo takimi pomysłami się ich po prostu upokarza. Prawda jest taka, że chrust powinien zostać w lesie. Las to nie tylko drzewa, gałęzie są ważną częścią ekosystemu, są elementem ściółki leśnej, dzięki nim rozwijają się mikroorganizmy, lasy żyją, a butwiejące drewno jest tego nieodzowną częścią. Poza tym palenie chrustem jest gorsze nawet niż palenie węglem. Powinniśmy ogrzewać domy czystą energią, dofinansowywać pompy ciepła, fotowoltaikę i inwestować w farmy wiatrowe.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Maciej Kopiec, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze Niedzielski! Zwracam się do pana z apelem w imieniu osób chorych na mukowiscydozę. Mukowiscydoza to ciężka choroba genetyczna, która uniemożliwia normalne, codzienne funkcjonowanie, a nieleczona prowadzi do śmierci. Chorzy każdego dnia zmagają się z silną dusznością, brakiem kondycji i ryzykiem infekcji podczas licznych wizyt w szpitalach. Choroba postępuje, a o normalnym życiu Ania może jedynie pomarzyć. Ciągłe infekcje oraz duszności nasilające się przy każdym ruchu spowodowały, że musiała zrezygnować ze studiów. Podstawowe czynności, takie jak zakupy czy sprzątanie, również sprawiają jej ogromny problem. Obecnie oczekuje na leki przyczynowe, które są dla niej ostatnią szansą na normalność. Niestety, nadzieja Ani gaśnie z dnia na dzień coraz bardziej, ponieważ Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, który ma ją pod opieką, wciąż nie otrzymał leku, bo proces porozumienia w sprawie refundacji wciąż się wydłuża. Wśród pacjentów panuje strach. Nie dość, że ich życie jest zagrożone chorobą, to nie wiedzą, czy w ogóle i kiedy ich leczenie będzie kontynuowane. Mają poczucie, że są pozbawieni wsparcia. To tylko jedna z ok. 3 tys. historii chorych na mukowiscydozę, z których zaledwie 1 tys. kwalifikuje się do leczenia refundowanymi lekami, a tylko te są sprawdzone, skuteczne i faktycznie ratują życie. Niestety chorzy z Polski są często zmuszani do samodzielnego organizowania zbiórek i wyjazdów za granicę w celu kontynuowania leczenia, którego koszt wynosi nawet 87 tys. zł miesięcznie. Mimo wcześniejszych apeli o zmianę tej sytuacji i zapewnień pana ministra o wsparciu do dziś osoby chore nie mają informacji, czy i kiedy będą mogły rozpocząć ratujące im życie terapie. Mukowiscydoza nie zna litości, nie czeka, postępuje i niszczy organizmy młodych ludzi takich jak Ania. Statystycznie chorzy na tę chorobę w Polsce żyją kilkanaście lat krócej niż w krajach zachodniej Europy. Ta drastyczna różnica to wstyd dla Polski. 1 marca tego roku chorzy po wielu latach codziennego cierpienia dostali obietnicę normalnego życia. Proszę pana ministra, aby ośrodki jak najszybciej otrzymały obiecane przez rząd środki na leczenie, a informacje dotyczące postępowania w sprawie refundacji leków były na bieżąco upubliczniane. Apeluję, aby procesy prowadzące do udostępnienia leków zostały natychmiast przyspieszone, ponieważ sytuacja chorych w Polsce jest dramatyczna, a każdy dzień opóźnienia może oznaczać wyrok śmierci dla kolejnej chorej osoby. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja.

Oświadczenie poselskie odnoszące się do obecności tutaj, w Wysokiej Izbie w dniu dzisiejszym pana wiceministra Waldemara Kraski. Pan Waldemar Kraska - wiceminister zdrowia lub, jak każe mi mówić doświadczenie ostatnich lat, wiceminister w resorcie choroby i nagłej śmierci składał tu dziś Wysokiej Izbie pewne wyjaśnienia, odpowiadał na pytania w ramach standardowego punktu: Informacja bieżąca. Zadałem panu ministrowi pytanie o jego biografię, o jego życie, dłuższe niż moje o ładnych parę lat, a tak jakby rozpoczynające się dopiero w roku 1989.

Zapytywałem resort i zapytywałem Instytut Pamięci Narodowej o oświadczenie lustracyjne Waldemara Kraski. Z korespondencji, która została skierowana akurat nie do mnie, ale do pewnego historyka, który podążył tym samym tropem, wynika, że oświadczenie lustracyjne przynajmniej jedno jest, owszem, w posiadaniu Instytutu Pamięci Narodowej, ale - uwaga - z analizy kontekstowej pisma wynika, że to oświadczenie nie było w ogóle weryfikowane. I za to z ostrożności i z troski o to, by Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie wysłuchiwał tutaj być może osób, których funkcjonowanie w życiu publicznym jest obciążone jakimś felerem prawnym, który by np., o zgrozo, mógł prowadzić do wniosku, że wszystkie decyzje Waldemara Kraski, w tym decyzje podjęte w latach walki z mniemaną pandemią, były bezprawne, bo obciążone tym felerem, tą wadą.

Już kończę, pani marszałek. Moje dzisiejsze oświadczenie poselskie proszę traktować jako doniesienie publiczne. Pani marszałek od tej chwili z urzędu posiada wiedzę o tym, że uzasadnione jest podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przez samego Waldemara Kraskę, albo przez osoby, które nie dopełniły obowiązku weryfikacji jego oświadczenia lustracyjnego. albo też przez inne nieznane mi osoby trzecie, czwarte i piąte. Tak czy inaczej składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, którym byłoby kłamstwo lustracyjne w przypadku Waldemara Kraski.

Może szkolenia, może działania, może służba dla resortu zielonego, niebieskiego - tego nie wie nikt, ale niechaj się dowie. Kto? Prokurator. Na wniosek pani marszałek, która z urzędu wiedząc, z urzędu ma obowiązek zawiadomić. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica.

Wysoki Sejmie! Moje oświadczenie dotyczy bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie. Dzisiaj pan premier, przedstawiając z tej mównicy osiągnięcia rządu, mówił m.in. o dopłatach do nawozów, pomocy w zakresie zakupu oleju opałowego czy pomocy dotyczącej energii elektrycznej. W tej chwili złożone wnioski o dopłaty do nawozów sztucznych nie są realizowane.

Ponadto dopiero rozpocznie się nabór wniosków, jeśli chodzi o pomoc suszową za ubiegły rok. Pieniądze na nawóz trzeba było wydać, zwiększone koszty związane z energią, gazem trzeba ponosić, cena 1 kg żywca spadła bardzo nisko i bardzo wiele gospodarstw zrezygnowało z hodowli trzody chlewnej. W związku z powyższym wiele rodzin jest w trudnej sytuacji materialnej, dlatego też chciałbym zaapelować do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, aby ogłaszane publicznie programy były w miarę sprawnie wdrażane przez administrację podległą panu ministrowi i nie doprowadzały do upadłości gospodarstw rolnych. Pani poseł Anita Sowińska, Lewica.

Mowa tu oczywiście o fabrycznie nowych samochodach, więc proces ten będzie następował stopniowo. Ta decyzja jest dobra z kilku powodów. Pierwszy powód to jest zbrojna napaść Rosji na Ukrainę, która wymaga od nas wszystkich odpowiedzialności. Każdy litr ropy zakupionej z Rosji to są zabici ludzie w Ukrainie.

Pamiętajmy jednak, że ta decyzja ma również swoje ekonomiczne konsekwencje. Ropa sprowadzana statkami jest co do zasady droższa, niż ta sprowadzana rurociągiem. Już teraz widzimy bardzo wysokie ceny paliw, a przecież jesteśmy dopiero na początku tej drogi, ponieważ Polska ok. 64% ropy kupuje z Rosji. Dlatego nie wystarczy zamienić jednego dostawcy na drugiego dostawcę. W dłuższej perspektywie z powodów ekonomicznych rozwiązaniem jest tylko rezygnacja z ropy naftowej w transporcie. Drugi powód, dla którego decyzja Parlamentu Europejskiego jest dobra, to ochrona planety dla naszych dzieci. Uniknięcie katastrofy klimatycznej jest możliwe tylko wtedy, gdy osiągniemy neutralność klimatyczną. W tym wyzwaniu kluczową rolę odgrywa transport, który jest odpowiedzialny za ok. 28% emisji gazów cieplarnianych w UE. Za smog odpowiadają przede wszystkim piece, ale zanieczyszczenia komunikacyjne też są istotne. W skali całego kraju samochody generują ok. 5%, 7% zanieczyszczeń powietrza, ale w dużych miastach to właśnie te toksyczne spaliny mają znaczący wpływ na liczbę przedwczesnych śmierci. Im szybciej zrezygnujemy z samochodów spalinowych w centrach miast, tym będziemy zdrowsi. Zadaniem państwa jest stworzenie takiego prawa i takich mechanizmów finansowych, aby ułatwić obywatelom sprawne odejście od kupowania drogiej ropy i drogiej benzyny. Sprawny, wygodny i tani transport publiczny, autobusy elektryczne lub na wodór, rozwinięta sieć linii kolejowych, ładowarki elektryczne na stacjach benzynowych i na parkingach, dopłaty do samochodów elektrycznych i oczywiście dekarbonizacja całej energetyki - to są działania, które powinniśmy wdrażać już teraz, tak aby osiągnąć zeroemisyjność najpóźniej do 2050 r. lub wcześniej (Dzwonek) i odpowiednio rozplanować ten proces w czasie. Pracy jest dużo, dlatego liczę na to, że polski rząd szybko przyjmie odpowiednie ustawy zaproponowane przez Parlament Europejski. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Górski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie!

Stefana Wyszyńskiego patronem powiatu ostrowskiego. Następnie miała miejsce uroczysta sesja rady powiatu, gdzie zostały odczytane uchwały wspierające wszystkie 11 samorządów gminnych oraz dekret ojca św. zezwalający na podjęcie takiej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie i, co jest warte podkreślenia, również gminy jednogłośnie podjęły tę uchwałę, aby wesprzeć powiat. Jestem zbudowany tą postawą i z tego miejsca pragnę podziękować radnym za podjęcie tej odważnej decyzji, tego zobowiązania, bo w dzisiejszych czasach nie jest łatwo, zwłaszcza w życiu publicznym, opowiadać się po stronie wartości katolickich, a ponieważ jeden przykład znaczy więcej niż tysiąc słów, to z tego miejsca, w którym obok Orła Białego wisi także krzyż, postanowiłem podziękować państwu radnym z powiatu ostrowskiego. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przypominam, że to szczególny dzień, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja. To święto obchodzone jest od 1890 r. dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago, które miały miejsce podczas strajku przeprowadzonego na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. W tym roku Lewica wraz z OPZZ po przerwie spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi zorganizowała pochód pierwszomajowy, który przeszedł ulicami Warszawy. Wiele osób idących bądź stojących obok nas pozytywnie reagowało na zorganizowany przez Lewicę przemarsz, ale niestety stało się coś, co mnie bardzo zasmuciło.

Pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzięki inicjatywie i zabiegom Polskiego Związku Działkowców rodzinne ogrody działkowe mogą otrzymać dotacje nawet do 100 tys. zł na proekologiczne inwestycje realizowane w częściach wspólnych ogrodów działkowych.

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach. Projekty mogą dotyczyć powiększenia powierzchni terenów zielonych, ograniczenia hałasu, zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, a także infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej. Rodzinne ogrody działkowe w miastach oprócz pełnienia tradycyjnej funkcji rekreacyjnej są też cennymi przestrzeniami naturalnej przyrody i stanowią nieodłączną część miejskiej zieleni użytkowej nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach Europy. Dlatego chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie pogratulować i jednocześnie podziękować wszystkim działaczom Polskiego Związku Działkowców, którzy zaangażowali się w pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Kujawsko-pomorscy działkowcy z Bydgoszczy, Inowrocławia i Świecia prosili mnie, żebym z tej trybuny sejmowej, czyli w sposób oficjalny, podziękował Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców za deklarację wsparcia jednostek terenowych w udzielaniu pomocy w wypełnianiu wniosków, bo wiele zarządów ogrodów działkowych będzie po raz pierwszy składało wnioski o środki publiczne. Ze swojej strony też deklaruję pomoc w przypadku wypełniania takich wniosków oraz w przypadku, gdyby konieczne było zwrócenie uwagi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na nieprzewidziane problemy związane z aplikowaniem bądź też z przejrzystością stosowanych procedur. Pani poseł Beata Strzałka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mija kolejny miesiąc od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Przed atakiem Rosji w naszym kraju mieszkało ok. 1 mln Ukraińców. Część z nich to mężczyźni, którzy wrócili do kraju, by go bronić. Część uchodźców wyjeżdża dalej do państw Europy Zachodniej, część zdecydowała się już na powrót do własnego domu, ale większość z nich zostaje w Polsce po to, aby dopiero po zakończeniu wojny wrócić do domu. Na wielki podziw i szacunek zasługuje postawa polskich obywateli, którzy przeorganizowali swoją codzienność, by nieść pomoc potrzebującym. To niezwykle budujące, że tak wielu z nas otworzyło serca i domy dla tych, którzy potrzebowali wsparcia i pomocy, dla tych, którzy w ucieczce przed wojną niejednokrotnie pozostawili dorobek swojego życia i przybyli do Polski jedynie z podstawowymi rzeczami. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim Polakom, którzy odpowiedzieli na potrzeby drugiego człowieka. Dziękuję wolontariuszom, którzy niestrudzenie niosą pomoc na przejściach granicznych, w ośrodkach dla uchodźców i dworcach. Dziękuję tym, którzy przyjęli kobiety i dzieci z Ukrainy pod swój dach, co daje im namiastkę normalnego życia. Wyjątkowa postawa Polaków została dostrzeżona i doceniona również poza zagranicami Polski. Jesteśmy jedynym krajem, który przyjmuje potrzebujących we własnych domach, a nie w obozach dla uchodźców. To pokazuje, jak szlachetne serca mają Polacy. Mając w pamięci bolesne doświadczenia I i II wojny światowej, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na niesprawiedliwość, jaka spotkała Ukrainę. Ta ogromna fala wsparcia jest tego przejawem. W kontekście totalitarnym zapędów Rosji jeszcze bardziej uwydatnia się bezcenna wartość - niepodległość i suwerenność, o które trzeba stale zabiegać. Pamiętajmy o tym szczególnie teraz, by zawsze działać ponad podziałami w interesie naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Głośnym echem odbiły się słowa hiszpańskiego eurodeputowanego Hermanna Tertscha, który stanął w obronie Polski: Ten nieustający szantaż związany z wypłatą pieniędzy dla Polski, gdy ta przyjęła 4 mln uchodźców i w dużej mierze właśnie dlatego musi ponosić te koszty, że Ukraina nie jest broniona. To Niemcy sabotują heroiczny opór Ukraińców. Tak, to Niemcy sabotują systematycznie ich wysiłki, dlatego Polska znalazła się w takiej sytuacji. Teraz jeszcze widzimy, jak Niemcy grożą Polakom, grożą Węgrom, bo ponoć źle się zachowują. A kiedy tu była mowa o łamaniu niezawisłości sądownictwa w Hiszpanii przez socjalistyczno-komunistyczny rząd Hiszpanii? Wypowiedź pana Tertscha, za którą serdecznie mu dziękuję, trwała jeszcze chwilę, po czym wyłączono mu mikrofon. Postawa hiszpańskiego polityka stoi w sprzeczności z zachowaniem polskiej opozycji na forum europejskim, ale przede wszystkim stoi w sprzeczności z postawą wielkich unijnych decydentów. Nikt nie zohydzi Polakom Unii Europejskiej bardziej niż sama Bruksela. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego nałożyliśmy szereg sankcji zarówno na Federację Rosyjską, jak i Białoruś. Celem ustawy była oczywiście solidarność z narodem ukraińskim, ale także uderzenie w gospodarkę rosyjską, z której finansowane są działania zbrojne na terenie Ukrainy. Tak krótki okres wejścia w życie ustawy sprawił, że przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego znalazły się w poważnych tarapatach. Północna część mojego województwa w dużej części czerpała korzyści z wymiany handlowej z obwodem kaliningradzkim. Teraz, w związku z wprowadzeniem rzeczonej ustawy wszelkie transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi a rosyjskimi zostały wstrzymane. Zatrzymanie łańcucha płatności jest niezwykle poważnym problemem dla firm z Warmii i Mazur. To embargo działa w dwie strony. Polskie przedsiębiorstwa nie są w stanie wyegzekwować środków za faktury, które zostały wystawione firmom rosyjskim. Z kolei nasze rodzime firmy nie są w stanie opłacić faktur firmom rosyjskim, które zostały wpisane na listę przedsiębiorstw objętych sankcjami. Należy sobie zadać pytanie, czy Krajowa Administracja Skarbowa czy też inne instytucje nie powinny odblokować rosyjskim spółkom kont, aby te mogły uregulować płatności wobec polskich przedsiębiorstw. Z powodu braku płynności środków dziesiątki firm zawiesiły swoją działalność. Aktualnie ponad 1200 pracowników żyje w strachu o swoje pensje, bo w tak dużą liczbę pracowników zgodnie z wyliczeniami samorządów uderzają sankcje. Firmy z północy Polski, których działalność nastawiona była na wymianę handlową z obwodem kaliningradzkim, nie są w stanie przebranżowić się w tak krótkim czasie. Mowa tu chociażby o terminalach przeładunkowych czy firmach transportowych, które zainwestowały dziesiątki milionów złotych w infrastrukturę. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma dla tych firm, przedsiębiorstw alternatywne rozwiązania? Czy rządzący mają plan na to, aby Braniewo pozostało suchym portem? Czy spółki Skarbu Państwa są w stanie przeprowadzić import towarów z zagranicy przez terminale przeładunkowe w Braniewie? Wysoka Izbo!

Mamy już czerwiec, a rzeczonej odrębnej rekompensaty nie ma. Nie znamy nawet jej treści. Kiedy Rada Ministrów planuje stworzyć specjalne tarcze dla firm pokrzywdzonych przez embargo? Mówimy tutaj o ponad tysiącu ludzi, którzy zostali na bruku bez środków do życia. Wnoszę do przedstawicieli rządu, abyśmy jak najszybciej przegłosowali ustawę, która zrekompensuje firmom Warmii i Mazur straty związane z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską i Białoruską. Pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Dzisiaj głosowaliśmy nad stanowiskiem Senatu odnośnie do Krajowego Planu Odbudowy. Właściwie gdzie jesteśmy, co się wydarzyło?

Niejako zostaliśmy w jakiś sposób odsunięci od możliwości udziału w tworzeniu i dopracowaniu tego planu, co było, uważam, błędem ze strony rządzących. Właściwie nic się nie mówiło przez prawie rok. Minęło lato, jesień, zima.

W pewnym momencie stanowisko Unii jest bardzo wyraźne - mówi o pewnych zobowiązaniach, o pewnych wymogach. Te wymogi są nazwane kamieniami milowymi, czy może kamyczkami, bo są różnej rangi. Są o charakterze zasadniczym, typu problemy z praworządnością, są też mniejszej wagi, aczkolwiek ważne, jeśli chodzi o sprawy związane z energią, z cyfryzacją, ze środowiskiem, a nawet sprawy społeczne, bo Krajowy Plan Odbudowy ma pomóc w naprawie tego, co zostało w jakiś sposób zaniechane, ograniczone przez pandemię, i chodzi o to, żeby nadrobić, przyspieszyć ten rozwój gospodarczy, który został opóźniony. Te negocjacje mają bardzo pogłębiony charakter, bo jest Parlament Europejski, jest Rada Unii Europejskiej, a więc ministrowie 27 krajów w tej sprawie też muszą się wypowiedzieć. Wydaje się, że tracimy dużą okazję skorzystania z możliwości finansowania inwestycji w rozwój gospodarczy.

I jest ogromnym błędem i stratą dla Polski, że nie korzystamy z tych środków, nie korzystamy z zaliczki. Już mogliśmy, tak jak inne kraje, składać kolejne rozliczenia z realizacji różnych projektów, które by mogły.

Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Olszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Punktem kulminacyjnym jubileuszu będzie uroczysta msza święta, która odbędzie się 12 czerwca. Będzie celebrowana przez ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej ks. bp. Romualda Kamińskiego. To ogromna okazja do świętowania nie tylko uroczystości religijnej, ale także historycznej i lokalnej. Region kołbielski położony jest w południowo-wschodniej prawobrzeżnej części Mazowsza, ok. 40 km od Warszawy. Na wschodzie sąsiaduje z Podlasiem, na zachodzie z doliną Wisły, zaś cały region leży w dorzeczu malowniczej rzeki Świder, prawobrzeżnego dopływu królowej polskich rzek Wisły, z ujściem pod Otwockiem. Pierwsza historyczna wzmianka o Kołbieli pochodzi z roku 1407, kiedy na tym terenie powstał kościół zbudowany i założony przez ród Kolibielskich herbu Jasieńczyk, należących do drobnej szlachty ówczesnych właścicieli. Na mocy aktu erekcyjnego z 1422 r. ustanowiona została parafia o rozległym zasięgu. W XVI w. została z niej wydzielona parafia Glinianka, a w okresie międzywojennym - parafia Celestynów. Kołbiel była wtedy wsią szlachecką leżącą w ziemi czerskiej przy historycznym szlaku z Czerska do Liwu. Nazwa miejscowości pochodzi od ludowego określenia grząskiego bagna.

Poważnie ucierpiało w czasie potopu szwedzkiego, powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich, a carski rząd pozbawił je praw miejskich w 1869 r.

Kołbiel jest więc zasadniczą częścią historii Mazowsza. Dlatego chciałbym z tego miejsca podziękować księdzu proboszczowi Krzysztofowi Abramowskiemu za jego (Dzwonek) codzienną pracę nie tylko duszpasterską, ale także poświęconą organizowaniu życia społecznego i kulturalnego w regionie. Wszystkim uczestnikom jubileuszu 600-lecia istnienia parafii w Kołbieli składam życzenia i gratulacje, dziękując państwu za codzienną pracę, jaką wkładacie w kultywowanie tradycji i historii naszych małych ojczyzn. Dziękuję. Pan poseł Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Właśnie dziś, 9 czerwca, odbywają się główne uroczystości związane z obchodami 750-lecia Lublińca. To jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, miasto powiatowe położone na rzekami Lublinicą i Małą Panwią, otoczone lasami, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. To miejsce niezwykłe wytrwale budowane przez kolejne pokolenia, w którym lubi nam się mieszkać, pracować, uczyć się, lubi się nam tu być - jak w 1272 r. powiedział założyciel miasta książę Władysław I Opolski. To przeszłość, czasami burzliwa, momentami dramatyczna, wojenna, powstańcza, ukształtowała nasz dzisiejszy dzień. Czas, który minął, oraz to, w jakim momencie historii się znajdujemy, określa naszą tożsamość. Dzisiaj z pokorą i wdzięcznością spoglądamy na naszych przodków, których wola i determinacja umożliwiły nam świętowanie tego wspaniałego jubileuszu. Przez wieki zmieniały się okoliczności i granice, zmieniały się budynki i mury, pamiętające jeszcze czasy Piastów opolskich, ale zawsze towarzyszyła nam niezwykła, przyjazna atmosfera miasta, która jest jednym z jego największych walorów. To miejsce, do którego chce się zawsze wracać. To miasto jest prawdziwym domem. Okoliczne lasy, liczne trasy rowerowe sprzyjają uprawianiu sportu i wypoczynkowi, a zabytki, bogata oferta kulturalna, muzeum, sanktuarium Edyty Stein i szeroka baza gastronomiczna i noclegowa zachęcają turystów do odwiedzania Lublińca. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w jego rozwój, dziękuję samorządowcom, członkom organizacji stowarzyszeń, ojcom oblatom i naszym parafialnym duszpasterzom, których historia od wieków związana jest z Lublińcem. Dziękuję żołnierzom jednostki wojskowej komandosów, którzy nadają miastu garnizonowego ducha i zawsze służą pomocą. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom. To wasze decyzje, to wasza postawa kształtują Lubliniec jako wspólnotę. Życzę wszystkim lublińczanom kolejnych lat satysfakcji, również z rozwoju miejskiej przestrzeni i infrastruktury. Oby św. Edyta Stein, patronka Europy i Lublińca, otaczała nasze miasto swoim błogosławieństwem, aby ci, którzy przyjdą po nas, mogli w szczęściu i dostatku świętować kolejne wspaniałe jubileusze. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Historia tego wspaniałego festiwalu sięga 1961 r., kiedy to z inicjatywy Janusza Ambrosa, ówczesnego kierownika artystycznego Filharmonii Rzeszowskiej, odbył się pierwszy cykl koncertów pod nazwą Dni Muzyki Kameralnej. Po 20 latach festiwalu nazwa została przekształcona na Festiwal Muzyki Łańcut, który przetrwał pod tą nazwą 10 kolejnych lat. Koncerty w ramach tego festiwalu odbywały się w sali koncertowej Filharmonii Rzeszowskiej oraz w sali lustrzanej zamku w Łańcucie - jednej z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce. W latach 80. dyrektorem majowych koncertów był Bogusław Kaczyński, który dbał o rejestrację telewizyjną koncertów, a przede wszystkim o poziom artystyczny festiwalu, występy znanych gwiazd estradowych, recitale wokalne i pianistyczne.

Ostatnie 2 lata zmieniły formułę festiwalu ze względu na czas pandemii, ale w obecnym roku festiwal powrócił do pełnej, tradycyjnej formy z koncertami w zamku w Łańcucie i w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani dyrektor Filharmonii Podkarpackiej prof. Marty Wierzbieniec odbyło się osiem pięknych koncertów, pełnych najwspanialszej muzyki i kreacji wybitnych muzyków.

Pani prof. Marcie Wierzbieniec gratuluję organizacji tego wspaniałego festiwalu, który jest wielką promocją naszego pięknego Podkarpacia. Bardzo proszę, pani poseł Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziś Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą uporczywego łamania prawa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i obaw co do finansowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Oto ważny fragment tej rezolucji, cytuję: Parlament Europejski wyraża poważne zaniepokojenie pozytywną oceną przez Komisję Europejską przedłożonego przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy, biorąc pod uwagę istniejące i wciąż trwające naruszenia przez Polskę wartości zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej, w tym praworządności i niezależności sądownictwa. Od wybuchu wojny w Ukrainie polskie władze podjęły szereg działań wprost sprzecznych z trzema warunkami postawionymi przez Komisję Europejską. Po pierwsze, 25 lutego zawieszono polską sędzię Annę Głowacką za stosowanie prawa europejskiego i wyroków sądów europejskich. Po drugie, polski prezydent wręczył nominacje ponad 200 nowym, nieprawidłowo powołanym na wiosek neo-KRS tzw. neosędziom, w tym cztery nominacje do Sądu Najwyższego. Po trzecie, upolityczniony i w pełni podporządkowany Trybunał Konstytucyjny podważył ważność art. 6 Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poprzez kwestionowanie jego kompetencji do badania prawidłowości powoływania sędziów i niezawisłości neo-KRS. Koniec cytatu. Dzisiejsze odrzucenie przez Prawo i Sprawiedliwość większości poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym najlepiej pokazuje prawdziwe intencje polskiego rządu. Polskie prawo wciąż będzie przez ten rząd łamane, a sędziowie - szykanowani. Premier Morawiecki wciąż będzie sojusznikiem Viktora Orbána, sojusznika Władimira Putina. Dzisiejsze głosowanie w polskim parlamencie to ważny sygnał dla pani i całej Komisji. Fundusz Odbudowy jest potrzebny Polkom i Polakom, ale nie za cenę bezprawia i niesprawiedliwości, które od 7 lat rujnują nasz kraj. Niepowstrzymane, teraz rozleją się na całą Europę.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Bąk, Prawo i Sprawiedliwość.

18 maja 1944 r. Polacy odnieśli tam zwycięstwo nad Niemcami, którzy mieli wyjątkowe umocnienia, byli pewni swego i próbowali lekceważyć nasze możliwości. Już po zwycięskiej bitwie dowódca korpusu polskiego otrzymał od dowódcy 8. armii list. Cytuję: Dzielność polskich oddziałów w tych zaciętych walkach oraz sposób, w jaki utrzymały one ciężki ogień moździerzowy i artylerii oraz uporczywe natarcia, były dla mnie rewelacją. Pewny jestem, że ten pamiętny czyn przejdzie do historii jako wspaniałe osiągnięcie oręża polskiego, a w naszej historii wojskowej na pewno zaliczony będzie do wybitnych sukcesów 8. armii. Wysoki Sejmie!

Chciałbym w tym miejscu wyrazić szacunek dla wójta Starej Błotnicy Marcina Kozdracha i dla księdza proboszcza parafii Kaszów Ireneusza Chmury, głównych inicjatorów tego przedsięwzięcia. W uroczystości wzięli udział znamienici goście. Przyjechał ambasador Polski we Włoszech, pani Anna Maria Anders, była senator RP, pan marszałek Stanisław Karczewski, oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego. Były sztandary ochotniczych straży pożarnych, sztandary szkół z terenu gminy Stara Błotnica, okoliczna ludność.

Tak dalej być nie może. Trzeba brać przykład z bohaterów Polski, a nie zapatrywać się na szkodzące Polsce postawy. Zapraszam, pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Regularnie spotykam się z samorządowcami z mojego okręgu wyborczego. Poruszamy różne tematy, omawiamy wspólne działania, ale zawsze wiem, że prędzej czy później padnie pytanie: Panie pośle Arturze, kiedy wreszcie Sejm zajmie się podatkami od tzw. apartamentowców? Jak długo mamy być robieni w konia? Otóż gminy i miasta żyjące z turystyki od kilkunastu lat przeżywają niebywały boom w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Niestety nie ma to nic wspólnego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców tych gmin i miast. Statystyki nabijają apartamentowce. Deweloperzy je budują. Nie ma w tym nic złego. Ludzie kupują w nich mieszkania, lokale czy - jak kto woli - apartamenty. W tym także nie ma nic złego.

Oczywiście w chęci osiągnięcia zysku również nic nie ma nagannego, natomiast naganne jest osiąganie tych zysków przy użyciu metod niemających nic wspólnego z uczciwą konkurencją.

Czy w takich warunkach można normalnie konkurować?

Dlatego nie można się dziwić samorządowcom, że próbują walczyć o należne lokalnym społecznościom podatki. W odpowiedzi otrzymałem dość obszerne wyjaśnienie co do zasad ustalania stawki podatku od nieruchomości, wskazano również orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących sporów między samorządem a płatnikami podatku od nieruchomości. Ponadto zawarta była też informacja, że od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie dyrektywa Rady Unii Europejskiej nakładająca nowe obowiązki na operatorów platform cyfrowych, które przyczynią się do uszczelniania systemu podatkowego, także w kontekście podatku od nieruchomości. Wszystko to wygląda obiecująco, ale tylko z pozoru. Bez zmiany ustawy o podatku i opłatach lokalnych samorządy będą skazane na przysłowiowe ciąganie się po sądach (Dzwonek) z próbującymi obchodzić przepisy podatnikami, a przecież nie o to chodzi. Dlaczego, żeby wyegzekwować należny podatek, samorząd ma iść do sądu, po co tracić czas i pieniądze? Według wielu samorządowców wystarczy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w art. 2a ust. 1 dodać warunek zameldowania się właściciela nieruchomości. Tylko tyle i aż tyle. To precyzyjnie zdefiniuje nieruchomość zaspokajającą potrzeby mieszkaniowe obywatela i pozwoli uniknąć sądowych utarczek. Od pewnego czasu Ministerstwem Finansów kieruje nowa pani minister, co daje nadzieję na nową jakość w tym resorcie. Dlatego zwrócę się do pani minister z interpelacją i zapytam, czy nie zechciałaby zlecić odpowiedniemu departamentowi podjęcia działań w tym ważnym zakresie. Pan poseł Krzysztof Śmiszek, Lewica. Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.